tego meteorytu, któryście sami ściągnęli na polską ziemię. Wywołaliście katastrofę gospodarczą, społeczną, kulturalną, polityczną pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Informuję pana, że oczywiście działamy na podstawie prawa, ale i odpowiedzialności za zdrowie i życie innych. Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do pytań. Konsekwencje pan zna. Zamykam listę osób chcących zadać pytanie. Jako pierwszy pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska.

Panie Ministrze! W budżecie, o którym dzisiaj mówimy, w jego nowelizacji, państwo zakładacie prawie 1300 mln zł w części 48 dotyczącej górnictwa. Chciałem się zapytać, czy te środki są już przeznaczone na realizację porozumienia, które rząd podpisał.

Kiedy nastąpi przekazanie zadań Centralnej Pompowni Bolko Spółce Restrukturyzacji Kopalń? Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Od lat narasta dziura finansowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a ściśle mówiąc, w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W pierwotnej wersji budżetu na ten rok przewidziano dopłatę z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 45 mld zł. Zgodnie z nowelą przedstawioną Wysokiej Izbie ta dopłata z budżetu - środków budżetowych - wyniesie 57 mld zł, ale to nie wszystko, ponieważ oprócz tego ZUS zostanie zasilony kwotą 38 mld zł z funduszu COVID-owskiego.

Chciałbym zapytać przedstawicieli rządu, jeżeli są tacy na sali.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na Śląsku sytuacja w służbie zdrowia jest taka, że już brakuje miejsc w szpitalach zakaźnych dla chorych na koronawirusa, więc umieszcza się ich w zwykłych szpitalach, w wyniku czego inni potrzebujący leczenia nie mogą na nie liczyć. Tak dramatyczna sytuacja jest w służbie zdrowia. To są oczywiste powody tego, że budżet wymaga nowelizacji i zwiększenia wydatków. Na wojsko. Nie na służbę zdrowia, nie na edukację, nie na wsparcie gospodarki, ale na wojsko. Naprawdę, co trzeba mieć w głowie? Dlaczego ten rząd postępuje wbrew żywotnym interesom społeczeństwa polskiego?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Nie wiem, kto będzie odpowiadał, ale chciałbym zapytać, czy państwo analizując i przygotowując tę nowelizację budżetu, zdiagnozowali potrzeby dwóch bardzo poważnych obszarów funkcjonowania naszego kraju w dobie epidemii. Bo ta mała kropla w morzu potrzeb jest zapewne niewystarczająca. Drugim obszarem, o który chcę zapytać, jest obszar edukacji. Czy państwo wiecie i możecie nas poinformować, ile pieniędzy muszą dołożyć samorządy do zapowiedzianych, zrealizowanych podwyżek dla nauczycieli przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, który obiecuje, realizuje, a nie daje na to pieniędzy samorządom? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Każdy dzień października przynosi nam nowe, zatrważające informacje o nowych zakażonych czy zmarłych z powodu koronawirusa.

Czy nowelizacja tego budżetu w jakikolwiek sposób odpowiada na wyzwania chwili? Pytam, ile środków przeznaczyliście państwo dla pracowników sanepidu, na wzmocnienie wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych? Ile środków przeznaczyliście na wsparcie ochrony zdrowia, szczególnie na uruchomienie nowych COVID-owych łóżek? Wreszcie ile środków zapewniliście na walkę z pandemią? W Małopolsce od marca przeznaczyliście na walkę z epidemią koronawirusa 6 mln zł. To jest po prostu wstyd. W tym budżecie nie ma na to ani grosza, za to robicie sobie poduszki po to, aby dalej robić sobie geszefty.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Miało wystarczyć pieniędzy na wszystko, mieliście nas więcej nie zadłużać. Okazuje się, że potrzebujecie pożyczyć 110 mld zł, aby wystarczyło na wszystkie wydatki w tym roku. Czy te pieniądze pójdą na walkę z epidemią, na wsparcie służby zdrowia, na wsparcie lekarzy sanepidu? Nie, te pieniądze pójdą na wypłatę trzynastych emerytur, na górnictwo węglowe, na policję i na armię, na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Skoro wydajecie pieniądze, których nie macie, to znaczy, że zwiększacie zadłużenie. Oznacza to, że każdy Polak będzie miał kredyt na 36 421 zł. Zadłużacie nasz kraj najszybciej w Europie. Czy to waszym zdaniem jest odpowiedzialne [[Dzwonek]] i czy zdajecie sobie sprawę z tego, że podążanie tą drogą prowadzi do scenariusza greckiego?

Pan Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska.

Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Jeżeli w kraju szaleje koronawirus, jeżeli mamy 3003 przypadki jednego dnia i 78 ofiar śmiertelnych, to co powinno być priorytetem w przypadku nowelizacji budżetu państwa? Oczywiście przeciwdziałanie koronawirusowi. Oczywiście walka z epidemią. Oczywiście zabezpieczenie tych najsłabszych, najbardziej narażonych. Szanowni Państwo! W tym budżecie pojawia się deficyt. Miał być rok bez deficytu, budżet bez deficytu. Problemem jest nieprzygotowanie społeczeństwa i państwa na jesienną pandemię. W Polsce jest 1 mln chorych na choroby onkologiczne. W Polsce jest kilka milionów osób starszych z wielochorobowością. Ile jest szczepionek na grypę? Szczepionki na grypę miały być priorytetem, elementem strategii państwa. Ich po prostu nie ma.

Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dyskusja o budżecie często biegnie obok tego, co to oznacza dla zwykłych ludzi, aktywnych, przedsiębiorczych, codziennie ciężko pracujących, czy dla seniorów. Czasem warto zadać sobie pytanie, co ta dzisiejsza nowelizacja oznacza dla takich ludzi. Bo ten wielki dług, który generuje dziś PiS, uderzy właśnie w tych, którzy codziennie ciężko pracują, a nie w leni i nierobów, bo oni oczywiście mają swoje zaszczytne miejsce w polityce PiS i im się nic nie stanie.

Każdy Polak, każda Polka, każdy senior, którzy mają dziś oszczędności, systematycznie je tracą z powodu polityki Prawa i Sprawiedliwości.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Natomiast w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej w związku ze skutkami pandemii COVID-19 przewidziano zwiększenie wydatków w tej części o kwotę prawie 2 mld. Tak to się ma globalnie. Gdy przegląda się zwiększeniu kwot na wydatki zaproponowane dla konkretnych województw, to okazuje się, że w 11 województwach faktycznie będą dodatkowe środki, natomiast w pozostałych pięciu, tj. dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i zachodniopomorskim, planuje się zmniejszenie wydatków. W związku z powyższym proszę o odpowiedź, najlepiej na piśmie, na pytanie: Jaka jest przyczyna, że jednym województwom zwiększa się budżety, a innym obniża? Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.

I proszę nie przekonywać nas, proszę nie przekonywać Polaków, że jedynym powodem tego ogromnego deficytu, którego nie mieliśmy w tej wysokości od 30 lat, jest wyłącznie epidemia. Chcę wiedzieć, jaki jest całkowity deficyt sektora finansów publicznych w Polsce, ponieważ ekonomiści mówią, że może on wynosić nawet 300 mld zł.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Jeżeli naprawdę zależy wam na nowelizacji budżetu, dobrej nowelizacji budżetu, to może najwyższa pora zostawić w spokoju spółki Skarbu Państwa. Kiedy zamierzacie skończyć z programem: rodzina PiS-u na swoim i nieudolnym zarządzaniem przedsiębiorstwami? Przypomnę, że od kiedy działa Ministerstwo Aktywów Państwowych, wartość największych państwowych spółek spadła o 22%, czyli o 57 mld zł. 57 mld zł to jest połowa tego, co w tym roku wydamy na służbę zdrowia, a to tylko straty do czasów pandemii, bo to kolejne 5 mld zł w dół. Mówię tylko o spółkach notowanych na giełdzie, a przecież w całym kraju są jeszcze tysiące państwowych instytucji tak samo nieudolnie zarządzanych i przynoszących straty tylko dlatego, że ktoś należy do jedynie słusznej partii. 62 mld zł strat - po to, żebyście mogli wypłacać sobie menedżerskie pensje. Odpuśćcie sobie. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Rozmawiamy dzisiaj o lawinowo rosnącym deficycie i zrujnowanych finansach publicznych, a na sali nie ma nawet ministra finansów. To, co dzisiaj trzeba zrobić, to ogłosić zero tolerancji, ale dla marnowania pieniędzy publicznych. Cały czas słyszeliśmy, przez 5 lat, propagandę sukcesu, o tym, jakie mamy zdrowe finanse publiczne, a tymczasem kryzys kompletnie to obnażył.

To jest rachunek po 5 latach waszych rządów i krótkim kryzysie. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Faktycznie, gdzie jest minister finansów? Tak ważna debata, niestety, nie ma ministerstwa w ogóle. W nowelizacji budżetu wprowadza się wiele zmian polegających na zwiększeniu środków na wydatki, które poniesione będą w roku 2021 - transfery socjalne, pieniądze na inwestycje - a tymczasem rząd nie zabezpiecza środków na wydatki, które są niezbędne w tym roku. Wysoki Sejmie! Dlaczego rząd nie zabezpiecza środków na edukację, na oświatę? Czy rządowi nie zależy na polskiej oświacie? Przecież samorządy nie pokryją tej ogromnej dziury budżetowej, która dotyczy polskiej oświaty. Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Premier Morawiecki mówił, że to będzie historyczny budżet z zerowym deficytem. Jest historyczny, ale z największym deficytem, ponad 100 mld zł. Państwo twierdzicie, że ten deficyt jest spowodowany pandemią. Państwo wydawaliście, jak chcieliście, komu chcieliście, bez przetargu. Pan minister zdrowia w piątek nam powiedział, że w październiku wrócą pieniądze za respiratory - przypomnę, chodzi o 70 mln zł. No i mamy projekt zmiany ustawy budżetowej na rok 2020, i szukam.

I mam pytanie do pana ministra: Dlaczego państwo tego nie wpisaliście, skoro jesteście pewni, że on te pieniądze odda? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Realny deficyt sięga dziś nie 110 mld zł, a 300 mld, bo należy dodać do tego zobowiązania zaciągnięte przez Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju. Na dodatek w tegorocznym budżecie zapisano również przyszłoroczne wydatki na 13. i 14. emeryturę oraz inne świadczenia. To po prostu kreatywna księgowość. Moje pytanie dotyczy konkretnie tego, na co przewidziane są środki, które są ujęte w tej nowelizacji. Mam również pytanie, jak się zdaje, retoryczne: Gdzie jest minister finansów? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Powtórzmy to jeszcze raz. Deficyt budżetu ma wynieść ponad 109 mld zł wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu, ale realnie ten deficyt wyniesie 300 mld zł. Należy do niego dodać zobowiązania zaciągnięte przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju. Dodatkowo zobowiązania przyszłoroczne - 13. i 14. emerytura - przenosicie na ten rok. Zamiast znacznie zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia i edukację, 3 mld zł dodatkowo trafią na armię. Te kwoty na armię wydane w roku 2020 to w sumie 52 mld zł.

Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. W takim razie pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! W poniedziałek w wielu miejscach w Polsce rolnicy odwiedzili biura poselskie i parlamentarzystów.

Przypomnę, że te dopłaty wynoszą 65% do 1 ha i jednego zwierzęcia gospodarskiego.

Dlatego też klub parlamentarny Lewicy wniósł poprawkę zwiększającą wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników o kwotę 250 mln zł. O tym mówili rolnicy na spotkaniu izby rolniczej w Słupcy, na spotkaniu w Gnieźnie i w innych miejscowościach wielkopolskich. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niedawno „Solidarność” przemysłu zbrojeniowego ogłosiła pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach zbrojeniowych w Polsce w związku ze złą sytuacją tej branży i śladowym udziałem krajowych zakładów w procesie modernizacji polskiej armii. Polski przemysł zbrojeniowy jest pomijany w wielu kluczowych programach modernizacji armii, a zakupy uzbrojenia dla polskiej armii w Polsce są wyłącznie na papierze i w propagandzie sukcesu uprawianej przez ministra obrony narodowej. Związkowcy z zakładów elektromechanicznych Belma i Nitro-Chemu z Bydgoszczy, z mojego okręgu wyborczego, publicznie twierdzą, że pieniądze na zakupy uzbrojenia wydawane w tej chwili wcale nie trafiają do polskiej armii. Mam w związku z tym pytanie: Kiedy minister obrony narodowej i minister aktywów państwowych spotkają się z przedstawicielami branży?

Nie wiem, jakie alibi ma minister finansów, że nie przychodzi na posiedzenie Sejmu, bo nie widzę żadnego uzasadnienia, żeby przysyłał wiceministra. A przecież rozmawiamy o zabezpieczeniu Polaków. Ten budżet to budżet skandaliczny, 300 mld zł długu, i państwo szukacie alibi. My zaproponowaliśmy 3 mld zł na zdrowie, bo nie ma ważniejszej rzeczy dla Polaków niż zdrowie i zabezpieczenie w okresie pandemii, i 2 mld zł dla samorządów.

Państwo nie potraficie przeprowadzić najprostszej rzeczy: koordynacji miejsc w szpitalach, a co dopiero zarządzania (Dzwonek) finansami. Pan poseł Wojciech Saługa. Wysoki Sejmie! Jaki jest stan finansów państwa, najlepiej widzi to każdy Polak, jak wyciąga pieniądze z bankomatu - najczęściej nowe dwusetki, czasami już pięćsetki. Drukujecie pieniądze na potęgę, psując tym finanse państwa, i wywołujecie gigantyczną inflację, inflację, która jest ukrytym podatkiem, który zapłacą najbiedniejsi, kupując towary w sklepach. Chciałbym zapytać: Jaki jest stan, wielkość tych skupionych obligacji w stosunku do tego, co było robione rok wcześniej i rok wcześniej?

Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kilka miesięcy temu premier Morawiecki mówił o zrównoważonym budżecie, pierwszym w historii. I dzisiaj nie mam żadnej satysfakcji z tego powodu, bowiem to, że państwo dzisiaj przyznajecie się, że brakuje ponad 109 mld zł, pokazuje jeszcze coś innego - że prawda jest dużo gorsza, że w tym budżecie brakuje dwa albo i trzy razy więcej środków finansowych. Drugi. Jeśli państwo chcecie teraz ten budżet w pewnym sensie modernizować, to popatrzmy, gdzie są dzisiaj wyzwania. Drugi element to przedsiębiorcy - tracimy miejsca pracy. Trzeci - gdzie [[Dzwonek]] jest wsparcie dla samorządów?

Wysoka Izbo! Podczas debaty na poziomie Komisji Finansów Publicznych i podczas tej debaty padło wielokrotnie stwierdzenie dotyczące zadłużenia państwa. Aby zrozumieć tę sytuację, trzeba przypomnieć historię długu publicznego PDP na przestrzeni ostatnich lat. W 2007 r., gdy Prawo i Sprawiedliwość kończyło rządy, dług publiczny wynosił 527 mld zł, czyli przez 2 lata rządów dług publiczny wzrósł o 60 mld zł, co daje wzrost roczny o 30 mld zł.

W takim razie lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania, które dotyczą bezpośrednio zagadnień związanych z zakresem kompetencji ministra finansów. Pierwsze pytanie dotyczyło dokapitalizowania i przeznaczenia dodatkowych środków na górnictwo. Z tego... miliarda 300... 879 mln to są środki na dokapitalizowanie spółki SRK. Według mojej najlepszej wiedzy te środki są również zabezpieczone na przejęcie tej przepompowni, o którą pytał pan poseł. Druga rzecz to kwestia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zwracam uwagę, że 38 mld to środki związane ze spadkiem makro oraz tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców. Ponadto zwracam uwagę, że w 2020 r. nie było reformy OFE i tych środków również nie uwzględniono w budżecie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w 2021 r. proponowana jest waloryzacja rent i emerytur. Dużo pytań dotyczyło wzmocnienia służby zdrowia.

Jeżeli chodzi o kwestie wydatków samorządowych, to zwracam uwagę, że w przyszłym roku subwencja rośnie o 3,4 mld zł, a w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego trafi dodatkowo 12 mld zł z funduszu COVID, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Padały także pytania o kwestie związane ze wzmocnieniem sanepidów. To wzmocnienie będzie miało swój dalszy ciąg w części ministra zdrowia w roku 2021. Dodatkowo kwestia dotycząca banku centralnego: zwracam uwagę na problematykę niezależności banku centralnego i jego polityki, ale narzędzie tzw. quantitative easing jest często wykorzystywane nie tylko przez Narodowy Bank Polski, ale również przez Europejski Bank Centralny czy przez rezerwę federalną Stanów Zjednoczonych. Jaki jest deficyt sektora finansów publicznych? Obecnie szacujemy to, łącznie z funduszami PFR-u i Banku Gospodarstwa Krajowego, na około 11% produktu krajowego brutto za ten rok.

Tak jak powiedziałem, środki w tym roku i w przyszłym roku na 6-procentowe podwyżki dla nauczycieli zostały zapewnione. Padło też pytanie o zwrot środków z tytułu zakupu respiratorów. Tutaj nie chciałbym wyręczać ministra zdrowia. Niemniej jednak zwracam uwagę, że dochody są tylko prognozą, więc gdy te środki się pojawią, to po prostu wpłyną na budżet państwa i przez to zmniejszy się deficyt. Padło też pytanie o zwiększenie środków dla rolnictwa.

Ze środków związanych z finansowaniem obronności mamy zapewnienia ministra obrony narodowej, że zdecydowana większość tych środków, bo ok. 2/3, trafi do firm krajowych. Padło też pytanie o niewielkie kwoty związane z przesunięciem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wysoki Sejmie!

Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 239 i 598) Proszę pana posła Dariusza Stefaniuka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych z druku nr 239 wpłynął do Sejmu 6 lutego 2020 r., na 10. posiedzeniu Izby 15 kwietnia br. odbyło się jego pierwsze czytanie. Następnie dokument skierowano do dalszych prac w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 4 maja br. komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do jego rozpatrzenia, której miałem zaszczyt przewodniczyć. Podkomisja pracowała nad projektem w trakcie dziewięciu posiedzeń. Projekt ustawy wprowadza nowe zasady doręczania korespondencji przez podmioty publiczne do podmiotów publicznych, jak również do podmiotów niepublicznych, w tym osób fizycznych. Celem projektu jest skrócenie czasu doręczania korespondencji, a także umożliwienie załatwiania spraw urzędowych na odległość, bez konieczności udawania się do placówki operatora pocztowego. Szczególnie w dobie pandemii widzimy, jak Polacy zmienili swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. W czasach, gdy za pomocą telefonu kupujemy bilety lotnicze, płacimy w sklepie, uczniowie i studenci mają zajęcia przez Internet, kontakt obywatela z urzędnikiem pozostaje taki sam jak niemalże 100 lat temu. Proponowane w projekcie rozwiązania zakładają, że e-doręczenie będzie pod względem prawnym równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego, m.in. za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja elektroniczna, czyli e-maile, zastąpią dotychczasową korespondencję listowną pomiędzy wszystkimi instytucjami państwa, urzędami i sądami, pomiędzy władzą a obywatelami i firmami, oczywiście za pomocą specjalnie stworzonego rejestru. Wynika to z kwestii bezpieczeństwa, rzetelności czy zachowania tajemnicy korespondencji. Na potrzeby wprowadzenia tych nowatorskich rozwiązań zostanie utworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Początkowo za organizację całego procesu korespondencji odpowiadałby narodowy operator, czyli Poczta Polska. Wynika to również z faktu, że w projekcie wprowadza się tzw. usługę hybrydową. Osoby wysyłające tradycyjny list do instytucji mają gwarancję, że zostanie on zeskanowany do systemu i przesłany instytucji. Podobnie jest w odwrotnej sytuacji. Jeśli obywatel życzy sobie, aby otrzymywać korespondencję tylko elektronicznie, to gdy jest ona wysłana w formie papierowej, operator, jakim jest Poczta Polska, odpowiada za zeskanowanie i przesłanie tej korespondencji elektronicznie. Oczywiście wejście projektu w życie wymaga dostosowania kilkudziesięciu innych ustaw. Stąd też długie vacatio legis, jakie wynika ze specyfiki kolejnych instytucji.

Zgłoszono również 24 wnioski mniejszości. Komisja przyjęła projekt ustawy z poprawkami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Witold Czarnecki. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu parlamentarnego mam zaszczyt przedstawić paniom i panom posłom stanowisko mojego klubu odnośnie do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 239 i 598) Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych to trudna i skomplikowana ustawa, nie tylko wprowadzająca nowe rozwiązania techniczne, ale także zmieniająca kilkadziesiąt ustaw w zakresie sposobu doręczania dokumentów. Zaproponowane w tej ustawie rozwiązania to milowy krok w cyfryzacji Polski. Dzięki tej ustawie cyfryzacja wchodzi w nowe, wcześniej nieregulowane lub słabo scyfryzowane dotychczas obszary. Wprowadzone rozwiązania będą miały zastosowania do najważniejszych procedur: administracyjnej, cywilnej i karnej. Jakie korzyści płyną z proponowanych w tym projekcie zmian? Po pierwsze, przyjęte rozwiązania zapewnią wszystkim, zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym - w szczególności osobom fizycznym - możliwość korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie można wykorzystać do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z doręczeń elektronicznych.

Po trzecie, skróci się czas potrzebny na doręczenie pism, podań, wniosków oraz odpowiedzi na nie. Zapewnią również pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo lub też tym, które nie są jeszcze gotowe na komunikację elektroniczną, możliwości korzystania z aktualnie dostępnej przesyłki listowej.

Dlatego na szczególną uwagę zasługuje przewidziana w projekcie ustawy zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego, która zapoczątkuje kierunek kolejnych zmian legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia tzw. domyślności cyfrowej w kontaktach z administracją. W zmianie dotyczącej Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono równoważność pism służących załatwianiu spraw bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej, czy na papierze. Ponadto stworzono podstawy do automatycznego załatwiania spraw dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi tj. środki identyfikacji elektronicznej i kwalifikowane pieczęcie elektroniczne organów. Zmierzając do podsumowania mojej wypowiedzi, chcę podkreślić, że brak uchwalenia tej ustawy spowodowałby pozostawienie dotychczasowego sposobu doręczania opartego na doręczaniu tradycyjnym, listowym oraz przy użyciu różnych systemów i adresów elektronicznych. W dalszym ciągu obywatel czy przedsiębiorca będzie zmuszony pamiętać o wysłaniu pisma do konkretnego urzędu, o informowaniu o każdej zmianie adresu, o wielu loginach, hasłach do różnych systemów teleinformatycznych i różnych adresów elektronicznych. Na koniec, co równie ważne, nie nastąpi tak wyczekiwane przyspieszenie wymiany korespondencji z administracją publiczną czy sądami.

To konieczność, a jednocześnie szansa na realizowanie zadań publicznych na rzecz obywateli w sposób ciągły i niezakłócony. Temu wyzwaniu czasów, jakim jest zapewnienie sprawnego działania państwa teraz i w przyszłości, odpowiada projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Mając na uwadze przedstawione argumenty, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za uchwaleniem ustawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Michał Gramatyka. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ta ustawa naprawdę tworzy nową jakość.

Przeniesienie urzędowych doręczeń do świata cyfrowego jest gigantyczną korzyścią dla środowiska. To jest korzyść mierzona w milionach zaoszczędzonych wozokilometrów, w dziesiątkach tysięcy zaoszczędzonych ryz papieru. Prawem opozycji jednak jest krytykować, warto więc wspomnieć, że ustawa w dalszym ciągu nie jest wolna od wad i elementów wątpliwych. Spore kontrowersje budzi np. wymóg odpłatności za usługę elektronicznego doręczenia. Nie przekonuje nas argumentacja ministerstwa wskazująca na konieczność zabezpieczenia przychodów Poczty Polskiej.

W dalszym ciągu ustawa ma wejść w życie - nazwałbym to - na raty, stopniowo obejmując kolejne obszary, kolejne ministerstwa i kolejne instytucje państwa.

Prowadziłem w tym zakresie kontrolę poselską, usiłując ustalić, jaki los spotkał dane osobowe setek tysięcy Polek i Polaków przekazane Poczcie Polskiej po słynnym mailu do samorządów z 23 kwietnia br. Poczta twierdzi, że zrobiła to na polecenie pana premiera, a w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie szef polskiego rządu nie miał prawa do wydania takiego polecenia. Winnych dzisiaj oczywiście brak. Trudno też dociec, co stało się z rekordami przekazanymi poczcie przez 532 polskie gminy. Wiadomo, że dane były przetwarzane, nie do końca wiadomo, przez kogo i w jaki sposób. I m.in. dlatego koncepcja wskazania tej państwowej firmy jako operatora wyznaczonego na kolejne 5 lat budzi tak głębokie wątpliwości. Oczywiście nie mniej ważne jest zachowanie pewnych nadrzędnych europejskich wartości: zasady uczciwej konkurencji, zasady równego dostępu do rynku, przejrzystości czy niedyskryminacji. Przy okazji rozważań na temat roli operatora wyznaczonego warto jeszcze raz podkreślić konieczność zabezpieczenia usługi tzw. doręczenia hybrydowego. To nic innego jak wydrukowanie elektronicznie nadanej przesyłki. To chyba najsłabszy punkt w całym systemie, który opisuje ustawa. Wymaga to fizycznego zaangażowania pracownika poczty. Czy i jak zostanie zagwarantowane nasze prawo do prywatności? Liczymy, że ta kwestia doczeka się precyzyjnego uregulowania w aktach niższego rzędu. W ramach wniosków mniejszości klub Koalicji Obywatelskiej zaproponuje państwu modyfikacje ograniczające monopol Poczty Polskiej. Jednakowoż klub ma świadomość wagi tej ustawy w budowaniu fundamentów cyfrowego państwa, dlatego nie będziemy się sprzeciwiać przyjęciu tych przepisów.

To jest poprawka o charakterze ściśle legislacyjnym, usuwa powielanie się zmian w tych samych przepisach. Gdybyśmy jej nie przedłożyli i nie przyjęli, ustawa pewnie wróciłaby z Senatu z jedną więcej zmianą do rozpatrzenia. W imieniu klubu Lewica głos zabierze pan poseł Robert Kwiatkowski. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! O ustawie o doręczeniach elektronicznych można mówić, cytując poszczególne zapisy tej rzeczywiście skomplikowanej ustawy, posługując się techniczną i legislacyjną nowomową. Można też próbować opowiedzieć o niej i ustosunkować się do jej zapisów, do tego, przypomnijmy, rządowego przedłożenia, językiem prostszym. Pozwólcie państwo, że spróbuję tej drugiej metody. Ustawa o doręczeniach elektronicznych to, szanowni państwo, nic więcej jak instrukcja obsługi korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną.

To jednocześnie, Wysoka Izbo, fundament e-państwa, państwa, które jest znacznie sprawniejsze, które działa w oparciu o elektroniczny obieg dokumentów nie tylko pomiędzy poszczególnymi organami, ale przede wszystkim na styku między państwem a obywatelem. Jeśli tak dobrze to wygląda, to chciałoby się zapytać, jak przebiegały prace nad tą ustawą, a przede wszystkim chciałoby się, Wysoka Izbo, zapytać, co na to organa administracji rządowej. Gdzie jest rząd, który powinien reprezentować to przedłożenie? Miałem okazję pracować w podkomisji powołanej w celu opracowania tej ustawy. To była trudna praca, bo ona przede wszystkim polegała na uzgodnieniu stanowisk legislatorów sejmowych ze zmieniającymi się kolejno wysokimi urzędnikami administracji rządowej. Chciałbym wyrazić ubolewanie, że na tej sali w trakcie dyskusji nad fundamentalną - i wszyscy, niezależnie od barw partyjnych, to podkreślają - ustawą, która ma na nowo regulować relacje między obywatelem a państwem, brakuje przedstawiciela administracji rządowej odpowiedzialnego za sprawy informatyzacji, czyli ministra odpowiedzialnego za te sprawy, tj. Mateusza Morawieckiego.

Szczęśliwie jest z nami pan minister Andruszkiewicz. Witamy.

Nie ma z nami także pani minister Wandy Buk, która zrezygnowała w odpowiednim czasie ze stanowiska w Ministerstwie Cyfryzacji. Ona pilotowała ten jakże trudny i wymagający projekt. Jednym słowem, nie dość, że doszło do rotacji na tych kluczowych stanowiskach, które z ramienia administracji rządowej mają zajmować się tym trudnym projektem, to jeszcze doszło do likwidacji samego Ministerstwa Cyfryzacji. Źle to, drodzy państwo, rokuje. Obiecuję w imieniu klubu Lewicy, że będziemy monitorować ten projekt, bo jego, że tak powiem, droga legislacyjna zapewne niedługo się skończy. Klub Lewicy, pani marszałek, będzie głosował za przyjęciem tego projektu, ale kluczowe nie jest uchwalenie choćby najlepszego prawa. Kluczowa jest realizacja tego prawa. Tu nasuwa się, pozwolę sobie jeszcze zaznaczyć ten wątek, sprawa vacatio legis. O tym mówił jeden z moich poprzedników, słusznie wskazując, że ono jest podzielone na kilka niezrozumiałych dla opinii publicznej etapów. Koniec końców ustawa ma wejść w życie dopiero po 9 latach.

Mam na myśli stronę administracji rządowej. Kończę swoje wystąpienie apelem do przedstawiciela rządu (Dzwonek), żeby zmobilizować te siły i środki, jakie są do państwa dyspozycji, i przypilnować, by po zakończeniu procesu legislacyjnego ten projekt był wdrażany z należytą starannością.

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych. Procedowany projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gospodarki i społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, iż należy zmienić sposób nadawania i odbierania przesyłek urzędowych i skończyć ze znienawidzonym przez wszystkich awizo i staniem w urzędach, jak również na poczcie. Chcę zwrócić uwagę Wysokiej Izby, iż jest to znacznie spóźniony krok w przyszłość. Rozwiązanie to od lat funkcjonuje w Estonii, Danii, Francji, Niemczech czy Czechach. Pani Marszałek! Moi poprzednicy zwrócili uwagę na zalety oraz wady tej ustawy. Ja chciałbym się skoncentrować na rzeczy najważniejszej dla Polaków, czyli na zaufaniu, któremu chciałbym poświęcić resztę mojego wystąpienia. Wysoka Izbo! Mija 5 lat, od kiedy Zjednoczona Prawica objęła stery Polski. Nie mogę pominąć pytania, dlaczego kolejny raz okazało się, że rząd nie dotrzymuje własnych obietnic. Procedowana ustawa miała być wdrożona już w roku 2019. Jest to ostatni z licznych przykładów zaniechań rządzących. Tu muszę wspomnieć chociażby o holdingu spożywczym obiecanym w 2016 r. Gdyby był on wdrożony, dzisiaj nie mielibyśmy problemu z galopującymi cenami w sklepach. Muszę wspomnieć o ustawie o oddłużeniu gospodarstw rolniczych, która niby została uchwalona, a dalej mamy liczne licytacje gospodarstw, czy o zbierającej tragiczne żniwo w gospodarstwach rolników pandemii ASF.

Minister cyfryzacji wielokrotnie podkreślał, że należy zagwarantować obywatelom poczucie bezpieczeństwa, poczucie i świadomość tego, że państwo ten proces kontroluje, i jeżeli moglibyśmy mówić o jakimkolwiek zagrożeniu, to zagrożenia te są pod kontrolą. Przypomnę, iż w listopadzie 2019 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Minister cyfryzacji zaproponował w niej zapis dotyczący uruchomienia systemu informatycznego dotyczącego instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne. Minister cyfryzacji wielokrotnie przekonywał parlamentarzystów i społeczeństwo, iż system ten będzie umożliwiał każdemu obywatelowi sprawdzenie przez Internet poziomu promieniowania elektromagnetycznego w domach i w miejscach pracy. System miał rozwiać wątpliwości, czy stacje telekomunikacji przekraczają dopuszczalne - przypomnę, obecnie 100-krotnie podniesione - normy granicznego pola elektromagnetycznego w Polsce. Przypomnę, miało to miejsce przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk naukowych w Polsce wyrażających swój sprzeciw w licznych opiniach przedstawionych Ministerstwu Zdrowia w trakcie konsultacji społecznych dotyczących rozporządzenia. Niestety, do chwili obecnej system nie jest dostępny dla obywateli. Ponadto ustawą - tarcza antykryzysowa 2.0 w kwietniu br. zwolniono organy ochrony środowiska i samych operatorów telekomunikacyjnych z konieczności wykonywania pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w lokalach mieszkalnych i użytkowych, pozbawiając tym samym państwo jakiejkolwiek kontroli nad tym kluczowym dla bezpieczeństwa obywateli elementem środowiska. Wydaje się, że hasło: kontroli nie ma, promieniowanie hartuje - z kontroli NIK-u dotyczącej działalności organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej - jest teraz bardziej aktualne niż rok temu. Reasumując, proponowane rozwiązanie jest bardzo dobre, i dobrze, że zostało wdrożone, aczkolwiek powinno być wdrożone lata temu. Ale istnieje duża obawa związana z poufnością przekazywanych wrażliwych informacji, gdyż sytuacja może się powtórzyć - i rząd, jak mówi, że zrobi, to tylko mówi. Nasze poufne dane będą źle zabezpieczone, a system będzie działał dobrze, ale podobnie jak to miało miejsce z innymi wcześniej wdrożonymi systemami, będzie działał tylko tam. W imieniu koła Konfederacja pan poseł Michał Urbaniak.

Na mównicę również bardzo proszę w maseczce, panie pośle. Panie pośle, bardzo proszę o założenie maseczki. Panie pośle, ja bardzo pana proszę o założenie maseczki. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że łamie pan ustalenia związane z noszeniem maseczki na sali posiedzeń. Ustalenia Prezydium.

Dziękuję uprzejmie. Najwyższy czas, żeby taki projekt w ogóle trafił do Sejmu, dobrze, że to się dzieje, więc Konfederacja jak najbardziej przyklaskuje temu faktowi. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowywało własny projekt.

Dzisiaj w całym kraju trwają protesty rolników i są one przeciwko piątce. Nie przedstawił on też skutków ekonomicznych wprowadzanych regulacji. Projekt ustawy nie był konsultowany z rolnikami, organizacjami rolniczymi i nie przewidziano negatywnych konsekwencji wprowadzenia tych przepisów. Autorzy piątki dla zwierząt, dając miesiąc na zamknięcie produkcji i mgliste obietnice odszkodowań, likwidują de facto całą branżę. Przypomnijmy, że cykl hodowli trwa 2 lata. Po wejściu w życie ustawy zakazujemy też uboju rytualnego w Polsce, zarówno bydła, jak i drobiu. Nasze zapotrzebowanie na wewnętrzny, polski rynek jest na tyle niewielkie, że w tym momencie prowadzenie takiego biznesu w Polsce traci rację bytu. Chciałbym przypomnieć też, że rynki eksportowe, zdobywane przez lata, nagle będą dla nas zamknięte. Mówimy tu też o rynkach w Unii Europejskiej.

Rząd Zjednoczonej Prawicy chce też siebie w tym momencie pozbawić źródła dochodu z podatków. Polska jako największy producent drobiu w Unii Europejskiej sprzedawała 855 tys. t drobiu z uboju religijnego.

350 tys. gospodarstw domowych może w tym momencie stracić źródło dochodu, to robi właśnie Zjednoczona Prawica.

Część zakładów będzie musiała zamknąć się w ciągu miesiąca, bo to wynika z polskiego prawa, które chcecie uchwalić.

Zakaz skutecznie pozbawił także kredytów bankowych - banki boją się tego, co wydarzy się na rynkach związanych z rolnikami. Kryzys dotknie także rynek zbóż, pasz, odpłatną utylizację odpadów, przetwórstwo rybne, mleczne, mięsne, to np. był także pokarm dla norek, które chcecie teraz przenieść - na to wychodzi - gdzieś za granicę. Wspominam o tym, bo ignorujecie protesty ludzi, którym po prostu zabieracie chleb. W tym momencie wiemy, że ci ludzie mogą już zwijać swoje interesy, bo Zjednoczona Prawica uważa, że lepiej wprowadzać lewackie prawo. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do pytań.

Bardzo dziękuję, pani marszałek. Chciałem zapytać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość znowu nie dotrzymuje swoich obietnic wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość w 2015 r., jak i ostatnio, wygrało wybory, mówiąc o reformie sądownictwa, a w tej ustawie reforma sądownictwa właśnie w zakresie doręczeń elektronicznych ma wejść w życie dopiero za 9 lat. Dlaczego tak kluczowa dla polskiego społeczeństwa reforma znowu zostaje odłożona tak naprawdę chyba na nigdy, bo 9 lat to jest bardzo długie czekanie na sprawiedliwość? Dziękuję. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Procedowana ustawa jest niewątpliwie krokiem w dobrą stronę, gdyż formuła doręczeń z zasady zapewni szybki i wygodny sposób komunikacji pomiędzy obywatelami i urzędami. W ustawie czytamy, że osoby, które na wymianę korespondencji elektronicznej z różnych przyczyn nie będą jeszcze gotowe, dzięki usłudze hybrydowej otrzymają możliwość odbierania tradycyjnej przesyłki listowej. Mówiąc wprost, list w postaci elektronicznej zostanie dostarczony na pocztę, a ta wydrukuje go i dostarczy w postaci papierowej. W jaki sposób zostanie zapewniona w tym przypadku ochrona tajemnicy, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności informacji?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pytanie: Dlaczego usługa doręczenia cyfrowego będzie płatna? Jaki jest tego sens? Gdzie koszty? Pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Co najmniej 4 lata przespaliście. Dziś oferujecie Polakom ustawę, która będzie wchodziła przez 9 lat. Wszyscy mówicie cały czas, że mamy być równi wobec prawa. A tu okazuje się, że różne instytucje państwowe nie są równe wobec prawa.

A dzisiaj, panie ministrze, przez 9 lat chcecie wprowadzać to, co jest proste, jasne i czytelne.

Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek!

W zasadzie jest on słuszny - tzn. na podstawie orzeczenia sądowego albo aktu administracyjnego.

Natomiast uwagę zwraca to, że w myśl tego przepisu nikt nie musi wykazywać żadnego interesu związanego z dostępem do mojej skrzynki. Nikt nie musi uzasadniać np. wniosku o tryb udzielenia takiego dostępu. Co więcej, udzielenie takiego dostępu nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Jak państwo widzą treść tego przepisu w kontekście przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej precyzujących ochronę tajemnicy korespondencji? Dziękuję bardzo. Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska, kolejne pytanie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To jest ustawa, która ma na celu wykorzystanie najnowszych technologii dla usprawnienia państwa. Natomiast pytanie i obawy budzi to, że wykorzystuje się też najnowsze technologie i technikę do tego, by zwiększać etatyzm funkcjonowania państwa. Dlaczego, jakie jest uzasadnienie tego, że wskazuje się precyzyjnie tylko jeden podmiot - Pocztę Polską - do tego, żeby to realizował? To jest pierwsze pytanie. A drugie brzmi: W jaki sposób ministerstwo przewiduje zapewnienie prywatności korespondencji osób, do których będą dostarczane przesyłki w formie hybrydowej? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Mam bardzo krótkie pytanie, ono dotyczy właśnie konkurencji. Bo rzeczywiście sytuacja wygląda następująco: ta ustawa wprowadza de facto monopol na rynku doręczeń elektronicznych wobec jednego podmiotu. Po pierwsze: Dlaczego ten monopol? Jakie będą kierunki działań w celu zniwelowania przewagi konkurencyjnej i zapewnienia rzeczywistej konkurencji na rynku doręczeń elektronicznych? Bo ponoć trzeba będzie w ogóle za to płacić, za doręczenie maila. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Parlamentarzyści!

Ta praca przebiegała i przebiega bardzo sprawnie. Z pewnością ustawa wprowadzająca e-doręczenia w Polsce jest projektem rewolucyjnym, nie ewolucyjnym.

To naszym zdaniem powoduje przede wszystkim to, że nie tylko dokonamy rewolucji w komunikacji na linii państwo - obywatel, czego sobie życzymy oczywiście wszyscy, tak jak mówimy na tej sali. Chcemy, aby Polska jak najszybciej realizowała założenia chociażby „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która zakłada powszechną cyfryzację państwa.

Uważamy, że przede wszystkim te zmiany muszą być wprowadzone solidnie.

Jako Ministerstwo Cyfryzacji, a teraz dział informatyzacji, który będzie włączany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mamy oczywiście na uwadze bezpieczeństwo danych. Opieramy się chociażby na regulacjach unijnych, które są bardzo w tym zakresie rygorystyczne.

To wynika również z ducha czasu, który mamy przed sobą. Wszyscy w tym kierunku podążamy.

Bardzo bym prosił, aby nie przeszkadzać.

Kończąc, dziękuję raz jeszcze członkom podkomisji za tę pracę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643) Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 643. Zmiany mają charakter zasadniczy i ewolucyjny, a wzorowane są na rozwiązaniach działających od 20 lat w Estonii. Proponujemy, aby od stycznia przyszłego roku zaczął w Polsce obowiązywać tzw. estoński CIT, czyli ryczałt od przychodów spółek kapitałowych. Jest to taki sposób opodatkowania małych firm, który gwarantuje maksymalną promocję inwestycji i minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Na czym on polega? Obecnie dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jest zasadniczo w momencie jego powstania, czyli memoriałowo. Oznacza to, że podatnik rozpoznaje przychód w momencie sprzedaży, nawet jeśli nie otrzymał jeszcze zapłaty od kontrahenta. W systemie estońskim tak długo, jak zyski pozostają w firmie, nie zapłaci ona CIT-u. Podatek pojawi się tylko wtedy, gdy osiągnięty w firmie zysk zostanie wypłacony wspólnikom. Brak podatku i pozostawienie środków w firmie ma dla niej dwa pozytywne efekty: po pierwsze, wzmacnia jej płynność, a przez to odporność na kryzysy, daje jej swoistą finansową poduszkę bezpieczeństwa, po drugie, pozostawia jej środki finansowe na dokonywanie inwestycji. Inaczej niż przy innych ulgach podatkowych nie ma tutaj ograniczeń - przedsiębiorca wydaje środki na to, co jest mu najbardziej potrzebne. Jest to sposób rozliczenia, który jest bardzo tani. Brak cyklicznej - comiesięcznej, cokwartalnej i corocznej - zapłaty podatku to również brak szeregu obowiązków, a przez to duża oszczędność czasu dla firm. Podatnik nie będzie zmuszony do prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji dla celów podatkowych i księgowych. Nie będzie liczył kosztów podatkowych i amortyzacji. Skorzysta również z ułatwień w zakresie raportowania MDR. Brak szeregu obowiązków oznacza dla firm niższe koszty obsługi prawnej. W Polsce samodzielnie, bez pomocy doradcy CIT rozlicza tylko 20% firm. W Estonii jest ich trzy razy więcej, ponad 60%. Czas rozliczenia CIT-u wynosi tam średnio 5 godzin rocznie, a w Polsce prawie 60. W sumie system estoński to potencjalna oszczędność prawie 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie przez polskie firmy na rozliczenie podatku CIT. Gospodarcze efekty reformy w Estonii były bardzo pozytywne. Z perspektywy mikroekonomicznej zmniejszyło się zadłużenie i wzrosła płynność przedsiębiorstw. W Polsce te rezultaty mogą być jeszcze lepsze, choć już osiągnięcie efektów podobnych do tych z Estonii byłoby dla polskiej gospodarki bardzo dużym sukcesem. Estonia była pierwszym państwem, które wdrożyło ten nowoczesny sposób opodatkowania. Jej drogą wkrótce podążyły kolejne kraje, m.in. Gruzja i Łotwa. Od przyszłego roku do tej grupy państw dołączy Polska. Proponowane przez nas rozwiązanie nie różni się od swojego estońskiego pierwowzoru. i taniość, pozostają takie same. W realizowanej w przyszłym roku pierwszej fazie wdrożenia w Polsce systemu estońskiego będzie on dostępny dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że warunki skorzystania z estońskiego CIT-u określone zostały bardzo inkluzywnie. Już w pierwszym roku jego działania będzie on otwarty dla ponad 200 tys. firm, czyli ponad 90% aktywnie działających w Polsce spółek kapitałowych. Zainteresowanie tym rozwiązaniem będzie duże, ponieważ estoński CIT jest rozwiązaniem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Zapewnia nie tylko możliwość odroczenia podatku na poziomie spółki, ale również niższe opodatkowanie na poziomie wspólnika i korzystne zasady rozliczenia podatku przy wyjściu z systemu estońskiego. Projekt jest efektem intensywnych konsultacji z przedsiębiorcami. W toku prac rządowych został tak ukształtowany, żeby był jak najbardziej korzystny, otwarty i dostępny dla jak największej liczby firm. Stąd niedawne zmiany w projekcie, m.in. dwukrotne podniesienie limitu przychodowego z 50 mln zł do 100 mln zł, stworzenie dodatkowych zachęt do inwestowania w zatrudnienie, do inwestycji w kapitał ludzki, a także zastrzyk środków na inwestycje poprzez możliwość rozliczenia zakumulowanej straty na 2 lata wstecz. Proponowane zmiany zwiększą wolumen inwestycji w polskiej gospodarce, zwiększą konkurencyjność i dokapitalizują sektor MŚP. Skorzystają przedsiębiorcy, którzy z uwagi na mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego cierpią z powodu niedoboru środków na realizację inwestycji. Przez to nie mogą rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem i znajdują się w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o konkurencyjność. Nowy model opodatkowania będzie dla tych firm elastycznym narzędziem, które rozbije barierę braku finansowania i wyrówna szanse mniejszych przedsiębiorców na rynku. Będzie to stanowiło impuls dla rozwoju całej gospodarki.

Zaproponowane w projekcie zmiany w pierwszym roku obowiązywania zmniejszą dochody sektora finansów publicznych o około 5600 mln zł. Bazując na doświadczeniach Estonii, przyjęto spadek dochodów tylko w pierwszych 3 latach obowiązywania nowej regulacji, natomiast szacuje się, że w kolejnych latach projektowane rozwiązania wpłyną pozytywnie, zwiększą dochody sektora finansów publicznych. Zakłada się, że zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie projektu ustawy w wersji zaproponowanej przez rząd. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Andrzej Szlachta. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 643. Celem wprowadzonych lub modyfikowanych przepisów jest wdrażanie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych wzorowanego, jak już pan minister powiedział, na rozwiązaniach stosowanych już od 20 lat w Estonii. W projekcie zaproponowano dwa alternatywne warianty opodatkowania na nowych zasadach, bez możliwości ich łączenia.

Jest to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Wariant drugi wprowadza specjalny fundusz inwestycyjny, który umożliwia szybsze rozliczenia amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych zasad opodatkowania. Oba warianty mają charakter proinwestycyjny, a tym samym wspierający wzrost gospodarczy. Projekt ustawy adresowany jest do grupy przedsiębiorców, która ma słabszą pozycję konkurencyjną i mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji. Są to podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a które chcą realizować proinwestycyjną strategię rozwoju w szczególności poprzez wzrost zatrudnienia oraz systematycznie ponoszone nakłady inwestycyjne. Przedsiębiorstwa te ze względu na brak powiązań kapitałowych napotykają na barierę dostępu do finansowania. Według badań OECD co trzeciemu polskiemu podmiotowi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie udaje się pozyskać potrzebnego finansowania dłużnego. Nie mogą one, jak w przypadku podmiotów prowadzących działalność w grupach kapitałowych, uzyskać finansowania od spółek powiązanych czy pozyskać gwarancji od spółek z grupy w zakresie uzyskania takiego finansowania od podmiotów sektora bankowego. Omawiany projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w pięciu aktach prawnych: ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawie o rachunkowości i ustawie - Kodeks karny skarbowy. Jeżeli chodzi o ustawę o podatku CIT, nowy przepis umożliwia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej wybór opodatkowania ryczałtem. Szczególne zasady opodatkowania ryczałtem oznaczają znaczną zmianę dotychczasowych zasad rozliczania. Zaproponowane zmiany zapewniają opodatkowanie rezerw i odpisów aktualizujących u podatników, którzy zakończyli opodatkowanie ryczałtem. Projekt zmian w podatku CIT przewiduje cztery podstawy opodatkowania: dochód z tytułu podzielonego zysku, dochód z tytułu ukrytego zysku oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dochód z tytułu zmiany wartości majątku oraz dochód z tytułu zysku netto. W ustawie o podatku PIT zachowane zostanie opodatkowanie podatkiem od dochodów od osób prawnych w momencie wypłaty zysku przez spółkę oraz podatkiem od dochodów osób fizycznych z tytułu odpowiadającego rodzajowi dokonanej przez spółkę wypłaty, np. dywidendy, odsetek, wynagrodzenia. W ustawie o rachunkowości wprowadza się obowiązek przekazywania informacji w ramach sprawozdania finansowego o wszystkich dochodach z tytułu ukrytych zysków. W ustawie - Ordynacja podatkowa projekt przewiduje zmiany w zakresie regulującym przedstawienie zobowiązania podatkowego. W ustawie - Kodeks karny skarbowy projekt przewiduje odpowiedzialność karnoskarbową podatnika, który nie składa spółce oświadczenia albo składa je po terminie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze przedmiotowy projekt ustawy w dalszych pracach legislacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Wojciech Saługa. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! CIT może i estoński, ale piekiełko regulacyjne na pewno polskie. Mówił pan tu z takim dużym entuzjazmem o Estonii właśnie, ale jak się wczytamy w ten projekt, to tej Estonii jest dość mało. W Polsce powszechnym się nie wydaje, ponieważ większość przedsiębiorstw w Polsce to nie spółki kapitałowe, a ten projekt dotyczy tylko spółek kapitałowych - wiadomo, jak chodzi o CIT, ale to nie będzie rozwiązanie masowe dla przedsiębiorców, a raczej bym powiedział: ekskluzywne.

Jest 15 wymogów, które trzeba spełnić, żeby z tego CIT-u estońskiego móc skorzystać. Nakłaniacie tym rozwiązaniem. Po co chcecie zmuszać ludzi do tego, żeby zatrudniali, jak np. nie muszą?

Raz, że to dość skomplikowane, natomiast też istnieje ryzyko, że przedsiębiorca nie będzie inwestował tyle, ile mu potrzeba, tylko będzie inwestował tyle, ile potrzeba, żeby móc się do tego CIT-u załapać. Też słyszymy o przeinwestowaniach, o za dużym zatrudnieniu. Prostota, powszechność. 25 stron przepisów, 50 stron komentarza.

W klasyfikacji łatwości prowadzenia biznesu jesteśmy bardzo nisko. Mamy szansę tą ustawą spowodować, że przynajmniej w tym obszarze będzie łatwo, właśnie będzie tak jak w Estonii.

Sam tego po prostu nie udźwignie, nie zrozumie. W Estonii jest rozwiązanie 20% i dość. Wypłata dywidendy 20% i nie płaci się już potem od dywidendy PIT-u. Komplikujemy ten system. Z entuzjazmem jeszcze raz mówię - pan minister mówił o Estonii - my wszyscy z entuzjazmem też czekamy na te estońskie rozwiązania, ale jak się wczytamy, to tu nie ma Estonii.

Byle to nie były błędy, które my tu popełnimy, wdrażając takie prawo.

Za dużo. I będziemy namawiać pana ministra, rząd do tego, aby w dalszych pracach, jakże potrzebnych, bo to rozwiązanie jest potrzebne, jest oczekiwane, tak pracować, żeby ten CIT estoński, polski był przyjazny i żeby te przepisy [[Dzwonek]] uległy maksymalnemu uproszczeniu w dalszym procedowaniu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko klubu parlamentarnego Lewica przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Anita Sowińska. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność zaprezentować stanowisko klubu Lewicy w sprawie druku nr 643 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzy się nasza gospodarka, jest mały kapitał własny polskich firm oraz związana z tym niewielka skłonność do wydawania pieniędzy na inwestycje. Jest to oczywiście problem znany nie od dziś, który sprawia, że polskie firmy nie inwestują w wystarczający sposób w innowacje i środki trwałe i przez to są mniej konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Drugim problemem, który również występuje od wielu lat, sprawą, która blokuje polskie firmy, jest skomplikowany system podatkowy wymagający ciągłego śledzenia zmian w przepisach i prowadzenia żmudnej ewidencji podatkowej. Sposobem na usunięcie obu tych barier może być estońska wersja podatku od przedsiębiorstw. Według tej koncepcji CIT odprowadzany jest nie od wypracowanego przez firmę zysku, ale dopiero w momencie wypłaty tego zysku z firmy w formie dywidendy. Czyli dopóki pieniądze pozostają w firmie, a zyski są inwestowane np. w rozwój, dopóty płacenie podatku CIT nie jest wymagane. W projekcie ustawy przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania do wyboru przez przedsiębiorcę. Wariant pierwszy to ryczałt od dochodów spółek, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego, polegający na znacznej modyfikacji zasad opodatkowania - m.in. zmianie ulega moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, a także stawki podatkowe. Wariant drugi to specjalny fundusz inwestycyjny, który umożliwia szybsze rozliczanie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. Co do zasady proponowane zmiany w ustawie, którą omawiamy, są pozytywne, ponieważ nie tylko obniżają wysokość opodatkowania, ale również zachęcają polskie firmy do inwestowania oraz upraszczają sposób rozliczania podatków. Jak wskazują doświadczenia estońskie, ale również innych krajów, rozwiązania te mają proinwestycyjny charakter i prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstw, poprawy ich płynności, zdolności kredytowej i produktywności, a tym samym wpłyną pozytywnie na wzrost gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki. Trzeba jednak wskazać, że zaproponowane rozwiązanie ma również wady. Wadą jest to, że nie będzie to rozwiązanie dostępne dla wszystkich firm, a jedynie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, które spełniają wszystkie kryteria łącznie, tj. nie posiadają udziałów w innych podmiotach, zatrudniają co najmniej trzech pracowników oprócz udziałowców, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej oraz które wykazują nakłady inwestycyjne. Zatem nie będą mogli skorzystać z tej preferencji podatnicy PIT, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ani też spółki, których udziałowcem jest inna spółka, czy to krajowa, czy zagraniczna. Musimy zdawać sobie sprawę, że takie rozwiązanie będzie prowadzić do zachwiania konkurencyjności w odniesieniu do przedsiębiorstw. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania w ciągu kilku pierwszych lat wpłyną na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

To dużo, należy się więc zastanowić, jak zrekompensować samorządom mniejsze wpływy do budżetu, zwłaszcza w pierwszych latach działania nowych regulacji podatkowych. Samorządy już teraz są w bardzo trudnej sytuacji finansowej nie tylko ze względu na pandemię, ale również ze względu na wzrost nakładów na edukację i ochronę zdrowia. Niestety za nowymi obowiązkami nakładanymi przez rząd nie idą dodatkowe wpływy z budżetu, trzeba to więc uwzględnić w nowej ustawie budżetowej. Podsumowując, Lewica popiera dalszą pracę w Komisji Finansów Publicznych nad tą ustawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 643.

Dotyczy wprowadzenia dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania, tj. systemu wzorowanego na rozwiązaniu estońskim, wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na znacznej modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umożliwi podatnikom szybsze rozliczanie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczanie podatkowe. Tzw. estoński CIT to nowoczesny sposób opodatkowania, który pozwala firmom inwestować i ograniczyć do minimum formalności przy rozliczaniu podatków. Zgodnie z tym rozwiązaniem podatek zostanie nałożony na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku. Oznacza to, że środki, które zostaną w firmie, będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy. Estoński CIT ma też przeciwdziałać negatywnym następstwom koronawirusa, czyli przyczynić się do zapewnienia stabilnych miejsc pracy i zwiększenia zatrudnienia. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Nowe rozwiązanie w polskiej wersji ma dotyczyć wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł. Dotyczy to ok. 90% polskich firm. Warunkiem skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u będzie zatrudnianie co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać nowy system opodatkowania na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 4-letnie. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim - czwartym - roku korzystania z tego systemu przedsiębiorca wciąż będzie spełniał wymagane kryteria. Z pewnością procedowany projekt przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw, tak jak wspomniałem: likwidacja barier rozwojowych, wzrost kapitałów własnych, poprawa płynności finansowej, mniej formalności, ale trzeba też nieco dziegciu do tego dołożyć naszym zdaniem, zdaniem klubu Koalicji Polskiej, mianowicie bardzo mocno wyartykułowany został głos w sprawie tego projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, które to ciało zwróciło uwagę na to, że niestety mamy, podobnie jak przy zerowym PIT w nieodległej przyszłości, również negatywne skutki, jeśli chodzi o finanse samorządów, jakie wiążą się z tym projektem. Jak wszyscy doskonale wiemy, finanse samorządów są już dzisiaj na skraju wydolności i bardzo ważne byłoby, myślę, na tym etapie - i my jako klub będziemy tego się domagać - żeby wprowadzić jakąś formę rekompensaty tych uszczuplonych dochodów samorządów. Co do zasady są to bardzo dobre rozwiązania dla przedsiębiorców, ale nie możemy po raz kolejny realizować szczytnych skądinąd założeń kosztem uszczuplania finansów i dochodów samorządowych. Myślę, że to jest główny argument, który w naszym przypadku będzie ważył na definitywnym poparciu tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Rozumiem, że prowokacyjnie oczywiście bez maseczki. Odpowiadają za protokół, wykonują swoje obowiązki służbowe, a pan po prostu bezczelnie narusza ich bezpieczeństwo. Rozumiem, że z pełną świadomością będzie pan chciał kontynuować swoje wystąpienie bez maseczki, tak? Przepraszam, panie pośle, jeszcze nie skończyłam.

Rozumiem, że pan zna. W związku z tym, panie pośle, chciałabym stwierdzić, że narusza pan spokój i porządek na terenie Kancelarii Sejmu, sali posiedzeń, co wiąże się z art. 22b.

Myślę, że zna pan konsekwencje. Bardzo chętnie.

Wczoraj wszystkie media zajmowały się prezesem Kaczyńskim, tym, że nie miał maseczki na zaprzysiężeniu, że zdjął rękawiczkę, wraz z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzisiaj pani marszałek wespół w zespół z tresowaną opozycją zajmuje się Konfederacją i maseczkami.

Nie. ...czasu, który musiałem zmarnować na polemizowanie z panią na tematy zastępcze. Mam tutaj raport Stowarzyszenia KoLiber, autorstwa Macieja Letkiewicza, na temat estońskiego CIT-u, a tak naprawdę na temat polskiego CIT-u, który powinien się nazywać antyestońskim CIT-em, gdyż takim w zasadzie jest. Pan premier Morawiecki ma taką zdolność: jest anty-Midasem podatkowym.

Co to jest estoński CIT? Pan premier mówi, że to jest rozwiązanie innowacyjne. Dzięki temu mają jeden z najprostszych systemów podatkowych, poświęcają na rozliczenia podatkowe sześć razy mniej czasu - a na rozliczenie podatku dochodowego dziesięć razy mniej czasu - niż Polacy. Podatek prosty jak budowa cepa: dopóki spółka nie wypłaca dywidendy, dopóty nie płaci podatku dochodowego. To jest uproszczenie przepisów, a w Polsce mamy rozbudowanie całej masy regulacji, bo w Polsce dochodzą dodatkowe elementy: musi być trzech pracowników z wyłączeniem udziałowców, muszą być odpowiednie rodzaje przychodów, nieprzekraczane limity przychodów, spółka nie może mieć udziałów w innych spółkach i udziałowcy tej spółki nie mogą być spółkami, muszą być odpowiednio zwiększane nakłady inwestycyjne, odpowiedni poziom. Szanowni państwo, w ten sposób, jeżeli wykluczają państwo duże firmy, które tak naprawdę zrobią różnicę, bo je stać na zagranicznych doradców, one uciekają z tym podatkiem dochodowym. Państwo sprawiają, że praktycznie nikt nie będzie korzystał z tego bardzo skomplikowanego rozwiązania, wymagającego wydania kupy pieniędzy na doradców podatkowych, bo ono jest zbyt trudne. Osobiście w 2016 r. byłem już w Ministerstwie Finansów na spotkaniu z wiceministrem finansów i przedstawiłem mu koncepcję podatku estońskiego. Na pierwszym spotkaniu powiedział, że to jakieś bajki. Spotkałem się z nim drugi raz, wówczas powiedział mi: rzeczywiście koncepcja bardzo ciekawa, ale my nie mamy teraz czasu, bo my musimy dociskać vatowców, poza tym w pierwszym okresie to będzie kosztowało. No i państwo pracowali 4 lata na to, by tak ten system skomplikować, żeby móc powiedzieć: wprowadzamy estoński CIT, ale w rzeczywistości nie wprowadzić nic. Tak wygląda państwa polityka podatkowa - coraz więcej podatków, coraz bardziej skomplikowany system podatkowy. Traci na tym gospodarka. Proszę tego nie nazywać estońskim CIT-em. Jeśli chodzi o te uwagi, ktoś w ministerstwie przeczytał na pewno ten raport, bo dwie drobne zmiany zostały wprowadzone - rzeczywiście limit delikatnie podniesiony, rzeczywiście definicja pracownika delikatnie zmieniona. Ale dalej nie jest to estoński CIT. Dziękuję bardzo.

Witam państwa na dzisiejszym balu maskowym. Jeszcze miesiąc temu wirusy nam nie szkodziły, teraz znowu nam szkodzą. Przyjmijcie do wiadomości, że jesteście śmieszni z tą maskaradą. Nie zostało mi wiele czasu, więc krótko. Ustawa, która wprowadza dodatkowe. Ta ustawa wprowadza różne wymogi, w związku z którymi wielu przedsiębiorców, zamiast skupić się na pracy na rzecz gospodarki, na rzecz wytwarzania dóbr i usług dla konsumentów, będzie się skupiało na tym, jak spełnić te wymogi i jak tak namieszać w firmie, jak tak przekształcić swoją działalność, żeby łapać się na jakieś wymogi.

Przechodzimy do pytań. Bardzo proszę. Przepraszam, panie pośle. Dziękuję. Panie Ministrze! Właściwie jaka jest tendencja rządu, jeśli chodzi o reformy podatków? Chcecie z jednej strony podwyższać, z drugiej - obniżacie. W tej kwestii rzeczywiście, jeśli to finalnie się skończy, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z obniżenia, a z drugiej strony wprowadzacie. Za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnym podatku CIT dla spółek komandytowych. Panie ministrze, oczywiście ta ustawa na przedsiębiorców nakłada pewne zobowiązania, trzeba spełnić 15 warunków, żeby można było w ogóle skorzystać z tego przywileju i wpisania się w to, trzeba utrzymać ludzi, trzeba realizować inwestycje. To pana zdaniem ilu przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tej ustawy? Ile i jakie konkretne środki finansowe będą mogli zaoszczędzić ci przedsiębiorcy? Wszyscy wiemy dobrze, że samorząd na tym na pewno będzie tracił, bo [[Dzwonek]] korzystał z tego podatku. Pytanie kolejne: Jak macie zamiar rekompensować te wpływy samorządów, które one utracą, jak ta ustawa wejdzie? Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Koalicja Obywatelska. Mamy połączenie?

Nie wiem, czy mnie słychać. Bardzo proszę o zadanie pytania. Dziękuję. Wysoka Izbo! W wystąpieniu pana ministra usłyszeliśmy bardzo dużo entuzjazmu i był to entuzjazm godny komiwojażera. Ale chciałbym zapytać o konkrety, bo planujecie państwo wręczyć bardzo kosztowny prezent spółkom kapitałowym, natomiast ja chciałbym usłyszeć, jakie są dowody, że ten prezent podniesie poziom inwestycji w Polsce. Podkreślam: w Polsce w 2020 r., bo my mamy inną gospodarkę i inną strukturę finansowania inwestycji, niż miała je Estonia 20 lat temu. To jest diablo kosztowna propozycja, która wyrwie i z budżetu centralnego, i z budżetów samorządów grube miliardy złotych. Czy warto, żeby tych pieniędzy na szpitale, na edukację było mniej? Chciałbym zobaczyć wiarygodne analizy, a nie usłyszeć entuzjazm rodem z broszurek lobbystów albo z podręcznika dla komiwojażera. Tych wiarygodnych analiz nie zobaczyliśmy. Tymczasem (Dzwonek) kapitał w Polsce ciągle jest opodatkowany dużo niżej niż praca, a jeżeli państwo wdrożycie tego typu rozwiązanie, to ciężar budżetu w jeszcze większym stopniu będzie się opierać na pracownikach. Tak działo się wszędzie, gdzie wprowadzano rozproszone opodatkowanie zysku. Chciałbym zapytać, jak chcecie państwo temu zapobiec, i prosić. Pan poseł Marek Rutka, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zacytuję uwagę Fundacji Startup Poland: Wprowadzony w projekcie wymóg zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej trzech osób zamyka możliwość stosowania estońskiego CIT-u przez wiele start-upów, zwłaszcza małych, które nie spełniają tego kryterium. Koniec cytatu. Stąd też pytanie. Zamysł i idea wprowadzenia estońskiego CIT-u są godne rozważenia, natomiast dlaczego w trakcie konsultacji społecznych start-upy oraz organizacje reprezentujące tego rodzaju podmioty nie miały większej możliwości wnoszenia uwag? Przecież to dzięki start-upom oraz małym, innowacyjnym przedsiębiorstwom pojawił się temat implementacji estońskiego CIT-u, w przypadku którego to dla tego rodzaju przedsiębiorstw wprowadzono największe ulgi i ułatwienia, zaś w polskim klonie CIT-u znalazły się obostrzenia i przeszkody dla tego rodzaju działalności. Innymi słowy, rząd starał się bardzo, a wyszło jak zwykle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Z roku na rok obserwujemy coraz mniejsze inwestycje wśród małych przedsiębiorstw.

Dlaczego nie pozwalamy wejść do tego systemu wszystkim, tylko komplikujemy go do granic możliwości, tak żeby zacieśniać tę możliwość korzystania z przyjaznych rozwiązań? Druga rzecz. Koszty wdrożenia tego pan minister szacuje na ponad 5 mld zł. Z CIT-u korzystają samorządy, głównie samorządy wojewódzkie. Jaki uszczerbek w budżetach samorządów wojewódzkich w związku z tym przewidujecie?

Wysoka Izbo! Procedowana ustawa w takim kształcie jak obecny nie ma nic wspólnego z estońskim CIT-em. Podatek ten nakłada obowiązek oddania pieniędzy fiskusowi w chwili wypłacenia zysku. Jeśli zostanie on przeznaczony na inwestycje, podatku od niego nie trzeba będzie płacić.

Od tej dywidendy fiskus pobiera swoją część w postaci PIT-u. Nowe rozwiązanie jest po części korzystne dla małych przedsiębiorców, niemniej jednak w związku z tym projektem po raz kolejny uszczuplone zostaną dochody jednostek samorządu terytorialnego, o czym moi przedmówcy już wspominali. Może idea tej ustawy jest dobra, lecz dla jednostek samorządu terytorialnego jest ona niekorzystna.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana wiceministra, który przeczytał nam z kartki walory estońskiego CIT-u oraz przedstawił nam, także z kartki, zalety tego estońskopodobnego produktu, PiS-owskiego CIT-u. Jakie są podobieństwa, ile jest tych podobieństw i ile jest różnic między tymi dwoma różnymi systemami? Chciałbym także pana ministra zapytać, która z branż najchętniej skorzysta z tego waszego estońskopodobnego produktu, PiS-owskiego CIT-u i jaki będzie miało to wpływ na budżety chociażby samorządowców. Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ja się zgodzę z tymi głosami, które dotyczyły nazywania nowego podatku estońskim, jakoby był kopią tamtego rozwiązania. To jest oczywista bzdura i takie intelektualne oszustwo. Oczywiście jest to krok, panie ministrze, w dobrą stronę, ale w takim typowo polskobiurokratycznym, znanym nam stylu i wydaniu.

Eksperci oceniają, że nawet z tej grupy 200 tys. firm tylko część z uwagi na te obciążenia biurokratyczne będzie chciała z tego korzystać. Dlaczego wykluczono spółdzielnie? Przecież mogłyby spokojnie z tego korzystać. Dlaczego PiS wyklucza [[Dzwonek]] z tej formy opodatkowania firmy innowacyjne, gdzie udziałowcami są np. fundusze? Często te firmy innowacyjne potrzebują kapitału, a ten kapitał oferują fundusze. Byłaby to naturalna przestrzeń do zastosowania tego opodatkowania, a państwo to wykluczacie. Dlaczego? Dziękuję bardzo. Panie pośle Braun, proszę nie pochylać się nad pracownikami, którzy są zmuszeni do kontaktowania się z panem, a jest pan bez maseczki. Czy pan słyszy, panie pośle Braun?

Konsekwencje pan zna. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek Gosiewska, narusza pani powagę tej Izby swoim istnieniem w tej Izbie i swoim tutaj dzisiaj zachowaniem. Proszę przyjąć do wiadomości... 5 minut przerwy, bardzo proszę.

Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czysto teoretycznie ta ustawa oczywiście idzie w dobrym kierunku. Estoński CIT jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem, ale polski estoński CIT niestety niezbyt wiele ma z nim wspólnego. Polski przedsiębiorca musi spełnić łącznie 15 warunków, o których wiele osób mówiło. Czemu w ogóle z VAT, czemu nie netto? Udziałowcami mogą być tylko osoby fizyczne, tak samo spółka nie może mieć udziałów w innych spółkach. Wiele poważnych spółek inwestuje w inne spółki. Konieczność inwestowania w środki trwałe. Tym samym wykluczacie państwo branże: szkoleniową, doradczą, konsultingową, finansową. Więc czemu to robicie? No i na koniec de facto 24% odsetek po 3 latach, jeżeli nie uda się spełnić któregoś z tych warunków. Który przedsiębiorca to zaryzykuje? No bo jest troszeczkę tak, że ogłaszacie teoretycznie dobre rozwiązanie, a następnie tworzycie tyle regulacji, tyle ograniczeń, [[Dzwonek]] że wykluczacie z niego prawie wszystkich. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Państwo z Ministerstwa! Idea podatku estońskiego to jest idea, która ma upraszczać system i zwiększać inwestycje firm. To jest idea. Dobra idea. Natomiast to, co państwo przygotowaliście, to jest slogan, który nie ma nic wspólnego z tą pierwotną ideą. Gdybyście porozmawiali z polskimi przedsiębiorcami, to wiedzielibyście, że największą barierą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce jest nadmierna regulacja. Ta ustawa jest przeregulacyjna. Pytanie pierwsze: Czy daliście do skonsultowania tę ustawę panu ministrowi Gowinowi, który kiedyś zajmował się deregulacją?

Pani poseł Monika Rosa, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Kiedy pan premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Polska stanie się idealnym miejscem do rozwijania biznesu, mówił o wprowadzeniu tzw. podatku estońskiego. Największym atutem estońskiego CIT-u jest jego prostota. Od 20 lat przepis stanowi, że wszystkie dochody spółki są nieopodatkowane tak długo, jak spółka nie wypłaca dywidendy jej właścicielom. Natomiast to, co państwo proponujecie, ma niestety niewiele wspólnego z tym estońskim CIT-em. Rozwiązania, które proponujecie, są bardzo skomplikowane. Polski przedsiębiorca, aby móc skorzystać z nowej formy opodatkowania, będzie musiał spełnić łącznie kilkanaście warunków. Bardzo proszę o informacje, dlaczego państwo tak mocno skomplikowaliście bardzo proste rozwiązanie i ilu przedsiębiorców wykluczycie z możliwości skorzystania z tego nowego podatku. Jest tu dość spora niespójność proponowanych przepisów. Dość daleko nam będzie do Estonii, jeśli chodzi o konkurencyjność systemu podatkowego. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Z oceny skutków regulacji, o których mowa w uzasadnieniu ustawy, wynika, że samorządy terytorialne, zwłaszcza samorządy powiatowe i wojewódzkie, stracą w najbliższych latach, najbliższych 3 latach, ponad 3300 mln zł.

W ten sposób państwo świadomie ograniczacie szanse rozwojowe społeczności powiatowych, społeczności lokalnych. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość.

Panie Ministrze! Niewątpliwie ten projekt ustawy jest dedykowany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Te podmioty będą beneficjentami tego projektu ustawy. Ale z drugiej strony w dyskusji pojawiły się krytyczne uwagi dotyczące wpływu skutków tej ustawy na sektor finansów publicznych, a w szczególności na samorządy. Dlatego bardzo proszę pana ministra o przedstawienie - wiem, że nie jest to łatwe, bo trudno precyzyjnie oszacować liczbę tych podmiotów, nie wiadomo tego - ile podmiotów z tego skorzysta, chodzi o jakieś takie wyważone proporcje, żebyśmy tego nie demonizowali, mówiąc, że przez to upadną samorządy. Czy inaczej to się kształtuje? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wiele słów padło już na temat uszczuplonych budżetów województw.

To jest pytanie, które chciałem zadać.

Pani Marszałek!

Ale troska o samorząd i jego kondycję jest obecna w tej Izbie, i to od lat.

Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Czy pan wie, co to jest wyrób czekoladopodobny? Państwo namnożyli przeszkód i zrobili swoisty tor przeszkód, aby przedsiębiorca nie skorzystał, a państwo mieli się czym pochwalić. Nie będę powtarzała tego, o czym mówił pan poseł Saługa i wszyscy krytycznie odnoszący się do tego projektu. To pierwsze. A drugie: pan może sobie nie przypomina, bo nie był pan w rządzie, ale kiedy Platforma Obywatelska zaproponowała rozwiązania dotyczące janosikowego, pierwszy był samorząd województwa podkarpackiego, który mocno protestował, jak tracił 30 mln. Dzisiaj straci 250 i nie słyszę protestu. Z Podkarpacia nie słyszę protestu. Czy i jakie samorządy do państwa napisały protest, aby państwo im to zrekompensowali? Wtedy będziemy widzieli, czy państwo sami tak chcecie robić i czy samorządy spolegliwie przyjęły państwa rozwiązanie. Dziękuję bardzo, pani poseł. I bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana ministra Jana Sarnowskiego. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Czy w rozwiązaniu proponowanym przez nas jest mało Estonii? Oczywiście, że nie.

Czy warunki wejścia w system estoński są skomplikowane? Warunki są przejrzyste, inkluzywne, takie, które sprawdzi każdy zatrudniony w firmie księgowy praktycznie od ręki. Gdyby ten podatek wdrożono w połowie bieżącego roku, natychmiast mogłoby z niego skorzystać 40 tys. zarejestrowanych w Polsce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przy drobnych zmianach struktury prowadzenia działalności np., zatrudnieniu przynajmniej jednego pracownika, mogłoby z niego skorzystać 200 tys. firm, czyli ponad 90% aktywnie działających w Polsce spółek komandytowych. Praktycznie każda branża, która jest zainteresowana rozwojem prowadzonej przez siebie działalności. Zauważmy: tutaj warunkiem jest nie tylko zwiększenie wolumenu środków trwałych, ale również inwestycje w kapitał ludzki, stąd zainteresowane będą zarówno branże produkcyjna, przemysłowa czy np. spożywcza, jak i branże usługowe, agencje reklamowe, usługi IT, a nawet firmy ochroniarskie. Przede wszystkim z 20-letniego doświadczenia Estończyków. To, co wdrożyliśmy, jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Finansów z Ministerstwem Finansów Estonii, które zwracało nam uwagę na trzy problemy, tzw. trójkąt bermudzki estońskiego CIT-u, a mianowicie: brak wpływu na dużych graczy, którzy nie zaczęli więcej inwestować, nieprecyzyjność wsparcia firm oraz nieszczelność systemu. Od wdrożenia tego systemu jak grzyby po deszczu w Estonii zaczęły się pojawiać spółki wydmuszki, które służyły do optymalizacji podatkowej, często międzynarodowej, agresywnej przez duże międzynarodowe koncerny. W Polsce chcemy tego uniknąć. Chcemy wdrażając system estoński w formule pilotażowej w przyszłym roku na pierwszym etapie jego wdrożenia, ograniczyć jego zastosowanie do tych firm, które najbardziej go potrzebują, a tak się składa, że będzie to aż 90% działających w Polsce spółek kapitałowych. Właśnie po to, żeby nie powstawały w Polsce firmy tak naprawdę nieistniejące, służące tylko międzynarodowym optymalizacjom, żeby nie było spółek wydmuszek, a także, żeby firmy, które z tego korzystają, działały realnie i żeby wejście w system estoński, oszczędność na podatku wiązała się z rzeczywistym, efektywnym wsparciem polskiej gospodarki, w tym zwiększeniem zatrudnienia. Pamiętajmy: nie mówimy już tutaj tylko o zwiększeniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tylko właśnie wsłuchując się w potrzeby sektora małych i średnich firm, w potrzeby start-upów, warunek ten został zmodyfikowany. Teraz wystarczy zatrudnienie każdego rodzaju skutkujące oskładkowaniem pracownika. Czy przepisy są długie? Warunki pozostawania w systemie estońskim opisane są tylko na pięciu stronach i to jest pięć stron, których powinien się nauczyć każdy przedsiębiorca, który jest w systemie estońskim, bo tylko z nich będzie korzystał, a nie z 278 stron, z których korzystać musi dzisiaj. Jakie są dowody, że to rozwiązanie przyniesie dobre skutki? Tutaj bazujemy nie tylko na badaniach dotyczących Estonii, ale również Łotwy, również Gruzji, również innych państw, w których funkcjonują podobne sposoby wspierania małego i średniego biznesu: niemieckie, austriackie czy węgierskie.

To są tylko przykłady, ale to są przykłady pokazujące, że te kraje, w których funkcjonuje tego rodzaju sposób wsparcia inwestycji dokonywanych przez firmy z sektora małych i średnich firm, radzą sobie nie tylko zdecydowanie lepiej niż Polska, ale też lepiej niż średnia unijna. Co do samorządów, to rzeczywiście nie przewidziano rekompensaty za spadek wpływów.

To jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby dać firmom maksymalnie korzystny sposób opodatkowania, który będzie wspierał zatrudnienie, który będzie wspierał inwestycje i który (Dzwonek) będzie również dawał firmom tę poduszkę bezpieczeństwa, która uchroni je przed ewentualnym wypadnięciem z rynku w trakcie trudności gospodarczych, które mogą przeżywać w kolejnych miesiącach. Pamiętajmy, co mówi nam przykład estoński. Z CIT-u rzeczywiście w pierwszym roku wpływów jest mniej, natomiast wpływy z PIT-u rosną właśnie poprzez wzrost zatrudnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 643, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Jana Sarnowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Szanowna Pani Marszałek! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 642. Proponowane zmiany korzystnie wpłyną na wywiązywanie się przedsiębiorców z obowiązków podatkowych, skutkować będą zmniejszeniem obciążeń małych firm, wyeliminują też wiele wątpliwości, które pojawiają się w stosowaniu przepisów podatkowych, i dostosowują obowiązujące regulacje do zmieniającej się rzeczywistości. W zakresie podatku dochodowego osób prawnych wskazać należy znaczne poszerzenie zastosowania preferencyjnej stawki podatku CIT. Dla tych podatników stawka wyniesie nie 19%, ale 9% podatku CIT. Skorzysta z tego 11 tys. podatników, a w ich kieszeniach zostanie ponad 400 mln zł. Jeszcze niedawno stawka CIT w Polsce wynosiła dla wszystkich firm 19%.

Pozytywną zmianą dla podatników CIT i PIT jest również przedłużenie zwolnienia z tzw. podatku minimalnego. Projekt zakłada, że zwolnienie stosowane będzie dalej, aż do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany. Ustawa przewiduje też zmiany dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt to uproszczony sposób rozliczenia podatku dochodowego. Podatnik nie oblicza dochodu, a zamiast tego stosuje obniżoną stawkę podatków wprost wobec osiągniętego przychodu, dzięki czemu unika żmudnych obliczeń, dokumentowania i ryzyka popełnienia błędu. Mniejsze firmy powinny jak najmniej czasu poświęcać na rozliczenie podatków, a jak najwięcej na dostosowanie swojego biznesu do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Postulują to od wielu lat m.in. rzecznik małych i średnich firm oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. My również podzielamy tę opinię. Stąd propozycje. Teraz limit podniesiemy aż ośmiokrotnie, do 2 mln euro. Po drugie, wyłączenia. Ustawa zawiera teraz listę aż 58 branż, które nie mogą korzystać z ryczałtu. Należą do nich np. usługi prawników, księgowych czy architektów. Usuniemy ogromną większość tych wyłączeń, pozostanie ich tylko kilka, wynikających ze względów bezpieczeństwa, np. prowadzenie kantorów czy handel częściami samochodowymi. Skorzystają osoby wykonujące wolne zawody, np. lekarze, tłumacze czy nauczyciele. W przyszłym roku chcemy pracować z rynkiem nad dalszym zmniejszaniem stawek ryczałtu, tak by korzystanie z niego było jeszcze bardziej atrakcyjne. W przyszłym roku dzięki tym zmianom z ryczałtu pierwszy raz w historii będzie mogło skorzystać aż 180 tys. firm. Dzięki temu w ich kieszeniach pozostanie prawie 900 mln zł. Wysoka Izbo! W czasie wychodzenia gospodarki ze spowolnienia kluczowe jest, aby firmom, szczególnie tym mniejszym, zapewnić równe warunki konkurencji z większymi podmiotami. To właśnie duzi rynkowi gracze mają największe możliwości oszczędzania na podatkach. Czasami dzieje się to przy użyciu nieuczciwych metod. Skutkiem jest ich jeszcze większa przewaga wobec mniejszego biznesu. Walka z unikaniem opodatkowania jest szczególnie pilna w czasach epidemii, ponieważ jest to czas, kiedy duże firmy wypychają z rynku mniejsze. Obniżki podatków dla małego biznesu i ostre kroki przeciwko unikaniu opodatkowania zapowiada teraz u siebie większość krajów Unii Europejskiej, w tym Niemcy, Francja, Austria, Włochy i Węgry. Polska już 4 lata temu wypowiedziała wojnę luce CIT-owskiej i rajom podatkowym. Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego dzięki uszczelnieniu podatków i reformie KAS luka CIT zmniejszyła się w ciągu 4 lat aż o połowę: z 2% do 1% PKB, ale wciąż wynosi ponad 22 mld zł rocznie, co oznacza, że do budżetu państwa nie trafia co trzecia złotówka, którą powinny zapłacić większe firmy. To duży koszt dla Polski, bo każda niezapłacona złotówka musi być rekompensowana przez uczciwego podatnika, najczęściej przez małych przedsiębiorców i pracowników. Chcemy wdrożyć sprawdzone w większości krajów Europy rozwiązania, które działają tam od wielu lat i są standardem cywilizowanych regulacji podatkowych. W sumie zmiany uszczelniające przyniosą ponad 2 mld zł i oznaczać będą zmniejszenie luki CIT z roku na rok o ponad 10%. To są środki, które pozostaną w Polsce (Dzwonek) i przyniosą korzyść polskiej gospodarce, szczególnie mniejszym firmom, w których jednocześnie obniżamy podatki.

W obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych, szczególną i istotną zmianą będzie wprowadzenie limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej. Od 2008 r. obowiązują przepisy, które preferencyjnie traktują dochody osób, które mieszkają w Polsce, ale przez część roku działają za granicą. W efekcie dochody uzyskiwane w wielu krajach są całkowicie zwolnione z opodatkowania w Polsce. Ulga abolicyjna często służy nieuczciwym firmom, żeby w ogóle nie płacić podatków w Polsce. Według informacji z kontroli podatku unika się np. poprzez transfer wypracowanego w Polsce zysku do zarejestrowanej w Holandii spółki. Zysk wypłacany jest potem z powrotem do jej polskiego właściciela, np. w formie wynagrodzenia dyrektora, które przez ulgę abolicyjną nie jest opodatkowane w Polsce. Brak podatków od dochodów z zagranicy staje się na świecie wyjątkiem. Polska zobowiązała się w ramach współpracy na polu OECD do zastąpienia go nowym globalnym standardem, czyli zaliczeniem podatku zapłaconego za granicą na poczet podatków do zapłaty w Polsce. Realizujemy nasze zobowiązania i zależy nam na tym, żeby w maksymalnym stopniu chronić osoby rzeczywiście pracujące przez część roku za granicą. Stąd przewidziana jest dla nich kwota wolna w wysokości 8 tys. zł rocznie. Podatek zapłacą jedynie osoby osiągające za granicą bardzo duże dochody. Według danych administracji osoby, których opodatkowanie się zwiększy, oszczędzają na podatkach do zapłaty w Polsce średnio aż 10 tys. zł rocznie. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie przedłożonego przez rząd projektu ustawy z druku nr 642. Projekt ustawy przewiduje zmiany w kilku ustawach podatkowych takich jak: ustawy o PIT, ustawa o CIT, ustawa o ryczałcie oraz ustawa o podatku tonażowym. Jednocześnie wprowadza zmiany w innych ustawach regulujących życie gospodarcze. Chodzi m.in. o ustawę o rachunkowości, Kodeks spółek handlowych, ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czy ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Głównym celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych zapewniające powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Tym samym przewiduje, że obejmie się zakresem podmiotowym ustawy o CIT mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP spółki komandytowe oraz te spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a w przypadku których podatnicy podatku dochodowego uczestniczący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się od opodatkowania. Proponowane regulacje nie obejmują spółek jawnych, w przypadku których tożsamość wspólników będących podatnikami podatku dochodowego, osób fizycznych lub prawnych, zostanie ujawniona organom skarbowym. W przypadku spółek komandytowych, których powiązania między wspólnikami nie wskazują na optymalizacyjny cel ich utworzenia, projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek, którego skutkiem efektywne opodatkowanie dochodów takich komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej pozostanie na porównywalnym poziomie do opodatkowania na podstawie aktualnych przepisów. Traktowanie spółek komandytowych jako podatnika podatku CIT jest rozwiązaniem powszechnie przyjętym w wielu krajach Unii Europejskiej i jest spójne z ogólnie przyjętą wewnątrzwspólnotową polityką podatkową. Kolejnym elementem uszczelniającym jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów akcji w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów. Na podstawie obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych trudno jest dochodzić należności od nierezydentów, dlatego w ramach uszczelnienia projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten dotyczy podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej niezależnie od osiąganych przez nią przychodów. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych proponowana jest zmiana dotycząca zwolnienia dla dochodów marynarzy pływających na statkach morskich, której celem jest zrównanie sytuacji prawno-podatkowej marynarzy będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego niezależnie od bandery, pod którą pływają. Zmiany w ustawie o ryczałcie polegają na podniesieniu limitu przychodów warunkujących wybór ryczałtu oraz limitu przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat ryczałtu, likwidacji większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym przez zmianę definicji wolnych zawodów, obniżenia i ujednolicenia niektórych stawek ryczałtu, doprecyzowania przepisów dla ryczałtu płaconego kwartalnie czy ułatwienia dla podatników na karcie podatkowej. Zakłada się, że zmiany spowodują poszerzenie grupy podatników mogących skorzystać z tej formy opodatkowania i zwiększą jej atrakcyjność. Proponowane są również zmiany w zakresie cen transferowych dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Polegają one na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej. Obejmują również rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych związanych z tymi transakcjami. Wprowadzone zmiany mają również na celu zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorstw (Dzwonek) w zakresie cen transferowych w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Michała Jarosa, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Omawiany projekt ustawy wpisuje się doskonale w charakterystykę postępowania rządu Mateusza Morawieckiego. Po pierwsze - traktuje przedsiębiorców i podatników jako potencjalnych oszustów. Po drugie - zaskakuje ich wprowadzanymi zmianami.

Wraz z rosnącym kryzysem zaufania do instytucji państwa większości obywateli i przedsiębiorców brakuje wiary, że cały system pracuje na ich korzyść. Lekką ręką sięgacie coraz głębiej do kieszeni przedsiębiorców i podatników, nakładając na nich coraz więcej danin, opłat, podatków, świadczeń, kontrybucji i obciążeń. Właśnie teraz, w czasie pandemii, podatnikom i przedsiębiorcom nie wolno przeszkadzać. Jeśli można, to trzeba im pomóc. Jak? Wyciągnijcie do nich rękę. Po prostu im zaufajcie. Zaufanie świadczy o poważnym państwie. W poważnym państwie nie wprowadza się zmian podatkowych od 1 stycznia, uchwalając je mniej niż 3 miesiące wcześniej, nie zaskakuje się zmianami podatników, księgowych, doradców podatkowych czy wreszcie sam fiskus. Głos ekspertów i strony społecznej, w tym przypadku przedsiębiorców, jest nie tylko słyszalny, ale przede wszystkim wysłuchany. W poważnym państwie systematycznie rośnie pozycja Polski w rankingach wolności gospodarczej.

To nie jest poważne państwo. Wiecie, co jest najgorsze? Że brniecie dalej. Dowodem na to jest ustawa, która wprowadza opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT, co bezpośrednio uderzy w polskie rodzinne przedsiębiorstwa, utrudniając im rywalizowanie z zagraniczną konkurencją.

To jest niezrozumiałe. Środowiska przedsiębiorców, środowiska pracodawców, zrzeszenia protestują przeciwko tej ustawie. Piszą do nas listy, wysyłają do nas informacje. Na sam koniec chcę państwu powiedzieć, że instytucja, którą powołaliście, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, też protestuje przeciwko tej ustawie.

Czego dotyczy ustawa? Panowie mówicie z taką łatwością o ludziach, którzy pracują za granicą, że są poza polskim systemem podatkowym. Przecież mówimy o ludziach, którzy często zostali wypchnięci do Wielkiej Brytanii, Anglii, Irlandii po to, żeby tam pracować. Resztę wysyłają do domu.

Dlaczego? Dlatego że wy sobie urządziliście bal, przez parę lat na wszystko was było stać, a dzisiaj okazało się, że pieniędzy nie ma, że pan Morawiecki już wszystkie je przejadł. Kto ma za to zapłacić? Mają zapłacić polscy emigranci, którzy pracują za granicą i co miesiąc wysyłają do Polski pieniądze, żeby utrzymać własne rodziny. To, co wy tutaj robicie, to jest wyjątkowa bezczelność. Okradacie ludzi, którzy w żaden sposób nie korzystają z państwa, tylko do tego państwa dokładają.

Będziemy robić wszystko, włącznie z obstrukcją parlamentarną w Senacie, żeby ta ustawa nie weszła w życie. To jest hańba, że żaden poważny człowiek - jakichś młodych ludzi tu przysyłają - nie jest w stanie uczciwie tutaj stanąć. Bardzo proszę, pani poseł Katarzyna Kretkowska, Lewica. Wysoka Izbo! Patriotyzm i wierność interesowi państwa polskiego można realizować na różne sposoby. W długiej historii naszych polskich dziejów Polki i Polacy walczyli zbrojnie w zrywach niepodległościowych, na wszystkich frontach wojennych świata, w ruchach oporu, w powstaniach, ale także dawali świadectwo swojego patriotyzmu w mozolnej odbudowie i umacnianiu polskiej gospodarki. Czynili tak zarówno w czasach niewoli, jak wielkopolscy pozytywiści w XIX w., jak i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. tymi patriotkami i patriotami odbudowującymi polską gospodarkę, jej konkurencyjność i konkurencyjność polskiego kapitału są właściciele polskich, rodzimych, często rodzinnych małych i średnich firm. To te małe i średnie firmy w największym stopniu budują dochód narodowy. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki znienacka postanowił wsadzić im nóż w plecy, konkretnie drugim najpopularniejszym w Polsce spółkom prawa handlowego, czyli spółkom komandytowym. Z dnia na dzień 70 tys. Polek i Polaków zatrudniających 3 mln pracowników i pracowniczek i generujących 300 mld przychodu dowiaduje się, że są oszustami, cytuję: agresywnymi optymalizatorami podatkowymi, funkcjonującymi tylko po to, by obejść prawo.

Rząd wpadł na pomysł, i to jest głównym założeniem tej ustawy, by te nasze spółki komandytowe podwójnie opodatkować, nie tylko podatkiem PIT, ale także CIT. Przypomina to jak żywo niechlubne „domiary” z czasów stalinowskich w Polsce, które ówczesna władza narzucała ledwo trzymającym się przy życiu resztkom prywatnych firm, by je ostatecznie dobić tym kolejnym podatkiem, oprócz podatku dochodowego i obrotowego. Uzasadnienie tego posunięcia w ustawie jest bałamutne i zmanipulowane. Odwrotnie do tego, co głosi rząd, ta zmiana wywoła głęboką asymetrię w opodatkowaniu polskich przedsiębiorców komandytowych w stosunku do ich zagranicznych odpowiedników oraz w stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których w Polsce jest sześć razy więcej niż komandytowych, z których to 72% w ogóle nie wykazuje dochodu, a więc nie płaci żadnego podatku, żadnego, a posiadają te spółki szereg przywilejów, których spółki komandytowe akurat nie posiadają. Bałamutne i cyniczne jest zapewnienie, że większość spółek komandytowych skorzysta z ulgi w podatku CIT, gdyż to te spółki, które nie załapią się na tę ulgę, wypracowują 90% przychodów wypracowywanych przez wszystkie spółki komandytowe w Polsce. I to te spółki będą teraz miały płacić 38% podatku, a ich zagraniczni konkurenci będą się tylko śmiać i zacierać ręce. Bałamutne jest również zapewnienie, że ta ustawa spowoduje, iż zagraniczne spółki komandytowe zaczną płacić w Polsce podatki, i tu rzuca się przykładami, np. Lidl.

Zresztą spółek komandytowych z jakimkolwiek udziałem zagranicznym jest mniej niż 2% wszystkich spółek komandytowych funkcjonujących na terytorium Polski. Ustawa ta wabi też zapowiedzią likwidacji ucieczek do rajów podatkowych, czego wszyscy byśmy sobie życzyli, sugerując, że także po to te spółki komandytowe powstały, ale tych spółek komandytowych, które są zarejestrowane czy na Cyprze, czy na Malcie, czy w Luksemburgu, jest w ogóle 0,4%.

Udział w podatku CIT gmin i powiatów jest sześciokrotnie niższy niż w PIT. Natomiast drugą sprawą, którą ta ustawa porusza, jest umożliwienie szerszej grupie podatników, konkretnie 175 tys. osób, korzystania z uproszczonej formy opodatkowania, czyli ryczałtu, a samorządy nie mają udziału w dochodach z ryczałtu.

Tu przed chwilą słyszeliśmy z ust przedstawiciela rządu, jakie to będzie fantastycznie korzystne. Natomiast ulga w krajach Unii Europejskiej jest pięciokrotnie wyższa, niż ulga w Polsce.

Ten projekt zaciska pętlę na szyi ledwo szamocących się z kryzysem, z lockdownem, z pandemią samorządów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Miejsce ustawy, która w dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego nakłada dodatkowe obowiązki podatkowe na polskich przedsiębiorców, jest, szanowni panowie ministrowie, w koszu. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska składam wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Jakie negatywne efekty przyjęcia tej ustawy się zmaterializują? Większość spółek komandytowych osiągających obroty powyżej 2 mln euro obudzi się w nowej rzeczywistości - podatku nie 19-, ale blisko 40-procentowego. Zdaniem przedstawicieli tych spółek to oznacza masowe bankructwa i przekształcanie się spółek w spółki jawne lub cywilne. Skokowy wzrost bezrobocia. Każda spółka komandytowa zatrudnia średnio co najmniej kilkudziesięciu pracowników, dlatego odrzucenie tego szkodliwego projektu ustawy jest wspólnym interesem pracodawców i pracowników. Zablokowanie inwestycji i nowych miejsc pracy. Czy o to w kryzysie, panowie ministrowie, chodzi? Liczne bankructwa polskich firm działających na niskiej marży. Zniechęcenie do wykazywania dochodów. Rozbudowanie szarej strefy. Znacząco obniży się zdolność konkurencyjna polskiego kapitału względem zagranicznych korporacji. Czy o to chodzi w dobie kryzysu?

Najpierw rząd przyznał pomoc, a teraz doprowadzi do tego, żeby ta pomoc była przez wiele upadających spółek komandytowych rządowi zwracana. Panowie Ministrowie! Co w praktyce dla tysięcy spółek komandytowych oznacza wejście w życie tej ustawy od 1 stycznia 2021 r. Po jej przyjęciu najpierw wspólnicy muszą mieć pewność, czy ten pomysł wejdzie w życie i w jakim kształcie. A o tym dowiedzą się dopiero, jak ustawa zostanie uchwalona. Czyli gdzieś w okolicach końcówki listopada. Następnie wspólnicy muszą siąść do stołu i przeprowadzić nierzadko długie negocjacje nad kształtem umowy nowej spółki, np. jawnej czy cywilnej. Następnie trzeba powołać nową spółkę, np. jawną, i są wszelkie z tym związane formalności. Krajowy Rejestr Sądowy musiałby ją zarejestrować, co w dużych miastach trwa nierzadko kilka miesięcy. Dopiero wówczas, już w nowym 2021 r., trzeba by przenieść cały majątek do nowej spółki, np. jawnej, zapłacić za pewne podatki z tym związane. Następnie trzeba podpisać nowe umowy z pracownikami.

Jest to niezwykle trudne, ponieważ nie wszyscy się na to zgodzą. Wielu będzie renegocjować warunki w części umów w ramach obecnej spółki komandytowej, są zakazy przenoszenia praw i obowiązków z obecnych umów na nowe podmioty. Ktoś o tym pomyślał w Ministerstwie Finansów? Jest to skrajnie nieodpowiedzialny skok na polskie firmy. I to jest brutalnie agresywne słowo, bo takim jedynie można to nazwać. Jest jeszcze czas, aby - tak jak powiedziałem na wstępie - w dobie rozkręcającego się kryzysu roztoczyć nad tą sprawą pewną refleksję, przemyśleć to, naprawdę wycofać się z tego projektu, bezwzględnie tragicznego dla spółek komandytowych. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Ze względu na szacunek dla polskich przedsiębiorców i polskich wyborców chcę poruszyć temat planów podwójnego opodatkowania spółek komandytowych. Puste ławy sejmowe pokazują szacunek dla polskich przedsiębiorców, jaki ma partia rządząca. Pokazują, jak wygląda rzeczywisty stosunek polityków opcji rządzącej, nie ten deklarowany w mediach, ale rzeczywisty, do kilkudziesięciu tysięcy polskich spółek komandytowych, do polskiego kapitału z branży transportowej, z branży budowlanej, z branży motoryzacyjnej, z branży przetwórstwa szkła i wielu, wielu innych, do ludzi, którzy prowadzą legalną dochodową działalność gospodarczą, efektywnie konkurując na rynkach europejskich, i teraz mają być zniszczeni w wyniku kaprysu rządu. Czy chodzi o to, że rozdaliście pieniądze z tarczy finansowej do spółek, brakuje wam w budżecie i to, co jedną ręką rozdajecie w ramach tarczy, teraz chcecie odzyskać? Czy chodzi o obejście regulacji konstytucyjnych, o to, że nie możecie wprost sfinansować długu rządowego? Jeżeli nie, to wytłumaczcie, jaka logika stoi za tym, że ta forma prowadzenia działalności gospodarczej przez 5 lat nie budziła waszych zastrzeżeń, a teraz nagle jej opodatkowanie ma wzrosnąć nie o 1 punkt procentowy, nie o 2, ale o kilkanaście? Prawie dwa razy. Jaki to ma sens? Po co chcecie to zrobić? Jak polscy przedsiębiorcy mają konkurować na rynkach międzynarodowych? Czy naprawdę chcecie te nowe przepisy wprowadzić od stycznia? Żadnych konsultacji? No jak można tak zrobić? Jak wam nie wstyd w ogóle? Jak nie wstyd wam wobec przedsiębiorców, którzy ciężko pracują? Setki tysięcy Polaków pracują w tym schemacie. Podobno pracujecie nad jakimiś programami mieszkaniowymi. Czy wiecie, że ponad połowa mieszkań w Polsce jest budowana przez spółki komandytowe, w które w tej chwili chcecie uderzyć? Jak w ogóle mogliście wpaść na taki pomysł? Jak mogliście nie zaprosić nikogo do żadnych konsultacji? Konfederacja nigdy nie zgodzi się na taki gangsterski standard uprawiania polityki, w jakim uczestniczą. Ubolewam nad tym, że widzę tutaj urzędników, nie widzę polityków, ubolewam, że musicie panowie firmować swoimi twarzami i swoimi nazwiskami, siedząc w ławach rządowych, tę haniebną politykę, której twarzy nie mają tutaj odwagi dać Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński ani inni politycy, którzy bawią się we władców marionetek, w panów życia i śmierci, w panów praw obywatelskich, w panów wolności gospodarczej, którą niszczą w Polsce.

Zwracam panu posłowi uwagę, że dzisiaj na sali obowiązuje nakaz zakładania maseczek i pan świadomie nie wykonuje zalecenia Prezydium Sejmu, biorąc odpowiedzialność za zdrowie pracowników Sejmu i posłów. Spokojnie, porozmawiamy o maseczkach po tym, jak 41 tys. spółek komandytowych zostanie rozwiązanych, bo do tego prowadzi ta ustawa. Czy panowie naprawdę sądzą, że podwójne opodatkowanie nic nie zmieni w tych spółkach, że oni śpią na pieniądzach, że - nie wiem - mają dorobione te pieniądze, mają maszynki do wyrabiania tych pieniędzy i po prostu sobie dodrukują? Ja też przez wiele lat prowadziłem spółkę komandytową i to nie jest tak, że zarabia się tam jakieś kokosy bez pracy i po prostu czeka się, na co je wydać. Nie wiem, czy pan pracował kiedyś na wolnym rynku, kiedy określa pan te spółki komandytowe jako coś, gdzie - nie wiem - pieniądze się wyprowadza czy nie płaci się podatków.

Jak pan sobie wyobraża jakiekolwiek biznesplany, jakiekolwiek kredyty? Jak państwo to sobie wyobrażają? Mają teraz renegocjować te kontrakty, powiedzieć swoim kontrahentom: wiecie, sorry, w Polsce zmienił się system podatkowy? Serio? Tak to ma wyglądać? Przecież ci ludzie wcześniej czy później po prostu wyprowadzą swoje firmy za granicę. Tam, powiedzą sobie, można te nasze firmy prowadzić, a tutaj się nie da. wobec 41 tys. spółek komandytowych, gdzie 95% to jest polski kapitał? A więc od kogo ściągacie? Od polskich przedsiębiorców. I do tego doprowadza nasz rząd. Czemu ma to służyć? Przecież tak się nie negocjuje. Nie da się tak prowadzić swojej spółki, jeśli wszystkie finanse są jawne. Dziękuję, panie pośle. Jeżeli nie, zamykam listę.

Chciałbym zapytać panów ministrów, czy mają świadomość, że Polacy, którzy uzyskują dochody za granicą, po prostu pracują za granicą, utrzymują swoje rodziny, pracując np. w Irlandii czy Wielkiej Brytanii, mogą wystąpić o tzw. rezydenturę podatkową w Wielkiej Brytanii. Pan mówi, że mogą? Ten prawie że nacjonalistyczny rząd spowoduje, że ich więź z Polską tak naprawdę zniknie. Oni zostaną straceni dla Polski, dla polskiego budżetu.

Chciałem zapytać, czy ta ustawa dotknie również polskich urzędników pracujących w instytucjach europejskich.

Wysoka Izbo! Podatki powinny być sprawiedliwe i proste. Jesteś pracownikiem - płacisz podatki, prowadzisz działalność gospodarczą - płacisz podatki, do tego odpowiadasz własnym majątkiem, jesteś udziałowcem w firmie - brawo ty, odpowiadasz jedynie do wysokości swoich udziałów, za ten przywilej obowiązuje cię podatek CIT, coś za coś, żeby reguły gry były sprawiedliwe dla wszystkich. Niestety spółki komandytowe to jest wyrwa w tych regułach, wyrwa kosztowna dla budżetu. W spółce komandytowej można jednocześnie nie płacić podatku CIT i nie odpowiadać za firmę majątkiem. A jak się dobrze zakręcić i zarejestrować spółkę matkę na Karaibach, to w ogóle nie płacisz podatku. To nie jest fair wobec pracowników ani wobec innych przedsiębiorców. Dziwi mnie stanowisko PSL-u, który broni spółki komandytowej jak niepodległości. Jak ten przywilej wprowadzono, to wasza posłanka wtedy pomstowała na to i mówiła, że to jest najprostsza droga do wyprowadzenia nieopodatkowanych zysków. Ustawa oczywiście doskonała nie jest, są też kiksy.

Bardzo proszę, pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani marszałek, jak również ja jesteśmy posłami okręgu warszawskiego, który obejmuje Polaków i Polki żyjących za granicą. Ta właśnie ustawa dotyczy tych osób, które zarabiają za granicą. Co jest w tej ustawie, Wysoka Izbo? Przede wszystkim jest to likwidacja ulgi abolicyjnej. Oznacza to, że niektórzy Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższe podatki. Ulga abolicyjna polega na umorzeniu określonej części bądź całości podatku w określonych sytuacjach. Obecnie najczęściej stosowana jest w kontekście rozliczania podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą. Mamy panią Annę, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam też płaci podatek dochodowy. W całości uzyskuje swoje dochody w Wielkiej Brytanii. Dlaczego dochodami Polek i Polaków pracujących za granicą chcecie łatać tę dziurę budżetową, ten deficyt, który tylko w tym roku wynosi już 110 mld zł? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Nie można karać tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą. Nie można karać tych, którzy pracują po 10, 12 godzin na dobę. Nie można karać tych, którzy tworzą miejsca pracy. Nie można karać tych, którzy ponoszą ryzyko. Naszym obowiązkiem jest wspieranie polskich przedsiębiorców. Ustawa, którą panowie proponujecie, ogranicza wsparcie dla polskich przedsiębiorców na rzecz przedsiębiorców z zagranicy. Nie można się na to zgodzić. Ostatnia rzecz - czas. Czy rząd PiS-u nie widzi, co się dzieje w Polsce? Nie widzi, że bardzo duża grupa spółek, bardzo duża grupa przedsiębiorców jest na pograniczu bankructwa, każdego dnia walczy o przetrwanie, walczy o swoich pracowników?

Bardzo proszę, pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Przepraszam, ale parują mi okulary. Chciałoby się przytoczyć klasyka, i to klasyka z tej strony sali, który kiedyś powiedział: wysłać tych ekonomistów na Saharę, to za miesiąc piasku zabraknie. Czy w ogóle ktokolwiek liczył, kiedy próbujecie wprowadzić ten projekt. Proszę państwa, spółki komandytowe w waszym projekcie zostały zrównane ze spółkami z o.o. Firmy, osoby fizyczne, które do tej pory nie płaciły dwóch podatków PIT i dywidendy, jeśli postanowiły wyodrębnić swoje działania związane z działalnością gospodarczą od majątku osobistego - bo o to chodziło, żeby wyodrębnić majątek działalności gospodarczej od osobistego - po zmianach dostaną dodatkowy podatek CIT.

Nie jest kosztem, panowie. Bardzo proszę, pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Po raz drugi w przeciągu godziny ograbiamy polskie samorządy.

Powiedział m.in., cytuję: mam nadzieję, że prace zakończą się jak najszybciej i wprowadzimy tę możliwość już od przyszłego roku podatkowego, czyli od rocznego rozliczenia za rok 2020. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo!

Konsultacje społeczne tak ważnego projektu w waszym wykonaniu to kpina i bezprawie, tak samo jak kpiną i bezprawiem jest danie przedsiębiorcom 3 miesięcy na dostosowanie się do tak istotnej zmiany.

Za co chcecie karać przedsiębiorców, sięgając brutalnie do ich kieszeni po pieniądze?

Rozdawnictwo rządu doprowadziło do tego, że gwałtownie szukacie pieniędzy w kieszeni podatników. Dlaczego robicie to kosztem przedsiębiorców i samorządów? Pan poseł Marek Rutka, klub Lewica. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Zgodnie z przygotowanymi propozycjami legislacyjnymi likwidacja obecnie przysługującej ulgi abolicyjnej będzie przejawem dyskryminacji przede wszystkim polskich marynarzy. Mówię to jako poseł ziemi pomorskiej. Powyższe działania rządu wskazują, iż polscy marynarze są traktowani wyłącznie jako obciążenie dla kraju. Należy wskazać, że to właśnie marynarze bardzo dotkliwie odczuli skutki światowego kryzysu spowodowanego pandemią. Warty podkreślenia jest fakt, iż marynarze nie posiadają uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego, a także z racji wykonywanego zawodu nie nabywają prawa do emerytury.

Likwidacja obecnie przysługującej ulgi abolicyjnej będzie przejawem dyskryminacji przede wszystkim cenionych w świecie (Dzwonek) polskich marynarzy. Skąd takie podejście? Czym marynarze podpadli dobrej zmianie? Tym, że nie pływają na statkach pod polską banderą? Zbudujcie obiecane promy i zarejestrujcie je w kraju, wówczas dacie im na to szansę. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze!

A zatem, szanowni państwo, Polacy, trzymajcie się za kieszenie. W spółkach komandytowych średnio - przy proteście - 15% dodatkowego podatku, tak skromnie. W tym roku już państwo podwyższyli VAT, o 8 mld zł, dla każdego.

Państwo zatrzasnęli drzwi przed Polakami pracującymi za granicą. Na nic słowa: wracajcie, tu jest rynek pracy, dzisiaj mamy bardzo trudną sytuację. Państwo nie szanujecie Polaków, którzy zarabiają pieniądze za granicą. Nie robicie żadnego kroku, aby można [[Dzwonek]] było im pomóc. To jest po prostu skandaliczne. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Kopiec, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nieobecni w pracy posłowie PiS i nieobecni w pracy ministrowie PiS! Kolejny raz chcecie mordować polski biznes, bo go nie rozumiecie, bo od lat zajmujecie się wyłącznie wydawaniem nie swoich pieniędzy. Po co wam te większe podatki? Na propagandę telewizji Kurskiego? Tam już poszło 8 mld zł. Na kolejne niepoliczalne stanowiska dla waszych rodzin w spółkach Skarbu Państwa? Na kupowanie koalicjantów? Na dopłaty do podwójnych fuch posłów wiceministrów, tych co wierniejszych? Na co? Opamiętajcie się, bo nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to grzech ciężki, a niegospodarność to zbrodnia przeciwko ciężko pracującym na wasze wyżywienie ludziom. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Przed kilkoma minutami powiedział pan z rozbrajającą szczerością, że musimy wspólnie ponieść tę odpowiedzialność za CIT estoński. Teraz mówicie państwo o tym, że pewnie wspólnie musimy ponieść kolejne ofiary. Argumenty nie mają dla państwa żadnego znaczenia - czy to będzie obniżka pensji, czy to będą bankructwa. Szanowni Państwo! Zostawcie tę gospodarkę w spokoju, nie psujcie jej. Nie psujcie jej, szanowni państwo, bo niczego dobrego z tego nie będzie. Zostawcie te spółki komandytowe. Podpisaliście się razem, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie zwierząt, a dzisiaj tworzycie nową koalicję. Polska Zjednoczona Prawica plus nowa Lewica. Szanowni państwo, współczuję.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej spotkaliśmy się wspólnie z przedsiębiorcami, którzy bazują właśnie na tej formie działalności, na spółce komandytowej. Czy rząd PiS-u zdaje sobie sprawę, że tą ustawą zarzyna kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzinnych firm, które bazują właśnie na tej formie działalności gospodarczej? Na spotkaniu byli przedstawiciele i transportu, i wyrobów szklanych, i prawników. Wszyscy podnoszą larum, wszystkim się wasza ustawa nie podoba. Jakie wy znajdujecie argumenty, żeby dzisiaj nas przekonać do poparcia tej ustawy?

dzisiaj - nowy podatek dla spółek komandytowych.

Bardzo dziękuję, panie pośle.

PiS dzisiaj atakuje polskie rolnictwo, polski przemysł mięsny, polski przemysł drobiarski.

Ta ustawa wprowadza podwójne opodatkowanie dochodów od spółek komandytowych. Ustawa jest tak absurdalna, że będzie promowała podmioty zagraniczne w Polsce, które nie będą opodatkowane podwójnie, natomiast będą opodatkowane podwójnie polskie podmioty gospodarcze. Mamy umowę zakazującą podwójnego opodatkowania między Polską i Niemcami. Czy te podmioty mają się przenieść do Niemiec? Wiadomo, iż ta ustawa spowoduje tylko jeden efekt, [[Dzwonek]] likwidację 40 tys. polskich podmiotów, rodzinnych firm, które z trudem budowały swój kapitał i polską gospodarkę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, klub Lewica. Pani Marszałkini! Ja mówiłam w imieniu klubu Lewica, że jesteśmy negatywnie nastawieni do tej ustawy, i dość szczegółowo tłumaczyłam dlaczego.

Chciałam zapytać, czy rząd posłucha Ministerstwa Rozwoju, które negatywnie zaopiniowało ten projekt, czy nie.

Chciałam zapytać po drugie i po trzecie: Dlaczego rząd nie słucha opinii osób, z którymi się konsultuje, i dlaczego konsultacje w tak ważnej sprawie były 2-dniowe? To jest kpina. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Debatujemy o podatkach i ich wpływie na działalność gospodarczą poszczególnych przedsiębiorców, ale jednocześnie warto i należy zapytać o skutki finansowe tych zmian.

W całym materiale nie znalazłam żadnej informacji, jak rząd zamierza zrekompensować te ubytki samorządom. Nie ma na ten temat żadnej informacji, a przecież regularnie samorządom dokłada się zadań i zabiera się pieniądze. Dlaczego? Dziękuję bardzo. Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To jest ustawa o grabieniu polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, fakty. To jest fundament naszej gospodarki. Skoro pracujecie ciężko, skoro zarabiacie, to my wam jeszcze dołożymy.

Po drugie: Czy ktoś z was w ministerstwie sprawdził, czy ta ustawa nie doprowadzi do skokowego wzrostu bezrobocia, zablokowania inwestycji, obniżenia pensji pracownikom? Bardzo proszę, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jesteście zwyczajnymi kłamcami. 1 lipca premier Morawiecki powiedział, że prezydent Duda jest gwarantem niepodnoszenia podatków w Polsce. 8 lipca prezydent Andrzej Duda w czasie kampanii powiedział, że zawsze będzie zmierzał do tego, by obniżać podatki. Kilka miesięcy minęło, okłamaliście Polaków i nie macie jeszcze honoru, aby stanąć przed nimi - bo ani jednego posła Prawa i Sprawiedliwości nie ma - aby spojrzeć Polakom w oczy i powiedzieć: tak, podnosimy wam podatki. 2,5 mln Polaków pracujących za granicą będzie musiało zapłacić dodatkowy podatek w Polsce kosztem swoich rodzin. 72 tys. polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniają 3 mln pracowników, nie będzie już tak dobrze konkurować z zagranicznymi koncernami, dlatego że zagraniczne koncerny mają [[Dzwonek]] zaledwie 1% rynku w spółkach komandytowych. Bardzo proszę, pani poseł Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W wystąpieniu pana podsekretarza nieustannie powielało się słowo „nieuczciwi” Ale chcę panu przypomnieć, że przedsiębiorcy chcą płacić w Polsce podatki proste i uczciwe, i sprawiedliwe. Może pan nie wie, ale większość obecnych spółek komandytowych to są polskie podmioty. Bardzo dużo z nich wyrosło na tyle, że skutecznie walczą o miejsce na naszym rynku z podmiotami zagranicznymi. Opodatkowanie spółek komandytowych posłuży tylko i wyłącznie pokryciu dziury budżetowej, którą kryształowi przedstawiciele rządu po prostu wygenerowali.

Budżety firm są już zaplanowane i te zmiany są dla nich zbyt nagłe, zbyt trudne do przeprowadzenia. To spowoduje u nich ogromny kryzys. Spółka komandytowa jest spółką na trudne czasy. Takie trudne czasy mamy teraz. Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Sytuacja firm w dobie pandemii jest naprawdę bardzo trudna. W firmach spadają przychody, spadają zyski, natomiast rosną wydatki. Wiele firm musi zwalniać pracowników, część z nich bankrutuje.

W uzasadnieniu piszecie o agresywnej optymalizacji podatkowej. Samo sformułowanie jest krzywdzące, ponieważ te firmy działają na podstawie polskiego prawa. To tak, jakby karać wszystkich kierowców za to, że jeden przekroczył prędkość. Piszecie również, że chodzi o kapitał zagraniczny, tymczasem zaledwie 3% z tych firm posiada ten kapitał zagraniczny.

Organizacja przedsiębiorców alarmuje, że to nie przyczyni się do wzrostów budżetowych, a jedynie spowoduje falę upadków spółek komandytowych, przekształceń i przejść w szarą strefę. Jaki naprawdę cel stoi za waszym działaniem? Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Ta faktyczna likwidacja, Wysoka Izbo, spółek komandytowych to absolutnie haniebny pomysł. Premier Morawiecki, który klęcząc na kolanach przed zagranicznymi korporacjami obiecał im, że nie będzie ich opodatkowywał, teraz w sposób absolutnie bezczelny sięga do kieszeni polskich małych firm rodzinnych, bo to o te polskie małe firmy rodzinne chodzi. To nie są wielkie zagraniczne korporacje, które nie płacą podatków, choć oni chcą nam to wszystkim wmówić. 97% spółek komandytowych to polskie firmy, małe firmy rodzinne. Co więcej, one wybierały to opodatkowanie, żeby płacić podatki, tylko płacić w sposób obiektywnie prostszy. Natomiast dziś, kiedy rząd mówi, że nie może opodatkować tych zagranicznych firm, sięga właśnie do kieszeni tych polskich małych firm. Tego projektu, szanowni państwo, nie da się naprawić. Mam nadzieję, że rząd przyjdzie po rozum do głowy i wycofa się z tego haniebnego projektu.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To skandaliczna ustawa, która powinna być natychmiast wycofana z procedowania w Sejmie. A tu mamy polskie rozwiązanie, z którego korzysta właśnie tyle firm, ile pan planuje przerzucić na ten estoński CIT. Zarzynacie po prostu firmy, które działają legalnie, płacą legalnie podatki w ramach systemu, który jest zbudowany w Polsce. Właśnie to rozwiązanie może być tym polskim estońskim CIT-em, jeżeli tyle firm wybiera taki sposób opodatkowania. Zastanówcie się, bo dobrobyt i dochody państwa biorą się z pracy. Wam to przeszkadza. Drukujecie pieniądze na potęgę i myślicie, że będziecie wiecznie ściągać z przedsiębiorców kasę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Michał Jaros, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! PiS chce dzisiaj tym projektem po cichu, skrycie ukarać 40 tys. polskich przedsiębiorców. Skandal! ...i do tego wyszarpać z ich kieszeni kolejne pieniądze, żeby załatać dziurę budżetową. Władza PiS-u wiele mówi o Polsce, o polskich firmach, o wsparciu dla Polski. Właśnie widzimy, jakie jest wsparcie dla polskich firm. Co robicie dla tych polskich firm? Panie Ministrze! Chciałbym zapytać, ile z tych 40 tys. polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w Polsce ma polski kapitał, a ile zagraniczny. Chciałbym zapytać też, bo mówicie o tym, że są dobre zmiany, że pojawia się niższy podatek CIT, ile firm skorzysta z tego niższego podatku CIT. Ten projekt jest zły, ten projekt jest skandaliczny. Skandaliczne było procedowanie nad tym projektem. Będziemy przeciwni temu projektowi i nie pozostawimy tego tak, że to będzie po cichu załatwione w Sejmie. Nawet jeśli nikogo z PiS-u na tej sali nie ma, będziemy głośno krzyczeli. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze!

Boją się, że dorobek ich życia pójdzie z dymem, bo kolejny przestój w generowaniu przychodów będzie po prostu oznaczał ich upadłość. Tak samo obywatele mają nawrót lęku dotyczącego utraty pracy, zarówno ci mieszkający w kraju, jak i ci poza naszymi granicami. Wyjechali, bo nie mogli tutaj znaleźć dobrej, godnej pracy. Opodatkowuje zarówno jedną, jak i drugą grupę. Jesteście naprawdę wyjątkowi na mapie świata i mapie Europy. Podczas gdy w innych krajach ułatwia się życie ludziom, przedsiębiorcom, zmniejsza się opodatkowanie, wy pracujecie na dwa podstawowe symbole (Dzwonek), symbole rządu PiS: po pierwsze, lawinowy wzrost zadłużenia kraju, po drugie, lawinowy wzrost liczby podatków będących w krajowym systemie podatkowym. Nie macie prawa mówić kiedykolwiek, że obniżacie Polakom podatki, bo wy je. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj przedstawiciele spółek komandytowych, którzy gościli w klubie Koalicji Polskiej, przedstawili dane pokazujące, że ponad 99% spółek komandytowych to są działalności gospodarcze kapitałowo związane z naszą gospodarką. Państwo staracie się przeczyć, dowodząc tego, że spółki komandytowe to jest jakiś obcy kapitał, to są jacyś spekulanci. To jest nieprawda. Chociaż widzę, że jesteście skuteczni, bo nawet niektórzy przedstawiciele Lewicy, jak pan poseł Konieczny, się na to łapią.

Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Jana Sarnowskiego o udzielenie odpowiedzi.

Rozpoczynając odpowiedź od kwestii ulgi abolicyjnej, chciałbym szanownym państwu posłom również przypomnieć, że ulga abolicyjna dotyczy polskich rezydentów podatkowych, tzn. osób, które mieszkają w Polsce ponad 183 dni, czyli ponad pół roku.

Szanowni państwo, nowa zasada rozliczenia, zasada, którą promuje OECD, do której wdrożenia zobowiązała się Polska, funkcjonuje w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej. Przyjęły ją również u siebie Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Austria, Litwa, Słowacja. To są kraje, w których ona już działa, i to są również te kraje, w których pracujący Polak, konkurując z mieszkańcami innych również tam działających państw, opodatkowany będzie na podobnej zasadzie, tzn. na zasadzie zaliczenia podatku zapłaconego od pracy na miejscu na poczet podatku do zapłaty w miejscu jego stałego zamieszkania, tam gdzie mieszka więcej niż pół roku - w wypadku ulgi abolicyjnej w Polsce. Co do marynarzy, szanowni państwo, w toku prac rządowych wprowadzona została do regulacji zmiana przewidująca zwolnienie niektórych grup zawodowych ze zmian w zakresie ulgi abolicyjnej. Przede wszystkim chodzi o tych, którzy nie wykonują swojej działalności na terytorium lądowym państwa, w którym pracują. Stąd marynarze nie będą objęci zmianami w uldze abolicyjnej. Co do gospodarki w czasie pandemii, szanowni państwo, to, czego potrzebują teraz firmy, to są trzy rzeczy. Po pierwsze, niskie opodatkowanie - niskie opodatkowanie, które, po pierwsze, da firmom poduszkę bezpieczeństwa, po drugie, zapewni im środki na inwestycje. Po drugie, jest to prostota rozliczeń - prostota rozliczeń, którą zapewni w przyszłym roku powszechny dostęp do ryczałtu oraz estoński CIT dla firm, które się rozwijają.

Pewne zmiany dotkną 40 tys., czyli dziesięciokrotnie mniej, przy czym nie zawsze będą to zmiany na minus. Zmiany uszczelniające łącznie z opodatkowaniem spółek komandytowych przyniosą do budżetu 2 mld zł.

Skąd wzięły się zmiany dotyczące spółek komandytowych? Według danych z kontroli prowadzonych przez administrację skarbową zarejestrowane w Polsce spółki komandytowe coraz częściej stanowią wehikuł służący wyprowadzaniu środków do rajów podatkowych, dokonują tego poprzez transakcje z zarejestrowanymi tam powiązanymi ze sobą podmiotami. Dotyczy to zarówno tych firm, których właścicielami są podmioty zarejestrowane w rajach podatkowych, których rzeczywiście jest bardzo niewiele, jak i tych, których właścicielami są Polacy - Polacy, którzy są jednocześnie udziałowcami lub pełnią funkcje menedżerskie w podmiotach zarejestrowanych w Holandii, na Cyprze czy w Luksemburgu. Według danych pochodzących z badanych przez Krajową Administrację Skarbową MDR-ów coraz częstsza jest praktyka polegająca na działaniu w formie hybrydy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej. W takim schemacie spółka komandytowa kamufluje jedynie rzeczywistą działalność przedsiębiorcy, która gospodarczo, ekonomicznie nie różni się od sytuacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to to samo zjawisko, które 6 lat temu było przyczyną objęcia CIT-em spółki komandytowo-akcyjnej. W roku 2014 tutaj również w Sejmie padały argumenty takie, że objęcie spółek komandytowych CIT-em to jest kwestia elementarnej sprawiedliwości podatkowej, to jest kwestia równości wobec prawa, kwestii konstytucyjnych. I padało to z ust ówczesnych ministrów finansów, którzy prezentowali ten projekt. Nie udało się tego zrealizować tylko dlatego, że podówczas spółki komandytowe nie były powszechnie używane w formule hybrydowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością do unikania opodatkowania. Ten problem, który zauważa Polska, pojawia się w wielu krajach, które starają się z nim walczyć. Popiera to OECD, które rekomenduje objęcie spółek osobowych CIT-em, zrobiło to już 12 państw Unii Europejskiej, zarówno na Zachodzie - Belgia i Hiszpania, jak i w naszym regionie - Litwa, Czechy, Węgry, Bułgaria i Rumunia. Oczywiście nie. Będą dalej służyć biznesowi do pozyskiwania kapitału. Mniejsze firmy zmiany nie odczują. CIT zapłacony przez spółkę będzie odliczany od podatku płaconego przez wspólników. Sytuacja komplementariusza się nie zmieni, odliczy podatek spółki od swojego, a komandytariusz otrzyma kwotę wolną. Dodatkowo dzięki prawie dziesięciokrotnemu zwiększeniu, dwukrotnemu, przepraszam, zwiększeniu limitu zastosowania preferencyjnej stawki 9%

Nie jest prawdą, że zagraniczne spółki działające w Polsce będą miały w efekcie tego lepszą pozycję konkurencyjną niż spółki polskie.

Szanowni Państwo! Mówią państwo czasami o przykładzie Niemiec. Ale pamiętajmy, że tam nie ma liniowej stawki 19% i to opodatkowanie na poziomie wspólnika sięga tam nawet 45%, bo tak ustalona jest w Niemczech progresja podatkowa.

Dziękuję. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu, proponuje. Przepraszam. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań.

Proszę ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej pana Tadeusza Kościńskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu.

Marszałek! Wysoka Izbo!

Gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów wymusiło aktualizację parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz uruchomienie nadzwyczajnych narzędzi do walki ze skutkami pandemii. Kluczowe parametry zawarte w ustawie budżetowej są pochodną aktualnej sytuacji makroekonomicznej oraz naszych oczekiwań i prognoz w zakresie jej rozwoju w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Przedstawię pokrótce Wysokiej Izbie najważniejsze informacje dotyczące projektu budżetu państwa na rok 2021. Sytuacja makroekonomiczna. Przyjęte przez nas założenia makroekonomiczne są dość konserwatywne. Zakładamy, że produkt krajowy brutto wzrośnie w przyszłym roku o 4%, co jest wynikiem zbliżonym do prognoz Narodowego Banku Polskiego, Komisji Europejskiej i co mieści się w przedziałach prognoz rynkowych. Jest to poziom podobny do poziomów osiąganych w ostatnich latach. W zakresie podstawowych wskaźników rynku pracy przewidujemy, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się na koniec bieżącego roku do 8%, a na koniec roku przyszłego spadnie do 7,5%. Przyjęliśmy, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5% w bieżącym roku oraz 3,4% w przyszłym roku. Jednocześnie zakładamy średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w tym roku, i o 1,8% w roku przyszłym. Przyjmujemy, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany wskaźnika inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP, to jest 2,5%. Wysokość dochodów budżetu państwa w przyszłym roku będzie determinowana przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Na stronę dochodową wpływ będą miały kontynuowane oraz nowe działania wspierające odbudowę wzrostu gospodarczego.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków budżetu państwa na rok 2021 wynosi 486,7 mld zł i jest niższy od planowanego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na bieżący rok o ponad 21 mld, tj. 4,2%. W kwocie tej zabezpieczono środki na kontynuację priorytetowych działań uwzględniających m.in. zwiększanie nakładów na zdrowie, naukę i obronę narodową. W budżecie na przyszły rok nastąpi powrót do stosowania limitów wyznaczonych stabilizującą regułą wydatkową, choć w zmienionej formie. Zgodnie z klauzulą uwzględniono połowę prognozowanej sumy skutków finansowych działań bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w bieżącym roku. Deficyt budżetu państwa wyniesie 82,3 mld zł. Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych liczony według metodyki unijnej prognozowany jest na poziomie ok. 6% PKB.

Wzrost zadłużenia wynika przede wszystkim z wydatków związanych z tarczą antykryzysową i tarczą finansową, czyli wydatków na ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy. Wysoki Sejmie!

Kontynuujemy politykę budżetową opartą na wspieraniu ożywienia gospodarczego i powrotu na ścieżkę wzrostu przy zachowaniu bezpieczeństwa finansów publicznych. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Dziękuję, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 15-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Pierwszy pan poseł Henryk Kowalczyk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

W 2020 r. notujemy spadek PKB w rozwiniętych krajach o ok. 10%, a w dużych krajach Unii Europejskiej, takich jak Włochy, Hiszpania czy Francja, ten spadek jest szacowany na 13%.

Wiem, że mogą się nie podobać, bo rzeczywiście Polska radzi sobie znakomicie na tle innych krajów w tej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej spowodowanej skutkami pandemii. Oczywiście jest tak, że przy konstrukcji budżetu na 2021 r. naprawdę trudno jest przewidzieć realne zdarzenia gospodarcze, jak dalej będzie rozwijać się pandemia. Jak to dalej będzie wyglądało? Jak długo potrwa?

Czy unikniemy kolejnego lockdownu? Bo to też jest niebezpieczeństwo.

Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę te wszelkie niepewności, skonstruowało budżet na 2021 r. w sposób niezwykle odpowiedzialny, powiedziałbym, chociaż było to zadanie bardzo trudne. Przyjęte w projekcie założenia makroekonomiczne eksperci określają jako rozsądne, rozsądne w tych warunkach, oparte na przewidywaniach takich, że po umiarkowanej recesji w 2020 r. w 2021 r. powróci wzrost gospodarczy - oczywiście wzrost gospodarczy porównywalny z rokiem 2020, a więc to nie jest nawet wzrost gospodarczy porównywalny do roku 2019, ale ten projekt w stosunku do roku 2020 przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 4% PKB. Te założenia, można by powiedzieć, są optymistyczne, ale też bardzo realne. Podobnie przewiduje się, że wzrośnie bezrobocie, ale w sposób bardzo umiarkowany, do poziomu 7,5%.

Myślę, że wpływ na poziom bezrobocia, na zatrudnienie, a tym sposobem i na finanse budżetowe - bo to nie tylko budżet, ale również składki w innych funduszach - powoduje, że.

Biorąc pod uwagę te prognozy wzrostu PKB i bezrobocia, szacowane dochody są planowane na takim realnym poziomie jak w 2020 r., więc niewątpliwie jest to prognoza bardzo ostrożna, ale taka ostrożna prognoza daje większą pewność zrealizowania jej bez korekty w czasie trwania roku budżetowego. Bo oczywiście korekta, która dotknęła budżet roku 2020, była naturalnym zjawiskiem i efektem pandemii, której nie dało się przewidzieć, nikt nie przewidywał tej pandemii w momencie, kiedy budżet na 2020 r. był uchwalany. Wydatki budżetu mają być realnie niższe od wydatków w roku 2020, czyli według tego znowelizowanego budżetu, ale też mają być wyższe w stosunku do roku 2019. To zwiększenie wydatków budżetu w stosunku do 2019 r. pokazuje, że to jest ta aktywność państwa w walce ze skutkami kryzysu.

Oczywiście jest to deficyt nieporównywalny z latami przed rokiem 2019 czy poprzednimi, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość sprawowało rządy, ale można powiedzieć, patrząc optymistycznie na porównanie, że on jest jednak mniejszy w stosunku do tego, który jest planowany w roku 2020 już po nowelizacji budżetu.

Co ważniejsze, relacja długu publicznego do PKB według projektu ma wzrosnąć do 52,7% i oczywiście jest to znaczący wzrost w stosunku do tego, co było jeszcze na koniec roku 2019, ale naprawdę jest to jeszcze dość daleki, dość istotny margines w odniesieniu do progu konstytucyjnego.

A więc widać bardzo wyraźnie, że mamy znaczny margines bezpieczeństwa. Oczywiście on jest bardzo potrzebny i wszyscy o tym wiedzą, bo zadłużenie w stosunku do PKB systematycznie, z roku na rok, malało, ale to właśnie dzięki temu, że przez ostatnie lata malało, teraz ten margines mamy i jest możliwość aktywnej interwencji w gospodarkę.

Teraz kolejna rzecz, niezwykle ważna, na której chciałbym się skupić. To dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Patrząc na doświadczenie, które mamy wszyscy.

Kredyty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgały wtedy 30 mld i więcej.

Właśnie teraz jest to przejrzyście, uczciwie pokazywane: dotacja z budżetu państwa. Nie jest ukrywany deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale jest to deficyt budżetu państwa, bo przewidziana dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2021 to prawie 60 mld zł. Nie zakłada się pożyczek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tak jak to było w poprzednich latach.

A więc widać bardzo wyraźnie, że w tych bardzo trudnych czasach rząd przygotował bardzo odpowiedzialny budżet. Oczywiście klub Prawo i Sprawiedliwość będzie ten budżet popierał. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska. Proszę, pani poseł. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Każdy kryzys, także ten wywołany pandemią, jest egzaminem dla rządu. Niestety tego egzaminu PiS nie zdał. Dowodem na to jest dzisiejszy stan finansów państwa, a przecież końca epidemii jeszcze nie widać. Gdyby nie chodziło o Polskę, miałabym pewnie satysfakcję. Z tej mównicy wiele razy ostrzegałam, że nie wolno lekkomyślnie wydawać pieniędzy, których się nie ma.

Rzeczywiście ma pan rację, panie przewodniczący, z liczbami się nie dyskutuje. Taki deficyt powinien być jak kubeł zimnej wody na rozgrzane kolejnymi kampaniami wyborczymi głowy populistycznego PiS-owskiego rządu.

Nikt nigdy nie zdewastował finansów państwa tak jak PiS. Ten budżet też nie jest żadną prognozą. To raczej mieszanina pobożnych życzeń, oszustw i manipulacji. Pierwsze oszustwo to zaniżona inflacja. Drugie oszustwo to zawyżony wzrost PKB. Oczywiście te dwa oszustwa, jedno w dół, drugie w górę, dla budżetu pewnie wyjdą na zero. Problem w tym, że zapłacą za to podatnicy z własnej kieszeni, bo pieniędzy z podatku VAT będzie więcej, niż zapisano w budżecie, bo inflacja będzie wyższa niż założona. Trzecie oszustwo to tradycyjnie już zawyżone inwestycje. Jeśli chodzi o inwestycje, to premier Morawiecki i PiS żyją w jakiejś równoległej rzeczywistości. Oni myślą, że to, co nazwali odpowiedzialnym rozwojem i 4 lata temu pokazali na slajdach, stało się. A przecież wy nie przeprowadziliście żadnej - powtórzę - żadnej inwestycji. Powiedzcie mi, jak to jest, że my dawaliśmy radę, a wam nic w inwestycjach nie wychodzi. Ostatnio wtedy jeszcze wicepremier Jadwiga Emilewicz zaapelowała do Polaków o pomysły na realizację i zagospodarowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Czy wy chcecie inwestować w formule pospolitego ruszenia? Reasumując, inflacja z sufitu, wzrost PKB z sufitu, wzrost inwestycji z sufitu. Czwarte kłamstwo tego budżetu też jest z sufitu. To są wydatki. Przecież w tym budżecie nie ma kilkudziesięciu miliardów złotych, które rząd planuje wydać w roku 2021. Po to, żeby pan przewodniczący Kowalczyk tu stanął i powiedział, że ten wielki deficyt, który wyniesie w przyszłym roku ponad 82 mld, jest przecież mniejszy niż deficyt tegoroczny, wynoszący 110 mld zł. Panie Pośle! To nieprawda. W przyszłym roku jest wyższy niż w tym roku. Piąte oszustwo tego budżetu polega na tym, że z roku na rok finansujecie coraz więcej ze środków pozabudżetowych. Chwali się pan tym ZUS-em, do którego dopłacicie w tym roku. Zła wiadomość, szczególnie dla młodych Polaków, jest taka, że każdego roku będziemy dopłacać więcej do rent i emerytur. Natomiast wracając do tego kolejnego oszustwa, czyli wydatków finansowanych spoza budżetu, chcę powiedzieć, że PiS namnożył tyle agencji, funduszy, państwowych osób prawnych, że już nikt nie wie, kto, ile i na co wydaje. Minister finansów nie ma o tym zielonego pojęcia. Dokładnie taką samą wiedzę o finansach miał minister finansów Grecji, kiedy w 2010 r. na posiedzeniu Ecofin przepytywali go, a on po prostu w ogóle nie miał pojęcia o prawdziwym stanie tych finansów. I wreszcie ostatnie kłamstwo, o którym zdążę powiedzieć, bo fakt, że mamy 15 minut, to jest w ogóle kpina, ale nie z Wysokiej Izby, to jest kpina z obywateli, a więc ostatnie kłamstwo, o którym zdążę powiedzieć, to kłamstwo o obniżaniu podatków. Ciągle słyszymy: obniżymy PIT, obniżymy CIT. Jeśli porównacie sobie nowe podatki, które wprowadzacie: cukrowy, od sprzedaży detalicznej i opłatę mocową, to wiecie, ile Polacy zarobią na obniżeniu PiS-owskich podatków?

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt budżetu na 2021 r. zakłada drugi największy deficyt w historii, po tegorocznym budżecie. Ale w uzasadnieniu próżno by szukać przyczyn, dla których ten deficyt ma wynieść aż 82 mld zł, czyli 4% PKB z grubsza licząc. Trudno zrozumieć, dlaczego przy wzroście PKB o 4% w stosunku do roku bieżącego i wzroście dochodów podatkowych o 5,5% sytuacja w budżecie musi być taka zła. Są dwa wyjaśnienia: albo to jest kolejny przykład nieudolności rządzenia Zjednoczonej Prawicy, która nawet przy wzroście gospodarczym 4%–4% realnie to jest 6% nominalnie - nie jest w stanie doprowadzić do zrównoważenia finansów, albo po prostu mamy do czynienia z kontynuacją tegorocznej polityki skoku na kasę pod pretekstem pandemii.

W tym i przyszłym roku dług według metodologii krajowej ma wzrosnąć łącznie - mówił o tym pan przewodniczący Kowalczyk - o ponad 250 mld zł, ale według metodologii unijnej ma on wzrosnąć o ponad 465 mld zł. Bardzo chętnie posługujecie się metodologią krajową, żeby po prostu zaniżyć faktyczne rozmiary długu i oszukać Polaków odnośnie do tego, na ile rzeczywiście zadłużacie ich, ich dzieci i ich wnuki.

Przede wszystkim są to oczywiście wydatki związane z zaciąganiem pożyczek przez fundusz COVID-owski i przez Polski Fundusz Rozwoju. No więc przyczyną tych rozbieżności jest wasza pokrętna polityka polegająca na przenoszeniu tych właśnie wydatków poza sektor finansów publicznych określony w ustawie. Ale metodologia oparta na tej definicji jest po prostu coraz mniej wiarygodna i nie pokazuje rzeczywistych rozmiarów długu. Natomiast metodologia unijna, bardziej obiektywna i zunifikowana dla całej Unii, pokazuje, że na koniec przyszłego roku dług wyniesie 1510 mld zł i to nie będzie 52% czy 54% PKB, tylko 64% PKB, panie przewodniczący, a to oznacza, że ten dług jest znacznie powyżej poziomu konstytucyjnego.

Ale ponieważ się tego boicie, robicie wszelkie sztuczki po to, żeby ukryć faktyczny stan finansów publicznych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Marek Hok, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Budżet państwa miał przejąć finansowanie polskiej ochrony zdrowia. Tak się nie stało. Dzisiaj w dalszym ciągu ochronę zdrowia utrzymują, finansują obywatele, Polacy, wszyscy pacjenci, którzy płacą składkę zdrowotną - to jest główne finansowanie ochrony zdrowia.

Dzisiaj polskie szpitale tylko w wyniku epidemii COVID. Na Śląsku 23 szpitale powiatowe zadłużyły się o kolejne 200 mln zł.

To były obietnice. Z czego mają otrzymać wynagrodzenia? Z finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia dla dyrektorów szpitali, którzy muszą się zastanawiać, czy kupić leki onkologiczne, czy kupić maseczki, czy pokryć koszty wzrastających opłat za gaz, za światło, za wszystkie dostawy?

Bez znaczącego, skokowego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia nigdy nie poradzi sobie z tą dramatyczną sytuacją. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! O budżecie na przyszły rok rozmawiamy w bardzo trudnym momencie dla polskiej gospodarki, nie tylko polskiej.

Po 5 latach życia na kredyt, nieodpowiedzialnej polityki, niesłuchania ekspertów i opozycji, po 5 latach ignorowania naszych gospodarczych poprawek i projektów ustaw, przedstawiacie budżet pokazujący głęboki deficyt i katastrofę.

Tak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki na wrześniowej konferencji prasowej. To sprawdźmy, jak to odbicie, panie premierze, będzie wyglądało.

Niespełna 19%.

Rząd PiS wprowadził już aż 34 nowe podatki - nie będę ich wymieniać, wszyscy o nich wiemy.

Dziś jest on gigantycznych rozmiarów i tym budżetem planujecie ten pożar ugasić. Skutki będą opłakane. Przedstawiony projekt ustawy jest antyrozwojowy. Jest on efektem waszej nieodpowiedzialnej polityki gospodarczej. Najsmutniejsze jest to, że skutki będą ponosić zwykli Polacy, o których tak dużo mówicie (Dzwonek), a nie wasi koledzy poupychani w spółkach Skarbu Państwa. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Wieczorek, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Chciałbym zobaczyć, jacy to eksperci, bo jeżeli rzeczywiście tacy są, to warto o tym podyskutować. Mam wrażenie, jak rozmawiamy o tym dokumencie, że to jest raczej dokument na ten moment przypominający literaturę fantastyczną, raczej powieść science fiction niż rzeczywiście dokument, który odzwierciedla realne finanse i poważne podejście polskiego rządu do finansów państwa w trakcie pandemii i po pandemii, bo mam nadzieję, że niedługo z tym wirusem, z tym problemem się uporamy.

Można powiedzieć, że pewnie w trakcie przygotowywania tego budżetu pan minister finansów nucił sobie piosenkę niczym ze Stadionu Narodowego: nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.

Mamy wrażenie, że niestety rządzący dalej uważają, że można prowadzić taką kreatywną księgowość, że można tworzyć wirtualne budżety, że można tworzyć wirtualne prognozy i że to wszystko będzie akceptowane.

Prawda jest taka, że lepiej znać tę najgorszą prawdę, niż żyć w świecie iluzji i wzajemnie się oszukiwać. Prawda jest taka, że jeżeli tak będziemy dalej robić, to przyszłe pokolenia, nasi następcy, ani wam, ani nam tego nie wybaczą. Więc, panie ministrze, dzisiaj przede wszystkim chcemy usłyszeć, jak wygląda rzeczywiście sytuacja finansów państwa.

Prawda jest taka, że dzisiaj każde dziecko narodzone w Polsce, także z programu 500+, którym tak się chwalicie, od razu ma na głowie 34 tys. długu państwowego, który będzie przez lata swojej pracy niewątpliwie musiało spłacać. Pytanie, czy to będzie tyle, czy będzie tego jeszcze więcej.

Przypomnę tylko, jaki był plan w styczniu tego roku, jeszcze raz, że to miał być budżet bez deficytu. Okazuje się, że już jest 109 mld zł, natomiast oczywiście wiem, znamy tę narrację, że to jest wina COVID-u, to jest wina pandemii. Jasne, niewątpliwie to ma ogromny wpływ na to. Tylko chcę też zwrócić uwagę, bo te same błędy popełniacie w tej chwili, w mojej ocenie, że to samo robiliście w przypadku tego budżetu zerodeficytowego, bo ileś tych wydatków - w formie pożyczek, tricków finansowych, przygotowanych przez ministra finansów, i trzeba to docenić - znalazło się poza budżetem. Wystarczy dowiedzieć się, jak wypłacono trzynastą emeryturę. Pożyczka z budżetu państwa dla Funduszu Rezerwy Demograficznej, Fundusz Rezerwy Demograficznej pożycza Funduszowi Solidarnościowemu, później Fundusz Solidarnościowy wypłaca trzynastą emeryturę. On oczywiście w tych dokumentach już zostanie rozwiązany i już widać jak, ale jeszcze będę trzymał państwa w niepewności, na koniec o tym powiem.

Tutaj plan dochodów jest na poziomie 404 mld, wydatki - 486 mld, deficyt planowany na 82 mld zł. I dzisiaj już rodzi się pytanie w tym kontekście: Czy to jest deficyt realny, czy czasami ten deficyt nie będzie większy? Rodzi się również pytanie: Czy rząd i rządząca większość mają pomysł na gospodarkę polską po pandemii? Czy pomysłem jest podnoszenie podatków? Czy pomysłem jest wstrzymanie inwestycji? Czy budżet na rok 2021 rzeczywiście odpowiada na pytanie, jak będziemy sobie radzić gospodarczo jako Polska po tym wielkim kryzysie? I żeby była jasność, odpowiedź jest bardzo prosta. Ten projekt budżetu na tym etapie - ale wierzę, że pan minister tych głosów słucha, i wierzę, że będzie też z tego wyciągał wnioski - ten budżet nie odpowiada na żadne z tych pytań. Bo w naszej ocenie, i to mówi polska Lewica, dzisiaj budżet na czas kryzysu, budżet na czas po pandemii, budżet na rok 2021 to powinien być budżet, my to nazywamy, 3P - budżet proinwestycyjny, budżet propracowniczy i budżet prozdrowotny. Bo dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z dwoma kryzysami - mamy do czynienia z kryzysem w ochronie zdrowia i mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym. I teraz zobaczmy, jak planujemy sobie poradzić z tymi dwoma kryzysami. Otóż jeżeli chodzi o stronę dochodową, 6 mld więcej w stosunku do roku 2020, czyli 404 mld zł.

Pytanie: Czy to jest realne czy nierealne?

Oczywiście to można tłumaczyć również jednym z projektów ustaw, który dzisiaj jest procedowany. Jeżeli chodzi o PIT, planujemy duży wzrost, w związku z czym jest pytanie: Czy wzrost wpływów z PIT-u to efekt planowanego wzrostu podatków czy dodatkowych obciążeń dla pracowników?

Czy rzeczywiście też realnie jest to ocenione? Myślę, że czas pokaże. I tutaj też mamy zastrzeżenia, że być może te założenia nie do końca są realne.

Otóż, żeby była jasność, tych środków z deficytu budżetowego, z tych pożyczek i tych kredytów na pewno nie wydamy na podwyżki dla sfery budżetowej, bo wskaźnik wynagrodzeń w sferze budżetowej jest planowany tak jak do tej pory na poziomie 100%. Nie wydamy tego na ochronę zdrowia, bo rzeczywiście jest planowane 5,3 PKB, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, a więc nadal będziemy na szarym końcu, jeżeli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia w państwach Unii Europejskiej. W związku z czym tych środków, mimo że mamy do czynienia z pandemią i z kryzysem, na to nie wydamy. A na co będziemy wydawać?

15 mld wydajemy na wydatki majątkowe dotyczące polskich Sił Zbrojnych. Jest pytanie, czy to jest najważniejszy dzisiaj problem. Czy rzeczywiście z koronawirusem będziemy walczyli F-35 czy armatami, czy pistoletami? Nie wiadomo, dlaczego to robicie, bo 63% wszystkich planowanych inwestycji zostanie zrealizowanych przez wojsko. Do tego wydatki majątkowe na drogi w tym kontekście to jest kwota 1,43 mld zł. Ja wiem, że pan przewodniczący mówił tu o 6 mld, ale zaraz zobaczymy, co tam się dzieje wokół tego budżetu i zobaczymy, że te 6 mld też jest iluzoryczne. Ale, żeby była jasność, stać nas na to, żeby przekazać papiery wartościowe dla telewizji publicznej na kwotę 1,95 mld zł. W związku z czym popełniamy dalej te same błędy, które popełnialiśmy w 2020 r. Jeżeli chodzi o obsługę długu - 28 mld zł, to tyle będzie nas kosztowała ta obsługa długu publicznego.

Ale w tym wszystkim rzeczywiście musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że de facto osobne dwa budżety znajdują się poza tym budżetem.

Pytanie: na co? Chcecie kupować TVN, czy chcecie kupować inne prywatne media? Wiele tych jednostek pozabudżetowych zakłada straty, w związku z czym, żeby była jasność, one i tak wcześniej czy później, w taki czy inny sposób, wrócą do budżetu i co do tego nie ma żadnej wątpliwości.

Na koniec jest rozwiązanie tej zagadki, o której na początku powiedziałem - Fundusz Solidarnościowy.

No i cóż te 11 mld deficytu? Coś się z tym musi stać, bo przecież jest 11 mld, coś się musi stać. A więc jak przejrzymy następny projekt ustawy, to się okaże, że tam się to staje. Tam się po prostu umarza te wszystkie pożyczki, więc jeżeli chodzi o ten cały bajer na początku o zrównoważonym budżecie, to tutaj się okazuje, że wcale nie był on taki zrównoważony, tylko zaciągaliśmy sobie pożyczki, które dzisiaj, mówiąc krótko, umarzamy. W związku z tym zwracamy się z apelem do pana ministra: zejdźmy na ziemię, zejdźmy z tego finansowego kosmosu [[Dzwonek]] i rzeczywiście pracujmy nad budżetem proinwestycyjnym, propracowniczym i prozdrowotnym. Tylko taki budżet poprze polska Lewica. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Szanowni Państwo! Projekt budżetu na 2021 r. powinien być kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym, europejskim, krajowym lockdownie, wywołanym przez COVID-19. Wymieniam tu świat, Europę, kraj, bo te gospodarki są powiązane. Problem w tym, że mamy drugą falę pandemii. Nie wiemy, jakie przyniesie skutki zdrowotne dla społeczeństwa i dla gospodarki, jak przełoży się na sytuację finansów publicznych.

Oczywiście są też optymistyczne założenia rządu co do działań proinwestycyjnych, kontynuacja programów społecznych, o czym za chwilę. Natomiast jeśli patrzy się na liczby, to chciałbym jeszcze raz podkreślić, że zadłużenie, dług sektora finansów publicznych według metodologii unijnej będzie na poziomie 6%, a zadłużenie - na poziomie 64,7% PKB.

Bo sytuacja jest wyjątkowa.

To musi być połączone. Oczywiście chodzi o to, o czym mówiłem: rząd zamierza kontynuować priorytetowe programy polityki społeczno-gospodarczej. Ja ich nie będę wymieniał, są powszechnie znane. Ale jakoś nie doczytałem się wielkości finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa. Wiemy, czym jest mieszkanie dla młodych ludzi, dla stabilizacji, to jest wyjątkowo ważne. Podobnie nie ma więcej informacji na temat zadań, jak będą finansowane sprawy, jakie obszary - z Funduszu Solidarnościowego.

Wreszcie sprawy związane z zadłużeniem. Mówił o tym pan poseł prof. Rosati. Ta wielkość jest rzeczywiście.

Wreszcie chciałbym przejść do problemów, jeśli chodzi o przejrzystość finansów. Jest ona utrudniona poprzez wykazanie niektórych przyszłych wydatków w roku 2021 w tegorocznym budżecie, kiedy - jak wiemy - nie obowiązuje nas reguła wydatkowa. A więc wymyślono strategię zapakowania do maksimum tegorocznego budżetu wydatkami na papierze, których ze względu na brak czasu nie da się zrealizować w ciągu tego kwartału.

Podatek cukrowy też będzie wchodził.

Pewne szanse daje nam to, że nasze funkcjonowanie na rynku unijnym jest związane z pewną zależnością od tego, co się dzieje w gospodarce niemieckiej czy w innych gospodarkach.

To nie udało się naszym negocjatorom.

Musi być pewne nowe podejście restrukturyzacyjne, które pozwoli na unowocześnienie gospodarki, na innowacyjność, na sprostanie wymogom inteligentnego rozwoju.

Bardzo mnie ciekawi, na ile za koncepcje, za rozwój, za strategię będzie odpowiedzialne Ministerstwo Finansów, a na ile będzie odpowiedzialne ministerstwo rozwoju. Po prostu ważne jest, żeby był autor, żeby były osoby odpowiedzialne, które będą czuwały nad prowadzonymi zmianami, bo te zmiany to jednocześnie pewna transformacja gospodarki, a nie tylko walka z kryzysem gospodarczym. Głos ma pan poseł Krzysztof Paszyk, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dobry budżet państwa to taki budżet, który odpowiada potrzebom mieszkańców kraju, którego dotyczy. Analizując ten budżet, który pan minister zaproponował, trudno odnieść wrażenie, że on faktycznie odpowiada tym potrzebom. Jeden przykład, który już w tej Izbie padał: dzisiaj potrzeby są po stronie polityki zdrowotnej, a nie polityki obronnej, panie ministrze.

Pytanie, dlaczego nie znajduje on zrozumienia po stronie rządu. Obawiam się, że ciągle bardzo znaczące, mentalne oddziaływanie mają słowa pana premiera, że epidemia już sobie poszła, że nie trzeba się jej bać.

Jeśli chodzi o rolnictwo, panie ministrze, to pan być może jest daleko od tych spraw związanych z rolnictwem, z wyzwaniami, które stoją przed rynkami rolno-spożywczymi. Pewnie to jest też trochę tak, że nowy minister zaczyna proces zamykania, zwijania polskiego rolnictwa, bo już jedna ustawa mu się prawie udała, ale zmniejszenie o 80% poziomu środków budżetowych na stabilizację rynków rolnych w stosunku do roku 2020 zakrawa na jakiś skandal.

Trzecia rzecz. Przed rokiem prezes Kaczyński bardzo mocny nacisk położył na transport, na rozwijanie połączeń.

To jest 65-procentowy spadek. A jak nie było w zeszłym roku, tak nie ma, np. połączeń autobusowych z Rzeszowa do stolic sąsiednich regionów, do Białegostoku, do Olsztyna. Jak ze stolicy województwa opolskiego nie było połączenia autobusowego do Warszawy, tak nie ma. Prezes Kaczyński z pewnością, panie ministrze, na to będzie zwracał pana uwagę. To miało być sztandarowe działanie rządu Zjednoczonej Prawicy skierowane właśnie w stronę samorządów. Już, widzę, przestało takie być, wybory się skończyły, nie ma. Zdumiewa to, dlaczego jest 200 mln mniej na Policję, 60 mln - na Państwową Straż Pożarną. Przecież wczoraj kto stał koło ministra zdrowia? Ano komendant główny Policji, który zapewniał o polityce zero tolerancji.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przede wszystkim uważam, panie ministrze, że tak ważna konstytucyjnie osoba jak pan w tym rządzie nie powinna w sposób lakoniczny potraktować informacji na temat najważniejszej ustawy w najbardziej trudnym czasie, w jakim znalazła się Polska. Uważam, że jest ujmą dla pana to, w jaki sposób pan zaprezentował ten budżet. Dlaczego pan z sercem nie podszedł do sprawy systemu ochrony zdrowia? Przecież są takie sytuacje w naszym kraju, że sanepid zawiesza jakąkolwiek inną działalność niż działanie na rzecz walki z koronawirusem. Są urzędy miast, które delegują na początku na szkolenia, a później do pracy w sanepidzie. To są dzisiaj najważniejsze sprawy.

Dzisiaj o tym powinien powiedzieć minister finansów. Są sytuacje ludzi, którzy przychodzą do mojego biura, i mówią, że nie mogą się dostać do publicznej ochrony zdrowia, idą do prywatnej, a tam jest ściana, a pieniądze od nich pęsetą się bierze.

Witam ponownie. Wracamy na bal maskowy, ale widzę, że dalej atmosfera drętwa. Lepiej się czasem dostosować. Ta zabawa musi się źle skończyć. Ale rząd się tym nie przejmuje. Roztrwoniliśmy pieniądze w czasie dobrej koniunktury, wydawaliśmy pod korek, żyliśmy od pierwszego do pierwszego, wtedy kiedy szło nam dobrze, to teraz, kiedy idzie gorzej, siłą rzeczy musimy się znaleźć pod korkiem. Ten budżet to jest jedno wielkie wyparcie rzeczywistości. Ten budżet to jest brnięcie w politykę, która zaprowadziła nas już na skraj bankructwa. I wy prosto w to bankructwo zmierzacie - w objęcia hiperinflacji i większego kryzysu. Zwracam uwagę na to, na co kilka razy już zwracałem tutaj uwagę, że nie da się samego siebie podnieść za włosy do góry.

Skoro państwo wierzycie, że w skali makro to działa, że wystarczy zebrać od ludzi więcej pieniędzy, potem im je rozdać i wszyscy będą dzięki temu bogatsi, zróbmy to samo w Sejmie. Zamiast sobie podwyższać wynagrodzenia zróbmy jakiś fundusz docelowy, wszyscy się zrzucimy, potem jacyś nasi najwybitniejsi przedstawiciele będą to rozdawać w postaci jakichś programów, funduszy, zapomóg stymulacyjnych i na pewno dzięki temu rozruszamy nasze budżety. Jeszcze się trochę zadłużymy na koszt przyszłych kadencji i na pewno będzie dobrze. Jeśli wierzycie, że to działa, to zastosujcie najpierw na sobie, a potem dopiero na żywej tkance organizmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan poseł Krzysztof Bosak.

To bardzo proszę zejść z mównicy i włożyć maskę.

W tej sytuacji przejdziemy do pytań.

Mam podstawę prawną w postaci jednogłośnego ustalenia Prezydium Sejmu.

No to mam przyłbicę. Proszę się nie bać krytyki ze strony opozycji. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Konieczny. O, bardzo proszę, ale czas panu już się wyczerpał. Tak więc, jak powiedziałem, pozwolę sobie wygłosić krytykę budżetu państwa mimo utrudnień ze strony pana marszałka.

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku!

Bardzo proszę, panie pośle. Rok 2021, nad którego budżetem teraz dyskutujemy, to będzie rok, w którym, mamy nadzieję, Polska wyjdzie z kryzysu gospodarczego. Jak pokazuje historia kryzysów gospodarczych, to muszą być inwestycje publiczne, bo z kryzysów rzadko wychodzi się za pomocą inwestycji prywatnych. Tymczasem budżet na inwestycje zaplanowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości to mniej niż 25 mld, to bardzo mało. Co jest najbardziej szokujące? Aż 63% z tej sumy to są inwestycje na wojsko. Że nie ma ważniejszych inwestycji w Polsce, że program „Mieszkanie+” okazał się tak gigantycznym sukcesem, że nie musimy już inwestować w mieszkania, że Polacy mieszkają w fantastycznych, przestronnych mieszkaniach i mają kłopot, żeby się w nich znaleźć? W tym momencie mamy ogromny problem z przeludnieniem, potrzebujemy inwestować w kolej, bo wciąż połączenia kolejowe w Polsce są niezadowalające i nieporównywalnie gorsze od tych chociażby na zachodzie Europy. Pomimo tego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce inwestować w transport publiczny, nie chce inwestować w kolej, nie chce inwestować w mieszkania, nawet po absolutnej klęsce programu „Mieszkanie+” Wydaje 63% sumy na inwestycje na wojsko. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Joński. Nadal nie ma pana posła? Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym na początku zapytać, w którym punkcie, w której pozycji tego budżetu są zapisane oszczędności wynikające z odchudzenia rządu, który wczoraj został zaprzysiężony.

Interesują mnie przede wszystkim obwodnice w województwie łódzkim: Brzeziny, Łowicz, Wieluń, Błaszki i Srock.

Bardzo wiele mówiliście na ten temat. Chciałbym także dowiedzieć się, ile pieniędzy zarezerwowaliście na wsparcie samorządów, szczególnie w wymiarze systemu ochrony zdrowia i oświaty.

Chciałbym uzyskać odpowiedź przede wszystkim na te pytania. Ile pieniędzy zarezerwowaliście na kupno w przyszłym roku szczepionek na grypę oraz na jedyny lek (Dzwonek) akredytowany przez Europejską Agencję Leków, czyli Remdesivir? Pani poseł Izabela Leszczyna, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Ze zdziwieniem słuchałam pana ministra finansów i przewodniczącego komisji finansów, którzy z takim samozadowoleniem opowiadali, że oto w roku pandemii, bo przecież koronawirus będzie z nami także w przyszłym roku, realizują swój mało ambitny plan dochodzenia latami do 6% PKB na zdrowie i oto w przyszłym roku będzie już 5,3% PKB. Pierwsze pytanie do ministra finansów: Czy pan minister uważa, i zgadza się z tezą, że system ochrony zdrowia potrzebuje więcej pieniędzy w czasie epidemii niż w czasach, kiedy epidemii nie ma? Jak już na to retoryczne, zdawałoby się, pytanie pan minister odpowie, to chciałabym, żeby pan minister wskazał, i proszę o odpowiedź nie tylko z mównicy, ale także na piśmie: Jeśli Polacy wpłacą na NFZ w przyszłym roku ponad 103 mld zł, to żeby zrealizować te 5,3%, ile miliardów złotych musi dopłacić budżet? Proszę wskazać miejsca, w których w budżecie te brakujące środki do 5,3% PKB państwo przewidujecie?

Pan poseł Robert Kwiatkowski, klub Lewicy. Dzień dobry. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jakże się cieszę, że jest z nami pan minister Piotr Patkowski, bo do niego adresowane jest pytanie. O co? O lukę VAT-owską, panie ministrze. To źródło sukcesu finansowego, dzięki któremu można było rzekomo sfinansować liczne programy socjalne rządu PiS-u. Dobrze, że je sfinansowano, ale argumentowano przy okazji, że dzieje się to w ten sposób, że gromi się liczne mafie VAT-owskie i dzięki temu są pieniądze na rzeczone programy socjalne.

Chyba że moje informacje są nieaktualne. Przyznacie państwo, że przy kwocie podatku od towarów i usług, wpływów przewidywanych na kwotę 181 mld, to te 40 mld robi wrażenie. Pytanie brzmi tak: Co z tym zrobicie? Zaangażujecie ministra Kamińskiego? Przedstawicie nową interpretację? Jakie będą odpowiedzi w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszyscy powtarzamy, że sprawy ochrony zdrowia i gospodarki powinny być najistotniejsze. A jak jest, szanowni państwo? Niewielki wzrost. Macie, szanowni państwo, niesamowitą okazję poradzić sobie z ogromnym, galopującym zadłużeniem szpitali powiatowych. Czy macie państwo realną propozycję? Nie, nie macie, szanowni państwo. Pochwała, panie ministrze, jeśli chodzi o inwestycje, tak. Musimy jak najwięcej na te inwestycje dawać, bo to pobudza naszą gospodarkę. Mamy tę szansę, możemy to zrobić.

To jest kilka miliardów złotych dopłacanych w sumie przez samorządy powiatowe do funkcjonowania tych szpitali.

To jest pewna refleksja, panie ministrze. Pan poseł w masce? Pani poseł Mirosława Nykiel, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, pan nie ma maski.

Być może coś w tym jest.

ponieważ to, co pan czynił nierozważnie, powtarza pan po chwili namysłu, na który dał pan sobie sam czas. Teraz, po namyśle, jest pan już przestępcą recydywistą i trwa pan w przestępczym uporze. Niech pan tego nie czyni, panie marszałku.

Sąd weźmie to pod uwagę jako okoliczność łagodzącą.

Panie pośle, proszę mi umożliwić wystąpienie. Bardzo proszę, pani poseł. Panie marszałku, dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! pani zajmuje czas przeznaczony dla mnie w tej debacie. Pani zajmuje ten czas, który przeznaczony jest dla mnie.

Proszę nie posuwać się do rękoczynów czy raczej tyłoczynów, panie pośle. proszę wezwać Straż Marszałkowską, ponieważ w tej sali dokonuje się czynów przestępczych już całkiem seryjnie.

Wysoki Sejmie, zwołuję Konwent Seniorów na godz. 17 w gabinecie marszałka. Ogłaszam przerwę do godz. 17.10.

Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 6. porządku dziennego.

Wysoka Izbo! Ja powrócę, z uporem maniaka do inwestycji, bo żeby realizować te piękne programy społeczne, to musimy mieć z czego. A jak nie będzie inwestycji, to z czego będziecie realizować te wspaniałe programy społeczne? Pamiętacie państwo „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którą z taką dumą prezentował premier Morawiecki, jeżdżąc po kraju? Jedną z pułapek rozwoju, którą zdiagnozował, jedną z ważniejszych, był niski poziom inwestycji, niska stopa inwestycji. Założył, że będzie to 25%.

Siłą napędową miały być te wielkie inwestycje: Centralny Port Komunikacyjny, elektrownia w Ostrołęce, 100 tys. mieszkań, milion aut elektrycznych. Żadna z tych inwestycji nie została zrealizowana.

Panie ministrze, pytam: Co ma być podstawą rozwoju gospodarczego [[Dzwonek]] Polski w 2021 r. Nie ma pana posła.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od kilku debat związanych akurat z kwestiami budżetowymi konsekwentnie pytam o kwestie spadku nakładów na rolnictwo w budżecie polskim.

Bo ten trend jest niepokojący, chociażby ze względu na liczne wyzwania, które stoją akurat przed szeroko pojętym działem - rolnictwo. No chociażby Inspekcja Weterynaryjna. Szerzące się choroby zwierzęce, które mają charakter epidemiczny, wymagają silnego wzmocnienia tejże inspekcji. Drugim elementem jest sprawa dotycząca wody i interwencji w tym zakresie. Tutaj mamy do czynienia z wieloletnimi oczekiwaniami w niektórych regionach. Podam przykład południowej Wielkopolski - zbiornik Wielowieś Klasztorna, który jest przygotowany od strony gruntowej, ale jednocześnie on też wymaga, że tak powiem, jeszcze wsparcia, żeby ten przewidziany termin rozpoczęcia realizacji - rok 2023 był realny, żeby to się rzeczywiście rozpoczęło, bo to jest jedna z największych inwestycji, jeżeli chodzi o Wielkopolskę w zakresie retencji wodnej. Pan poseł Jakub Kulesza, koło Konfederacji. Nie ma pana posła. Pan poseł Arkadiusz Marchewka, klub Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Doskonale pamiętam, jak z tej mównicy premier Morawiecki mówił o tym, że pieniędzy wystarczy na wszystkie obietnice i nie trzeba będzie zaciągać żadnego długu. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

To rekord. Dla przeciętnego Polaka to są liczby abstrakcyjne, ale żeby powiedzieć, co to znaczy, to trzeba powiedzieć jasno, że każdy z was: pan, panie pośle, pan, panie pośle, wszyscy Polacy będą mieli kredyt w wysokości 40 tys. zł. Zadłużacie Polskę w rekordowym tempie. W ciągu ostatnich 5 lat zwiększyliście dług publiczny o ponad 500 mld zł. Chciałbym zadać pytanie: Czy uważacie, że to jest odpowiedzialne prowadzenie polityki państwa? Czy to jest prowadzenie spraw kraju z myślą o przyszłym pokoleniu? Nie. Mam takie poczucie, że myślicie tylko o tym, co zrobić tu i teraz, żeby wypełnić obietnice, na które nie ma dziś pieniędzy. Musicie te pieniądze pożyczyć i później się tym nie musicie martwić, bo pewnie to spadnie na waszych następców, a te długi będą musiały spłacić [[Dzwonek]] kolejne pokolenia. Bardzo dziękuję. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! W czasie pierwszego czytania nowelizacji tegorocznego budżetu, odpowiadając na moje pytanie dotyczące wsparcia Krakowa i Małopolski w organizacji europejskich igrzysk olimpijskich w 2023 r., powiedział pan, że zamierza zwiększyć budżet Ministerstwa Sportu na rok 2021 o kwotę 56 mln zł. Kiedy przyglądam się tej projekcji na rok 2021, to w części 25 tego nie dostrzegam. Co prawda jest pozycja dotycząca rezerwy celowej nr 37, ale tam jest 30 mln, i jest ta rezerwa pt.: upowszechnianie sportu. Myślę, że tu chodzi głównie o wsparcie infrastruktury sportowej oraz przygotowanie logistyczne tej dużej europejskiej imprezy.

Na 2021 r. zaplanowano tylko kwotę 400 mln zł.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Czesław Siekierski, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Czy to jest szacunek NBP-u? Bo dotychczas te wpływy były większe, w zależności oczywiście od roku.

Jeśli chodzi o samorząd, to państwo mówią, że rosną wpływy dla samorządu z tytułu zwiększonych podatków i inne wpływy, a samorządy mówią, że przez obniżki różnych podatków mają mniejszy udział. Jak to w rzeczywistości jest? Ile będzie finansował rząd, a ile muszą dopłacić samorządy? Wreszcie pan poseł Grzyb pytał o zielony ład.

To są istotne informacje dla rozmowy o przetargu w Unii, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy inne możliwości pozyskania środków z Unii. Bardzo dziękuję. Pani poseł Klaudia Jachira, klub Koalicja Obywatelska. Wicepremierze Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać, kiedy rząd, zamiast zadłużać Polskę, pomyśli wreszcie o oszczędzaniu, szczególnie w czasie pandemii. Oto paragon wydatków PiS-u, niepotrzebnych wydatków PiS-u.

W niecałą minutę znalazłam państwu w zaokrągleniu 29 mld zł oszczędności, a ta lista niepotrzebnych wydatków jest długa, bo te długi, nomen omen długi, będziemy spłacać latami, tak jak nasi rodzice spłacali pożyczki Gierka.

Wysoka Izbo! Podczas dzisiejszej debaty na temat nowelizacji tegorocznego budżetu zwracaliśmy uwagę na naszym zdaniem kuriozalne pomijanie potrzeb systemu edukacji w warunkach kryzysu. Dokładnie te same zarzuty można byłoby powtórzyć pod adresem przyszłorocznego budżetu, choć przynajmniej my na lewicy mamy nadzieję, że kryzys w 2021 r. nas jednak opuści. Państwo jednak wydają się robić bardzo dużo, żeby przynajmniej w edukacji ten kryzys dalej trwał.

Jak szacują związki zawodowe, jak podają kuratoria oświaty, we wrześniu ze szkół odeszło nawet 10 tys. nauczycieli. Moje pytanie do państwa jest takie: Jak chcecie zatrzymać tę katastrofę kadrową w edukacji, jeżeli nie przewidujecie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, których już teraz, już w tym roku zaczyna brakować? Dziękuję. Pani poseł Zofia Czernow, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dwa pytania konkretne. Pierwsze: Jakie środki finansowe rząd zabezpieczył na realizację narodowej strategii onkologii w 2021 r. I drugie: Co dalej z finansowaniem polskiej oświaty? Dlaczego rząd, wiedząc, że wysokość subwencji oświatowej jest niewystarczająca i powoduje zapaść finansową w polskiej oświacie, nie zabezpiecza niezbędnych środków na ten cel w 2021 r. Szacuje się, że niedobór w oświacie wynosi ok. 20% przyznanych środków w 2020 r., a tymczasem wzrost w projekcie budżetu na rok 2021 wynosi zaledwie 4%. Samorządy nie mają absolutnie pieniędzy, żeby dofinansować brakujące środki na prowadzenie oświaty, a jest to zadanie państwa. Proszę, panie ministrze, o odpowiedź, co dalej z finansami w polskiej oświacie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przewiduje się, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o ponad 36 mld zł, tj. o 8,4%, w tym dochody podatkowe budżetu będą niższe o ponad 40 mld zł, tzn. o 10,3% w stosunku do kwot pierwotnie planowanych na bieżący rok.

Stąd też moje pytanie.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W budżecie na przyszły rok znajdują się też środki dla nowego ministra do spraw samorządów. Na razie nie wiemy, czym zajmować się będzie minister Michał Cieślak. On sam w rozmowie w Radiu TOK FM przyznał, że jeszcze nie zna zadań, jakie postawił przed nim premier, ale zapewnia, że chciałby przygotować jakiś zarys reformy samorządowej. Od dłuższego czasu krążą jednak informacje, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach parlamentarnych weźmie się za samorządy w celu ich zawładnięcia i ograniczenia kompetencji. Za chwilę minie właśnie pierwszy rok tej kadencji Sejmu, dlatego mam pytanie: Czym zajmować się będzie nowy minister do spraw samorządów i jakie zadania będzie miał do zrealizowania? Czy został powołany po to, by wspierać i pomagać lokalnym samorządom, czy też, broń Boże, jest wręcz przeciwnie i włodarze gmin i powiatów powinni zacząć się bać? Pani poseł Monika Falej, klub Lewica. Wysoka Izbo! Czy został on skorelowany z potencjalnymi skutkami pandemii i zwinięcia gospodarki, co pociągnie za sobą spadek popytu na rynku konsumpcji detalicznej? To moje pierwsze pytanie. Kolejne pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, ile środków rząd zamierza przeznaczyć na rekompensatę dla samorządów za utracone wpływy. Szczególnie interesują mnie samorządy województwa warmińsko-mazurskiego.

Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Krzysztof Truskolaski, klub Koalicji Obywatelskiej. Uprzejmie informuję Wysoką Izbę, że nie będę uwzględniał usprawiedliwień, chyba że ktoś uczestniczy w posiedzeniu komisji.

Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oznacza to, że nasz kraj na każde wypracowane przez obywateli 4 zł będzie musiał pożyczyć 1 zł.

Ile w rekordowym budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie przeznaczone na polskie zakłady zbrojeniowe, które w chwili obecnej są na granicy upadku? Ile z tych środków zostanie przeznaczonych na polski przemysł obronny, a ile wzmocni przemysł obronny Stanów Zjednoczonych? Pytanie drugie. Dziękując panu premierowi za ujęcie drogi S10 na odcinku pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, mówiłem, że będę ciągle pytał o to, jakie są środki na tę inwestycję. W związku z tym pytam, ile tych środków będzie w roku 2021. I trzecie pytanie: Ile środków zostanie przeznaczonych w poszczególnych ministerstwach na zatrudnienie makijażystek? Chciałbym w imieniu moich wyborców zapewnić pana premiera Sasina, że ilość pudru nie będzie oceną pana ministra, [[Dzwonek]] tylko ilość środków finansowych wygenerowanych przez firmy, którymi pan zarządza.

Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na koniec grudnia 2018 r. wartość wszystkich akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa przekraczała 190 mld zł. W budżecie na 2021 r. zaplanowano zaledwie 386 mln wpływów z dywidend. Z taką efektywnością pracuje ten rząd. Właściciele wyrzuciliby taki zarząd po pierwszej takiej informacji, a minister, premier Sasin kupuje puder, żeby rzeczywistość przypudrować. Klęska w programach mieszkaniowych, w odtwarzaniu połączeń kolejowych, autobusowych, ale ministrowie pozostają bez zmian. Budżet 2021 r. to także znaczące ograniczenia środków na inwestycje infrastrukturalne. Wprowadzacie nowe podatki, zawłaszczacie spółki Skarbu Państwa. Kiedy wreszcie zaczniecie pracować, bo na razie nieudolność goni klęskę, a klęska zapisana jest w każdym kolejnym budżecie, także w tym najnowszym, na 2021 r. Konkretne pytania: Ile państwo przeznaczycie na funkcjonowanie karetek wymazowych? Jakie środki zostały zarezerwowane na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej? Obiecaliście. Jakie środki zarezerwowano [[Dzwonek]] na utrzymanie oddziału psychiatrii dziecięcej w szpitalu w Bielsku-Białej? Jakie środki w południowej części województwa śląskiego zaplanowano na walkę ze smogiem?

Wysoka Izbo! Dlaczego subwencja oświatowa na przyszły rok jest na tak samo niskim poziomie jak tegoroczna? Zaplanowano 52 mld zł w tym roku. Patologię przyjęto za normalność. Pandemia spowodowała większe koszty po stronie szkół, których w tym roku budżetowym budżet centralny nie pokrył. Wielu samorządom brakuje na płace, wiele samorządów się zadłuża.

17 września w tej Izbie przyjęliśmy kolejną COVID-ową ustawę, która zakładała, że dźwignią z pandemii, z zapaści gospodarczej będą właśnie wydatki na transport, na łączność, na kolej. Na gospodarkę mieszkaniową - 44% mniej. Pytanie, jeśli chodzi o transport i łączność, co dla Wielkopolski.

Panie i Panowie Posłowie! Kryzys obnażył zrujnowane finanse publiczne. To najlepiej udowadnia, że nigdy nie było pieniędzy na piątkę Kaczyńskiego.

Pytałam już o to w Komisji Finansów Publicznych. Pan przewodniczący sobie zażartował, że luka VAT wynika z budżetu. Rozumiem, że można ją odczytać z budżetu, natomiast pytałam, z jakiego powodu nagle nam tak bardzo urosła. Podatek VAT spada szybciej niż PKB i to tak wygląda, jakbyście po wyborach mafii VAT-owskiej oddali pieniądze, które niby premier Morawiecki im przed wyborami zabrał. Teraz moje kluczowe pytanie, panie ministrze. W poprzedniej kadencji cała komisja pod wodzą pana posła Horały zajmowała się tym, jak to PO kradło pieniądze. Komu i ile pozwoliliście ukraść, że ta luka [[Dzwonek]] znowu urosła?

Wysoka Izbo! Od gigantycznych wydatków na wojsko, ponad 50 mld zł, nie będziemy ani zdrowsi, ani mądrzejsi, ani szczęśliwsi. Ochrona zdrowia w przyszłym budżecie stanowi zaledwie 5,39% PKB, i to czasie, kiedy mamy zapaść służby zdrowia, ludzie nie są badani, a operacje są przekładane. Służba zdrowia leży na łopatkach. Na inwestycje przeznaczacie o 10 mld mniej niż w 2020 r., a na domiar złego aż 63% to inwestycje w wojsko. Ale kupno kolejnych amerykańskich samolotów i tak nie pomoże wam w amerykańskiej ocenie waszego traktowania LGBT. Ze Szczecina i Koszalina do Warszawy od lat jedzie się 7, 8 godzin przez Rzepin i Kostrzyn. Mierzeja Wiślana to 465 mln. Ile szczepionek, oczywiście z wiarygodnego źródła, można za to kupić? Kiedy zatem skończycie z wojennymi obsesjami, a zaczniecie wydawać na nasze zdrowie, edukację, gospodarkę i kulturę? Dziękuję. Pan poseł Michał Szczerba, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Ministrze! I nie ma ważniejszej sprawy, Wysoka Izbo, dla Polek i Polaków, szczególnie w czasie pandemii, niż zdrowie. Zdrowie powinno być priorytetem państwa. I te 5,3% PKB to są wydatki na zdrowie absolutnie niewystarczające. Bardzo często jest tak, że osoby starsze, osoby z otępieniem, chore na chorobę Alzheimera, a jest ich w Polsce pół miliona, potrzebują opieki drugiej osoby. To są dorośli opiekunowie osób niepełnosprawnych. Gdzie w tym budżecie na rok 2021 jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2014? To pierwsza sprawa. Druga sprawa to rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego. Tak naprawdę państwo poprzez ustawy, które przyjmowaliście, obniżyliście dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Wysoka Izbo! Budżet państwa to również budżet lokalnych społeczności. To budżet mieszkańców Tucholi, Żnina, Bydgoszczy, Inowrocławia. To budżet ludzi, którzy często swoje problemy lokują w nadziei. Nadziei, że tutaj, w parlamencie, będziemy przyjmowali ustawy dobre i służące tej społeczności.

Dzisiaj w województwie kujawsko-pomorskim jeden z największych problemów to dofinansowanie szpitali. Szpitali, które mierzą się nie dość, że z pandemią koronawirusa, to jeszcze mają ordynarne braki w wyposażeniu, brakuje także możliwości zatrudnienia nowego personelu. Dlatego zwracam się z pytaniem do pana ministra: Jak dużo środków dla szpitali powiatowych planujecie przeznaczyć, które będą dedykowane na wyposażenie i wzrost wynagrodzeń? Druga rzecz to sprawa dotycząca edukacji widzianej oczyma rodziców i dzieci. Czego im najbardziej brakuje? Laptopów, tablic interaktywnych, ale też środków finansowych na dofinansowanie różnych inicjatyw.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie będzie dotyczyć realizacji „Programu dla Śląska” Zapewne pan minister pamięta zapowiedzi z 2019 r. - 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 62 mld zł. A moje pytanie brzmi: Czy nastąpi w końcu taki moment, może w 2021 r., że zaczną się państwo z tych zapowiedzi rozliczać, nie opowiadać niestworzone historie o środkach zaangażowanych, nie definiując tego pojęcia, ale właśnie precyzyjnie się rozliczać? Kiedy opozycja porównała wasze zapowiedzi z tym, co się dzieje w rzeczywistości, po prostu przestaliście publikować kolejne dane. Jeszcze w lipcu tego roku minister odpowiedzialny za politykę regionalną informował mnie, że sprawozdanie za cały 2019 r. jest w trakcie opracowania i zostanie udostępnione posłom, prawdopodobnie, jak mówili starożytni, ad calendas Graecas, czyli po polsku: na święty nigdy. Dodam tylko, że kosztem ponad 120 tys. zł stworzyli państwo stronę „Programu dla Śląska” Ostatni dotyczy posiedzenia rady wykonawczej tego programu. Jak pan myśli, panie ministrze, czy poseł polskiego Sejmu może zobaczyć protokół z (Dzwonek) tego posiedzenia? Nie może. Może czekać, pytać, apelować.

Chciałabym zapytać, czy zapisując w budżecie wydatki na ochronę zdrowia, uwzględnili państwo zwiększone ryzyko, które wynika i z kwestii drugiej fali pandemii, i tym samym ze wzrostu kosztów leczenia, ale także z otoczenia gospodarczego, czyli spadku wpływów przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększonych kosztów wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia, ale też z ciężaru utrzymania szpitali jednoimiennych zakaźnych. Chciałabym państwa zapytać w związku z tym, że realnie spadła liczba wydawanych zielonych kart diagnostyki leczenia onkologicznego, jaką kwotę przeznaczają państwo w budżecie na leczenie onkologiczne, na chemioterapię, na finansowanie narodowej strategii onkologicznej. Ile pieniędzy w budżecie państwa w porównaniu do roku 2020 przeznaczacie państwo na psychiatrię, także na psychiatrię dziecięcą? I chciałabym zapytać, czy w tym budżecie zrealizują w końcu państwo obietnicę wyborczą sprzed wielu lat dotyczącą realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od tego, w jakim wieku ta niepełnosprawność powstała.

Panie Ministrze!

Bo pan doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że pan firmuje i daje twarz polityce realizacji bieżących interesów (Gwar na sali, dzwonek) politycznych kosztem przyszłości kolejnych pokoleń. I to jest zbrodnia wobec państwa, wobec społeczeństwa, ale przede wszystkim wobec następnych pokoleń, naszych dzieci i wnuków.

Na tym posiedzeniu Sejmu, dzisiaj, rozmawialiśmy o dwóch kolejnych podatkach. W poprzedniej kadencji to było kilkadziesiąt nowych podatków, które zostały wprowadzone przez rządy Prawa i Sprawiedliwości.

Po trzecie, chciałbym się dowiedzieć, czy w przyszłym roku też będzie prowadzona taka polityka wobec Funduszu Sprawiedliwości, który powinien pomagać ofiarom przestępstw, a w gruncie rzeczy służy do realizacji polityki finansowania Tadeusza Rydzyka. Pani poseł Marta Golbik, klub Koalicji Obywatelskiej.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Pytam, ponieważ wszystkie dane, które spływają do nas, mówią o tym, że właśnie w trakcie pandemii ten problem jeszcze bardziej się pogłębia, mówią o tym wszyscy specjaliści i wszystkie raporty. Państwo na pewno zapoznali się szczegółowo z raportem NIK-u, który jest miażdżący dla systemu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, w którym można dowiedzieć się o tym, że na Podlasiu nie ma szpitala dziennej opieki psychiatrycznej. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, czy uwzględnili państwo taki koszt w tym budżecie, czy nastąpiła realna wycena usług za świadczenia, ponieważ niestety mamy wciąż do czynienia z odpływem specjalistów do sektora prywatnego. To powoduje, że na 400 tys. dzieci - bo tak szacuje się dziś zapotrzebowanie na usługi specjalistów - mamy zaledwie 416 psychiatrów.

Wysoka Izbo! W grudniu 2017 r. premier Morawiecki szumnie ogłosił i przedstawił „Program dla Śląska” Przedstawił ten program jako strategiczny program, którego realizacja ma doprowadzić do zmiany profilu gospodarczego Śląska.

Chcecie likwidować dalej huty. Panie Ministrze! Jakie wsparcie finansowe otrzyma sześć miast w województwie śląskim, które - jak zaznaczyliście w tym programie - tracą funkcję społeczną i gospodarczą, a wśród nich są m.in. Jastrzębie-Zdrój i Rydułtowy? 9 stycznia br. tu, w Wysokiej Izbie, dyskutowaliśmy o obywatelskim projekcie ustawy przyznającej dodatek do emerytur dla wieloletnich członków ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie kluby parlamentarne były za. Mało tego, prezydent Duda podczas kampanii wyraźnie obiecał wsparcie dla tego projektu. Pan poseł Artur Łącki, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy rząd wprowadzał swoje tarcze antykryzysowe, dziurawe tarcze antykryzysowe, zastanawiałem się, kiedy przyjdzie miecz podatkowy, bo jak jest tarcza, to i miecz. Nie minęły 2 miesiące i jest. Dzisiejszy dzień zostanie zapisany w historii mikro- i małych polskich przedsiębiorstw jako czarna środa. Po pierwsze, CIT estoński, a właściwie polskie wariacje na temat CIT-u estońskiego. Po drugie, koniec spółek komandytowych, czytaj: upadek kilkudziesięciu tysięcy polskich mikro- i małych firm. Zwracam się do marynarzy, którzy wszyscy korzystają z ulgi abolicyjnej, bo ponad 180 dni w roku pracują poza granicami kraju: już nie będziecie jej mieli, będziecie dwa razy płacić podatki. No i ustawa budżetowa - raczej rozmontowywanie reguł finansowych, kreatywna księgowość i propaganda. Moje pytanie jest takie: Ile w tej ustawie budżetowej, panie ministrze, zapisaliście środków na zakup ewentualnych szczepionek na COVID-19, które się pojawią w roku 2021?

Drugie pytanie dotyczy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym się po raz kolejny upomnieć o Polskę wschodnią.

Ale chodzi również o to, by kraj był rozwijany w sposób zrównoważony. To jest pierwszy element.

Daję też pod rozwagę, jeśli mówimy o rozwoju Polski wschodniej, budowę nowego przejścia granicznego Zbereże - Adamczuki. Od dłuższego czasu o tym mówimy, ale niestety kończy się tylko i wyłącznie na mówieniu. Kolejny element to rzecz niezwykle ważna. Chełm jest jednym z nielicznych dużych miast, które wciąż nie ma obwodnicy. Wierzę głęboko w to, że środków finansowych na ten cel nie zabraknie, ale również apeluję o zwiększenie środków na drogi samorządowe. Pan poseł Michał Krawczyk, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Budżet, projekt budżetu państwa to nie tylko spis cyferek, to nie tylko spis wydatków i przychodów na kilkaset miliardów złotych.

Czy poprawicie funkcjonowanie oddziałów położniczych, o których NIK w swoim raporcie pisze: nie zapewniają pacjentkom i noworodkom wymaganej jakości świadczeń medycznych?

Czy dzięki temu budżetowi w szkołach przybędzie lepiej wyposażonych klas? A może przybędzie żłobków? Ale nie tych prywatnych. Państwo w raportach lubicie mówić o tym, że w Polsce przybywa żłobków. Chodzi o to, czy przybędzie żłobków państwowych, publicznych, takich, na które Polki i Polaków będzie stać. I jeszcze chciałem zapytać o jedną kwestię, o drogę wodną E40. Jaka jest kwota przeznaczona na budowę tej inwestycji, która zdegraduje ekologicznie Lubelszczyznę, a której dokumentację (Dzwonek) skrzętnie państwo ukrywacie? Pani poseł Krystyna Skowrońska, klub Koalicja Obywatelska.

Czy pan minister wie? Czy pan marszałek wie?

To jest wsparcie na zdrowie z budżetu państwa. A ile na obsługę długu? Panie ministrze, czy pan pamięta?

I dzisiaj są zamykane szpitale. Państwo powinni wiedzieć, ile szpitali jest zamkniętych i jakie mają długi. Przecież minął wrzesień i samorządy musiały zapłacić za długi swoich szpitali, których są organami założycielskimi. A przecież jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2019 r., który mówi, że za finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiada Skarb Państwa.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Deficyt w tym roku wyniesie niemal 110 mld zł, a w przyszłym - ponad 82 mld zł. Tempo wzrostu zadłużenia Polski macie istnie szokujące. Ogólnie rzecz biorąc, aż połowa zadłużenia naszego kraju jest to dzieło rządów PiS. Przez ostatnie 5 lat nie przygotowaliście Polski na kryzys, a roztrwoniliście wypracowane przez Polaków pieniądze na populizm, na propagandę, na zarobki swoich ludzi obsadzanych w spółkach Skarbu Państwa. Nie wspomnę już o 70 mln zł, które minister Sasin wydał na wybory, które się nie odbyły. Mimo deficytu teraz brakuje pieniędzy na wszystko. Nie będzie podwyżek w budżetówce, co faktycznie oznacza spadek zarobków, bo jest inflacja i wzrost kosztów utrzymania. Brakuje środków na przeciwdziałanie COVID, brakuje na ratowanie gospodarki, na służbę zdrowia, na zapobieganie innym katastrofom, takim jak powódź. No i nic dziwnego, że brakuje pieniędzy, skoro w czasach koniunktury nie stosowaliście się do stabilizacyjnej reguły wydatkowej i roztrwanialiście pieniądze zarobione przez Polaków. Teraz nagle, gdy jest kryzys, twierdzicie, że będziecie się stosować do tej reguły, więc znów wydajecie pieniądze. Pytam: Kto za to wszystko będzie płacił? Jakie kroki - poza optymalizacją księgową oraz nakładaniem dodatkowych podatków, co dzisiaj próbujecie uczynić, na firmy - zamierzacie poczynić celem ratowania budżetu i podupadającej gospodarki? Pani poseł Hanna Gill-Piątek, poseł niezależna. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam tutaj dwie ustawy, nad którymi pracujemy obecnie w Sejmie. Tę ustawę, ustawę mieszkaniową, akurat zdjęliśmy dzisiaj z porządku obrad, ale pewnie uchwalimy ją w tym roku, ponieważ jest to ustawa, która nie budzi wątpliwości, ona zawiera dobre rozwiązania i w Komisji Infrastruktury właściwie dostała jednogłośne poparcie. I ta ustawa nie widzi się zupełnie z drugą ustawą, którą tutaj trzymam, nad którą dzisiaj właśnie w tym miejscu debatujemy, ponieważ w tej ustawie, ustawie mieszkaniowej, zapisane jest, że do 2020 r. na fundusz rozwoju mieszkalnictwa będzie zapewnione 1,5 mld, a do Funduszu Dopłat rocznie ta ustawa przewiduje dołożenie 1 mld zł, czyli mamy 2,5 mld na mieszkalnictwo rocznie, natomiast tutaj tego nie ma. Ja sprawdzałam. Naprawdę. Największe, co jest, największa kwota, która jest w ustawie budżetowej, to jest rezerwa 300 mln. I nikt nie potrafi mi tego wytłumaczyć. A więc chciałam zapytać - w związku z tym, że mieszkalnictwo jest dziedziną bardzo u nas zaniedbaną, która naprawdę wymaga dużych pieniędzy, a jednocześnie są to inwestycje małe, lokalne, mogące zostawić pieniądze na miejscu, pobudzić lokalne firmy budowlane - dlaczego nie ma w tym budżecie pieniędzy na mieszkalnictwo, natomiast są na takie pomniki władzy, na takie gigantomańskie inwestycje, jak np. przekop Mierzei Wiślanej albo też następne prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym. I bardzo proszę o udzielenie mi tej odpowiedzi na piśmie. Pan poseł Dariusz Joński, klub Koalicji Obywatelskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

3 miesiące po tym dziś mamy 3003 nowe przypadki koronawirusa i 75 osób, które zmarło. Bo dzisiaj to pan minister Kościński mówi tak: o tej porze za rok będziemy już po recesji. Już zakopaliśmy wszystkie skutki, a większość krajów Unii Europejskiej będzie jeszcze pewnie 2–3% do tyłu. Chciałbym zapytać pana ministra, u której wróżki pan był. Bo jeśli tak, to państwa seanse uspokajania po prostu nie działają. To, co państwo robicie, to nonszalancja w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, chociażby jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. Teraz pan wychodzi na tego, który mówi i uspokaja, że wszystko będzie w porządku, tylko nie mówi pan, na jakich danych i wskaźnikach pan się opiera. Więc apeluję do państwa, żebyście nie uprawiali fikcji, nie uprawiali PR-u tylko i wyłącznie, tylko mówili, jaki jest stan faktyczny. Teraz głos ma minister finansów, funduszy i polityki regionalnej pan minister Tadeusz Kościński.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawda o stanie finansów jest taka, że na koniec września mieliśmy ponad 120 mld na rachunkach budżetu państwa. Mamy ponad 98% naszych potrzeb pożyczkowych już wykonane. Recesja w Polsce - my jako Ministerstwo Finansów prognozujemy, czy będzie to 4,6, zgodnie z tym, co Komisja Europejska tak samo prognozuje. Również dane z Komisji Europejskiej, z Banku Światowego: Polska będzie miała najniższą recesję ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy jedynym krajem, który będzie miał poniżej 5%, a średnia jest ok. 9%. Również Polska wyjdzie z tej recesji najszybciej pewnie ze wszystkich krajów. To są dane, które pochodzą z Komisji Europejskiej, z Banku Światowego. Przypominam, że 11 września międzynarodowa agencja Moody’s podtrzymała rating dla Polski z perspektywą na poziomie stabilnym, co znaczy, że finanse publiczne są dobrze zarządzane w Polsce.

2 października, w ostatnim tygodniu, Standard & Poor’s, ostatnia z tych dużych trzech, również podtrzymała perspektywę Polski na poziomie stabilnym.

I ponownie potwierdzam, że nie ma żadnych prac w Ministerstwie Finansów nad zwiększeniem żadnych podatków. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zamykam dyskusję. Zgodnie z art. 106 regulaminu Sejmu projekt ustawy budżetowej Sejm kieruje do rozpatrzenia do Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne części projektu rozpatrują także właściwe komisje sejmowe, które przekazują Komisji Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 641) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Sebastiana Skuzę o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wraz z projektem ustawy budżetowej Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Główne rozwiązania zawarte w omawianym projekcie dotyczą mrożenia wynagrodzeń w budżecie państwa na 2021 r. W państwowych jednostkach budżetowych, w tym w ministerstwach i urzędach, przewiduje się, co do zasady, utrzymanie wynagrodzeń na poziomie roku obecnego. W związku z tym w projekcie ustawy okołobudżetowej na rok 2021 zawarto przepisy zamrażające wynagrodzenia w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych oraz organach, o których mowa w art. 139 ustawy o finansach publicznych, tj. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunale Konstytucyjnym, Najwyższej Izbie Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy i Instytucie Pamięci Narodowej. Ponadto, mając na względzie zasadę sprawiedliwości społecznej, proponuje się utrzymanie na poziomie roku 2020 m.in. wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, w tym w stanie spoczynku, oraz maksymalnych wynagrodzeń osób wymienionych w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz osób zatrudnionych w podmiotach podlegających pod przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W projekcie zawarte są też regulacje, które zmieniają zasady dotyczące nagród o charakterze uznaniowym. W roku 2021 proponuje się w miejsce planowanego, tworzonego funduszu nagród wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych utrzymanie możliwości przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowanie wyłącznie ze środków na wynagrodzenia, które nie zostały wydatkowane z przyczyn obiektywnych, jak np. pozostawanie na zwolnieniach, urlopach wychowawczych, czy też z wakatów. Działania te przyczynią się do ograniczenia wzrostu wydatków budżetu państwa. Przewiduje się również utrzymanie podstawy naliczenia funduszy socjalnych na poziomie analogicznym do tego z roku bieżącego, poziomie podstawy naliczenia z roku 2018, i te rozwiązania dotyczyłyby nauczycieli, emerytów i rencistów żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin, jak również pracowników cywilnych, w odniesieniu do naliczenia których jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kolejnym elementem proponowanej ustawy okołobudżetowej jest umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. Chciałem tu tylko wskazać, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w tym samym roku, czyli w 2019 r., dokonał wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej, tak że te środki zostały uzupełnione.

Działania te umożliwią kontynuację programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” W projekcie zawarto również przepis umożliwiający umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze przedstawione przepisy, zwracam się do Wysokiej Izby o uchwalenie proponowanych rozwiązań. Dziękuję. Bardzo dziękuje, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Henryk Kowalczyk w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, druk nr 641. Oczywiście zasady zapisane w tej ustawie, a więc m.in. zamrożenie wynagrodzeń, czy zamrożenie naliczania funduszu socjalnego odnoszące się do roku 2018 są naturalną konsekwencją sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Można wspomnieć o uproszczeniu procedury wypłat ekwiwalentu z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pani poseł Marta Golbik. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! Ustawa przewiduje zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, samorządowych, komunalnych. Zaproponowane przez rząd zmiany będą miały wpływ m.in. na wysokość wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych, na wysokość uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Zamrożeniu będą też podlegały diety członków Krajowej Rady Sądownictwa i ławników biorących udział w rozpoznaniu. Warto też powiedzieć o liczbach, bo konsekwencje zamrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniesie ok. 13 354 nauczycieli szkół rządowych i 527 196 nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponad 3 mln pracowników sektora publicznego i ponad 6,5 mln pracowników sektora prywatnego poniesie konsekwencje zamrożenia podstawy odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych na poziomie z 2018 r. Konsekwencje poniosą również służby mundurowe, emeryci służb mundurowych i członkowie ich rodzin. To ponad 411 tys. osób. Można by się spodziewać, że ograniczenia budżetowe będą dotyczyły wszystkich zbędnych wydatków państwa. Tymczasem w tym samym projekcie ustawy znajdujemy zapis o środkach budżetowych dla szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeznaczonych na remonty w nieruchomościach, np. wykonanie węzła komunikacyjnego w budynku Perkoz na terenie ośrodka wypoczynkowego Łańsk albo modernizację wnętrz lobby recepcyjnego w budynku głównym Puszcza w ośrodku wypoczynkowym Łańsk. Szanowni Państwo! Pieniądze, 57 mld, idą na przeróżne cele.

Dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! Szkoda, że pan minister finansów nas opuścił, bo chciałam go zapytać, czy jest tak dobrze, że wszyscy nas chwalą, jak uważa i tu stwierdzał, czy jest tak źle, że trzeba mrozić wszystkie pensje w budżetówce, o czym mówiła przed chwilą moja koleżanka. No bo skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Prawda jest taka, że faktycznie dług publiczny rośnie lawinowo, szybciej niż rósł kiedykolwiek wcześniej. Tak jak nasi rodzice spłacali długi Gierka, tak my będziemy spłacać długi Kaczyńskiego i Morawieckiego, i całego PiS-u. W trakcie debaty budżetowej mówiłam o tym, że w ogóle poza finansami publicznymi zrujnowaliście również system ubezpieczeń społecznych i przy okazji - jest jeszcze trochę czasu na dyskusję, którą i tak zawęziliście do minimum - parę słów o tym. A więc z budżetu tegorocznego wydamy na renty i emerytury dodatkowo, poza tym, co obsługują ZUS, KRUS i inne dedykowane temu jednostki, 126 mld zł.

Bo nie ma na to pieniędzy i tak jak powiedziałam wcześniej, pochodzą one z długu, co jest na koszt przyszłych pokoleń. Solidarnie byłoby myśleć o emerytach i rencistach nie tylko dziś, ale również za parę lat, kiedy przestaniecie rządzić, bo wtedy również ZUS musi być wypłacalny.

Dziękuję bardzo.

Pan poseł Dariusz Wieczorek w imieniu klubu parlamentarnego Lewica. Proszę bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście to dobrze, że temperatura tutaj jest jakaś taka w miarę ludzka, ponieważ jak słyszę o tym zamrażaniu, to aż ciarki przechodzą, bo widzę, że teraz słowo „zamrażanie” będzie bardzo charakterystyczne dla polskiego rządu i dla ministra finansów. Jest tylko pytanie czy w sytuacji, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, jest to najlepsza polityka, jaką powinniśmy przyjąć. Jest pytanie, czy właśnie w momencie kiedy jest problem, jeżeli chodzi o recesję gospodarczą, nie powinniśmy napędzać gospodarki poprzez właśnie zlecenia dotyczące budowy infrastruktury, budowy dróg, budowy kolei, czy nie powinniśmy również odpuścić tego zamrażania, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w sferze budżetowej, bo przecież to napędza konsumpcję, napędza koniunkturę, przecież to są podatki, to są odpisy na ZUS, to jest cały mechanizm gospodarki, który w takim momencie powinien zafunkcjonować, a wiele jest przykładów krajów, które były w takiej dużej recesji, kiedy rzeczywiście te publiczne inwestycje ratowały i pomagały wyjść z tej recesji. Oczywiście ten projekt ustawy wprost jest związany z projektem budżetu, który przedstawiliście państwo, ten projekt budżetu na rok 2021, w związku z tym on wprost, mówiąc krótko, uznaje te wszystkie, w naszej ocenie błędne, zapisy, które w tym budżecie się pojawiły. Mówiliśmy tutaj o inwestycjach, zobaczmy więc: w tej ustawie jest „Program modernizacji Służby Więziennej lata 2017-2020”, „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020”, natomiast nie ma już kontynuacji tych programów, a to są setki milionów zł na inwestycje właśnie w powiatach, właśnie w gminach. A więc tego nie realizujecie.

No bo przecież tą ustawą umarzacie pożyczkę dla Wód Polskich, czyli, mówiąc krótko, kolejne 780 mln pojawia się jako umorzenie tej pożyczki. Jeżeli chodzi o umorzenie i mechanizm umarzania w tej chwili pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej - o tym mówiłem w pierwszej części i nie chcę już tego powtarzać - to jest dokładnie ten sam mechanizm, który za chwilę wystąpi, czyli zakładany deficyt w Funduszu Solidarnościowym. Kompletnie niezrozumiałe jest zamrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

No co to jest za wpis „nie mniej niż” Rozumiem, że dzisiaj są inne potrzeby, widzimy, co się dzieje, widzimy jakie są kłopoty.

Przecież są inne potrzeby. Nagle traktujemy to jako wielką świętość. Nie dość, że zamrażacie wynagrodzenia w sferze budżetowej, to likwidujecie te wszystkie fundusze nagród, które, mówiąc krótko, też są mechanizmem, jeżeli chodzi o pracodawców, do kreowania polityki kadrowej. Dlatego jeszcze raz apeluję o to, ażeby przeanalizować przede wszystkim budżet, bo z tego będzie wynikał ostateczny kształt tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska chciałbym przedstawić nasze stanowisko dotyczące projektu ustawy okołobudżetowej.

Tylko tak się zastanawiam, panowie ministrowie, czy ci wykonujący zawody mieszczące się w tej kategorii, którym zamrażacie wynagrodzenia, jak lekarze, jak pielęgniarki, jak ratownicy medyczni, jak cały sztab osób pracujących w diagnostyce, są dzisiaj dobrymi adresatami zamrażania wynagrodzeń? To są dzisiaj, w tych wyjątkowych realiach, te zawody, ci pracownicy, którzy naprawdę zasługują na to, żeby poziom ich wynagrodzeń był dopasowany, po pierwsze, do wysiłku, który na co dzień podejmują, po drugie, do skali zagrożenia i do perspektyw, które nie są, wszyscy się zgodzimy, najlepsze, chodzi nie tyle o tygodnie, co nawet miesiące czy lata. To jest pierwsze nasze zastrzeżenie i chciałbym to w imieniu klubu Koalicji Polskiej bardzo jasno zasygnalizować.

Łóżka są ważne, karetki są ważne, ale jak nie będzie ludzi należycie wynagradzanych za wysiłek, to tylko przyspieszy erozję tego systemu. Druga sprawa również na pozór wydaje się racjonalna, czyli podniesienie limitu wydatków dotyczących realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zakupu szczepionek, pojawia się, jeśli chodzi o program szczepień ochronnych. Panie Ministrze!

Ja trochę i swój okręg wyborczy, i region, z którego pochodzę, jakim jest Wielkopolska, zjeździłem, troszkę się z samorządami, z rolnikami naspotykałem w ostatnim czasie, kiedy jeszcze było można, a już w najlepsze Wody Polskie funkcjonowały. Muszę powiedzieć, że nie znalazłem ani jednego przykładu na to, że Wody Polskie, już nie mówię, że zrealizowały, ale nawet podjęły najmniejszy wysiłek, żeby przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi.

Pani marszałek, kończę, jeszcze tylko ostatnie zdanie. Klub Parlamentarny Koalicja Polska nie widzi możliwości poparcia tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. W związku z tym pan poseł Grzegorz Braun w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja. Przechodzimy do pytań. Zamykam listę osób chcących zadać pytanie. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Nie ma pana posła. Pan poseł Marek Rutka, Lewica. Nie ma pana posła. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie ma. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Co ta ustawa wnosi? Po pierwsze, pozwala na wyprowadzenie środków z funduszu CEPiK, czyli tych środków, które przy każdym badaniu technicznym wpłacają kierowy. Po drugie, w ustawie znajdziemy również takie prawne podstawy do oszustwa związanego z przeznaczeniem 2% PKB na obronność. Czytamy, że do tych wydatków PiS zaliczy wydatki na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe czy na kształcenie cywili na uczelniach. To wielkie oszustwo, jeżeli chodzi o zdolności obronne w Polsce. PiS uderza także w urzędników, bo likwidacja funduszu nagród za wybitne osiągnięcia jest de facto pochwałą przeciętności.

Dziwię się, że rząd przedłożył takie skandaliczne projekty budżetowe, [[Dzwonek]] bo można je opisać tak: zero wizji, zero rozwoju, zero odpowiedzialności. My tych ustaw budżetowych nie poprzemy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! W ostatnich latach rząd nie liczył się z pieniędzmi publicznymi, wręcz odwrotnie, był bardzo rozrzutny. Teraz, kiedy przyszedł trudny czas, kto najbardziej ucierpi? Oczywiście sfera budżetowa, pracownicy sfery budżetowej, którzy nigdy dobrze nie zarabiali, bo następuje zamrożenie wynagrodzeń na poziomie tego roku, zamrożenie podstawy naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych czy też rezygnacja z tworzenia oddzielnego funduszu nagród. A w takich służbach jak Służba Celno-Skarbowa czy Policja oraz inne służby nagrody zawsze były i powinny być. Przecież praca organów celno-skarbowych w dużym stopniu jest nagradzana, co zachęca do aktywności, do efektywności. Niestety tworzy się, jak kolega powiedział, taką filozofię jak pochwała przeciętności. Pytam się, jakie będą skutki takich niesprawiedliwych działań wobec pracowników sfery budżetowej, takich decyzji, które są bardzo krzywdzące, które nie powinny mieć miejsca, bo tu są takie służby, które są nisko wynagradzane. To jest [[Dzwonek]] wielki błąd, proszę państwa. Dziękuję bardzo, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Odniosę się do innego artykułu, bo moim zdaniem ten ośrodek w Łańsku to jest tylko przykrywka dla dużo większego skandalu, który jest w tej ustawie. Otóż chodzi o art. 73, w którym czytamy o umorzeniu długu Funduszu Solidarnościowego wobec Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Szanowni Państwo! Polityka musi być na pokolenia, a nie na kadencje. Jednocześnie informuję, że złamała pani zalecenia Prezydium i Konwentu Seniorów co do obecności na sali posiedzeń. Prosiłabym, żeby to się nie powtarzało. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Wiceministrze! Panie Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, który z PiS-u jesteś sam na tej sali! Chciałam się pana ministra zapytać: Zaczęliście od siebie? Czy zaczęliście od siebie, od waszych wynagrodzeń, od organizacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od oszczędności? Zaczynacie państwo i mówicie: 10,5 mln osób będzie dotknięte np. mrożeniem funduszu świadczeń socjalnych, ale państwo u siebie oszczędności przy rekonstrukcji rządu nie robicie żadnej, bo podobno z 20 resortów będzie 14 i dodatkowo inne jeszcze urzędy. I skandalem jest, tak jak m.in. mówił kolega [[Dzwonek]] z Koalicji Polskiej, że dotyczyć to będzie również pracowników ochrony zdrowia. W okresie pandemii? Bardzo proszę. Panie Ministrze!

Urzędnicy powinni być dobrze wynagradzani, żeby pełnić odpowiedzialnie swoje funkcje, odpowiedzialnie podejmować decyzje, żeby ludzie kompetentni, chcący pracować, zaangażowani pracowali nie dla idei, ale dlatego, że muszą utrzymać z czegoś swoje rodziny i siebie. A więc proszę mi wyjaśnić, dlaczego 2 mld idą na telewizję publiczną kosztem zamrożenia płac w budżetówce. Z drugiej strony piszecie państwo w ustawie budżetowej bardzo optymistycznie: przyspieszone tempo spożycia prywatnego popytu krajowego, ale planujecie zamrożenia w administracji publicznej i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ta ustawa jest smutnym podsumowaniem bieżącego posiedzenia i w zasadzie całego roku waszej kadencji, bo dzisiaj mieliśmy podniesienie podatków, przeregulowanie gospodarki, a na koniec dyskusję o budżecie, wyjątkowo zadłużonym budżecie, przy jednoczesnym bardzo optymistycznym przedstawianiu tego przez ministra finansów. A ta ustawa pokazuje, że jesteśmy w bardzo głębokim kryzysie, więc wasze dobre samopoczucie pokazujące, jak to właśnie wychodzimy z tego kryzysu, jest po prostu ściemą.

Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać, dlaczego pomimo obietnic w budżecie na rok 2021 nie przewidziano ani złotówki na podniesienie uposażenia nauczycieli. Rząd bez problemu znalazł środki na wypłatę wynagrodzeń dla górników, którzy mają je otrzymać za niechodzenie do pracy, tymczasem deklaracje wygłoszone dla nauczycieli mają się nijak. Każda złotówka wydana na oświatę owocuje większą świadomością i wiedzą społeczeństwa. Niedługo obchodzić będziemy dzień komisji edukacji, święto polskich nauczycieli. Zapewne odbędą się uroczystości. Wtedy kiedy będą pytali państwa, posłów PiS-u, jak zachowaliście się wobec nauczycieli, wobec podwyżki dla nauczycieli, to niech pan poseł mówi szczerze, że Lewica apelowała, abyście jednak zrewidowali swój pogląd w tej (Dzwonek) sprawie. Dziękuję, panie pośle. Ostatnie pytanie, pan poseł Marek Rutka, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czy rząd pod nazwą szczególnych rozwiązań służących realizacji ustawy budżetowej ma zamiar wprowadzić podobne rozwiązania, tak jak było to w przypadku tarczy antykryzysowej, która umożliwia budowę osiedli mieszkaniowych na terenach wcześniej wyłączonych z budowy, tak jak ma to miejsce nad morzem, w Mechelinkach koło Gdyni, gdzie na terenie zalewowym powstaje luksusowe osiedle. W związku z projektowanym w 2021 r. zamrożeniem na poziomie bieżącego roku wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych proponuje się dodanie dodatkowego przepisu - jest to art. 10 - uniemożliwiającego zwiększenie wynagrodzeń w trakcie roku 2021. Kiedy jednym z najważniejszych czynników wzrostu dochodów państwa ma być konsumpcja, po raz kolejny wprowadza się zamrożenie wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania pań i panów posłów odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o pytanie dotyczące przeznaczenia 0,2% na obronność, to te rozwiązania mają raczej charakter systemowy niż finansowy z tego względu, że zaliczane są tam niewielkie wydatki, takie jak wydatki agencji wojskowych, uczelni wojskowych i pogotowia lotniczego, które jest wykorzystywane również przez służby wojskowe. Sfera budżetowa w roku bieżącym otrzymała 6-procentowe podwyżki. Podobnie podwyżki otrzymali nauczyciele, i tu są zapewnione skutki przechodzące na rok następny. Tak jak mówiłem, prezentując projekt ustawy okołobudżetowej, nagrody będą mogły być przyznawane, ale nie poprzez tworzenie z funduszu wynagrodzeń dodatkowego funduszu, tylko z naturalnie powstałych oszczędności, takich jak np. oszczędności etatowe. Zwracam uwagę, że ustawa okołobudżetowa na rok bieżący zawierała takie zapisy. Niezbędne jest dla instytucji gospodarki budżetowej stworzenie materialnej podstawy prawnej, żeby mogła otrzymywać dotacje, i taka podstawa była w tym roku. Jako że ze względu na sytuację pandemiczną nie udało się tej inwestycji zrealizować, przechodziłaby ona na rok następny.

O rzetelnej sytuacji państwa dotyczącej ustawy budżetowej rozmawialiśmy przy omawianiu ustawy budżetowej na rok 2020, na rok 2021. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań, czyli o godz. 20. Do tego czasu ogłaszam przerwę.

Wznawiam obrady. Przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał. że Sejm propozycję przyjął. Czy słyszałem sprzeciw? Proszę? Dziękuję bardzo. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, - o Funduszu Medycznym. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 666 i 669. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin (druki nr 611 i 658) Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Jarosława Rzepę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pozwólcie państwo. Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac nad poselskim projektem uchwały w sprawie upamiętnienia Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę jego urodzin. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 22a ust. 2 i ust. 4 pkt 4 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierowała w dniu 16 września 2020 r. projekt uchwały zawarty w druku nr 611 do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 6 października wnosi do Wysokiego Sejmu o przyjęcie tej uchwały. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować posłowi wnioskodawcy Pawłowi Szramce za przygotowanie projektu, a całej Komisji Kultury i Środków Przekazu - za merytoryczną pracę nad projektem i wniesione poprawki. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin. 12 września 1820 roku w majątku Mileszewy w powiecie brodnickim urodził się Ignacy Łyskowski - wybitny działacz społeczny, polski poseł, pozytywista. W 1848 roku został delegatem powiatów brodnickiego oraz lubawskiego do Frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie nad Menem. Był zaangażowany w rozwój działalności Ligi Polskiej na Pomorzu. W 1861 roku przyczynił się do powstania Towarzystwa Agronomicznego Ziemi Michałowskiej, którego działalność polegała na zakładaniu biblioteczek ludowych oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zmiany sposobu uprawy roli, tj. przechodzenia z trójpolówki na płodozmian. W 1867 roku, razem z Teodorem Donimirskim i Hiacyntem Jackowskim, zwołał w Toruniu pierwsze posiedzenie sejmiku gospodarczego Polaków z Prus Zachodnich. W celu krzewienia oświaty, ochrony języka polskiego oraz podnoszenia fachowej wiedzy rolników i rzemieślników w 1869 roku, wraz z Ludwikiem Ślaskim i Leonem Czarlińskim, powołał Towarzystwo Moralnych Interesów Ludności Polskiej pod Panowaniem Pruskim. W 1875 roku został pierwszym prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Przez blisko 20 lat swojej kariery na tym szczeblu był uważany za jednego z najlepszych mówców i najbardziej wytrawnych polskich parlamentarzystów. Przez długie lata sprawował funkcję prezesa Koła Polskiego. Pełniąc funkcję posła, stanowczo występował przeciwko germanizacji w szkolnictwie, sądownictwie i administracji, domagając się równouprawnienia w odniesieniu do języka polskiego. Jako poseł powiatu brodnickiego aktywnie przyczynił się do powstania gimnazjum w Brodnicy z prawem fakultatywnego nauczania języka polskiego. W uznaniu wielkich zasług Ignacego Łyskowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje mu cześć w przypadającą w tym roku 200. rocznicę jego urodzin i wyraża głęboką nadzieję, że jego życie i działalność staną się godnym do naśladowania wzorem” Dziękuję panu posłowi. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy wobec tego do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 658, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 636-A. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Skierowano ten projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Bardzo dziękuję panu posłowi. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 636. Komisja przedstawia również wniosek mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. W 1. poprawce do części tekstowej projektu ustawy wnioskodawcy proponują w załączniku nr 10 do ustawy „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym” dodanie lit. j. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 4 mld zł. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki w pozycji 5: Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki o kwotę 10 mln zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej. Przystępujemy do głosowania.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki o kwotę 10 mln zł na realizację zadań ustawowych w zakresie rozpoznawania zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisji wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. We wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują zmianę w części 83: Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 13. poprawce wnioskodawcy proponują zmianę w części 83: Rezerwy celowe w pozycji 56: Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 363, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 451 posłów. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 598-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Witolda Czarneckiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrywała 16 poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania ustawy o doręczeniach elektronicznych. 15 poprawek zgłosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, jedną poprawkę Koalicja Obywatelska. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 598. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 450 posłów. Sejm wnioski odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 442, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 9. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. W 8. poprawce wnioskodawcy proponują inne brzmienie art. 124. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 439, przeciw - 1, wstrzymało się 9. Sejm poprawkę przyjął. W 10. poprawce wnioskodawcy proponują nadać inne brzmienie art. 143. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 436, nikt nie był przeciw, 9 posłów się wstrzymało. Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Z poprawką tą łączą się poprawki 13. i 15. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 442, nikt nie był przeciw, 9 się wstrzymało. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 598, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych. Panie i Panowie Posłowie! Państwo Ministrowie!

Czy naprawdę nowy rząd - bo my nie - chce to nałożyć, czyli zlikwidować abolicję dla pracujących za granicą? Jak państwo spróbujecie zachęcić Polaków pracujących za granicą, żeby wrócili do kraju i tutaj pracowali? Przecież państwo mówili: nie wyjeżdżajcie, pan premier mówił: nie wyjeżdżajcie, a robicie rzecz odwrotną. Tak jak wycofaliście się z projektu dotyczącego bezkarności urzędników, wycofajcie się z tego projektu. To jest najwyższy czas, żeby o tym rozmawiać. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 642, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 641, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druki nr 653 i 666) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senat zgłosił 20 poprawek. Komisja rekomenduje 6 poprawek odrzucić, 14 poprawek przyjąć.

Dziękuję, panie pośle. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. W 1. poprawce do art. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej Senat proponuje uchylić ust. 5 w art. 37m ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Z poprawką tą łączą się poprawki 14. i 19. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Senat uchwalił do art. 16 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 16. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym (druki nr 656 i 669) Proszę pana posła Tomasza Latosa o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym. Senat zgłosił 37 poprawek, z których część komisja rekomendowała przyjąć, a część - odrzucić. Dziękuję panu posłowi. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął.

Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Kto jest przeciw?

Sejm poprawki przyjął.

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 7. i 13., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 9. i 14., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 16. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Senat zgłosił do art. 35 ustawy zawierającego zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 17. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Senat proponuje, aby świadczenia opieki zdrowotnej udzielane poza granicami kraju przysługiwały świadczeniobiorcom. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 19. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Senat zgłosił do art. 37 ustawy zawierającego zmiany do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 22. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 24. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 27. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Z poprawką tą łączy się poprawka 33.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 30. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 34. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 35. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 1, przeciw - 443, wstrzymał się 1. Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 36. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym.

Wznawiam obrady. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 18. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy jeszcze ktoś z pań i panów posłów pragnie wygłosić oświadczenie? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwszy oświadczenie wygłosi pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie ma pana posła. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ogromnie się cieszę, że na sali jest pan premier, albowiem moje oświadczenie będę kierował do pana premiera. Jestem posłem z Bydgoszczy, z Kujaw i Pomorza i codziennie jestem pytany przez wyborców, kiedy znajdą się obiecane przez rząd szczepionki na grypę i kiedy znajdą się one w polskich aptekach i hurtowniach. Pytają o to osoby, które szczepiły się regularnie w ostatnich latach, pytają rodzice, a przede wszystkim pytają seniorzy, dla których szczepionka miała być za darmo, [[Oklaski]] pytają też samorządowcy i pracodawcy, którzy chcieli nieodpłatnie zaszczepić chętnych nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia i innych grup podwyższonego ryzyka. Szanowny Panie Premierze! Wszyscy oni dostają w aptekach i hurtowniach taką samą informację: szczepionek na grypę było kilka na aptekę i teraz nie wiadomo, kiedy będą i czy w ogóle będą. A wszystko to dzieje się w czasie wielkiego przyrostu zarażeń, liczby zgonów zarażonych pacjentów. Dzisiaj formalnie wykryto ponad 3 tys. zakażeń w Polsce. W niektórych województwach już ok. 80% respiratorów jest zajętych przez chorych. Wojewoda kujawsko-pomorski w dniu dzisiejszym ogłosił, że w województwie kujawsko-pomorskim zajętych jest 21 z 25 respiratorów. Zatem lekarze już niedługo będą stawali przed wyborem, komu przydzielić taki respirator. Szanowny Panie Premierze! Polski system opieki zdrowotnej nie udźwignie dwóch epidemii - grypy i COVID. Rząd wiedział o tym już od marca. Wyborcy chcą, bym zapytał pana premiera i ministra zdrowia: Gdzie są szczepionki na grypę? Razem z respiratorami w rządowych magazynach czy może w narciarskiej szopie handlarza? A może po prostu ich nie ma i nie będzie dla wszystkich, bo minister Szumowski, popularnie mówiąc, zawalił sprawę i pojechał na wczasy. A jeżeli nie będzie szczepionek dla wszystkich, to kto je dostanie? Tylko młodsi czy tylko starsi, czy ci ze skierowaniami i ze skierowaniami od kogo? Wczoraj pan minister zdrowia szumnie ogłosił w mediach politykę zero tolerancji dla Polek i Polaków. A ja się pytam: Kiedy minister zdrowia rozpocznie politykę zero tolerancji wobec samego siebie i swoich urzędników? Pytam się: Kiedy będzie zero tolerancji dla kłamiących, że radzą sobie najlepiej na świecie z epidemią i ta epidemia jest w odwrocie i pod kontrolą? Pytam się wreszcie, to pytanie trzecie: Kiedy będzie zero tolerancji dla tych, którzy zlekceważyli zakup szczepionek na grypę i zmarnowali publiczne pieniądze w dziwnych, prywatnych interesach przy zakupie maseczek i respiratorów? Te odpowiedzi pan premier i pan minister winni są Polkom i Polakom. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Dzisiaj na terenie całego kraju rolnicy strajkowali, wyjechali ciągnikami, maszynami, wyrażając swój zdecydowany sprzeciw wobec ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw. W Sejmie prace nad tą ustawą trwały bardzo krótko. Nie wzięto pod uwagę wielu aspektów i skutków tej ustawy. Ubój rytualny jest zgodny z prawem w Unii Europejskiej. Wykonuje go bardzo wiele krajów Unii Europejskiej, m.in. Francja, Hiszpania, Irlandia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Węgry.

Senat zamówił ekspertyzy, czekamy na nie. Dzisiaj także odbyła się debata w Top Agrar Polska, gdzie biorący w niej udział byli zdecydowanie przeciwko tej ustawie. O sytuacji w rolnictwie mówią nie tylko banki, pytają o płynność finansową, zatory płatnicze. Sytuacja w rolnictwie jest ciężka. Wczoraj rozmawiałem na posiedzeniu komisji rolnictwa z jej przewodniczącym Robertem Telusem o pilnym zwołaniu komisji rolnictwa celem omówienia wszystkich aspektów tej ustawy. Potrzebna jest debata na temat tej ustawy. Nie chcą podpisywania ustawy w tym kształcie.

Dzisiaj na transparentach były hasła: Ekolodzy i posłowie, ile wam płaci Zachód za niszczenie polskiego rolnictwa? Te dramatyczne hasła i to motto niech przemówi do posłów i senatorów, zanim dojdzie do głosowania [[Dzwonek]] w Sejmie i w Senacie nad tą ustawą.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z tej mównicy już niejednokrotnie mówiliśmy na temat sytuacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Tam rozgrywa się ludzka tragedia. Pana ludzie przygotowali właśnie wniosek o to, aby sprzedać część tego zakładu, zakład w Świnoujściu, w którym pracuje ponad 130 osób, zakład, który kiedyś został połączony, składał się z oddziału w Świnoujściu i w Szczecinie.

Pracownikom stoczni remontowej w Świnoujściu proponuje się pracę w Szczecinie. Każdego dnia 2 godziny wcześniej musieliby wstawać do pracy i tyle samo wracać.

Apeluję do pana, by nie pozbywać się tego zakładu. Branża remontowa ma przyszłość w Polsce, a Świnoujście jest tym miejscem, gdzie można to robić i robi się od 50 lat. Dzisiaj ktoś, kogo pan wyznaczył na miejsce prezesa, chce zlikwidować ten zakład. Jemu nie zależy na tym, żeby utrzymać remonty statków w Świnoujściu, tam jest tylko i wyłącznie kwestia finansów i budowy kolejnej megalomanii, wielkiego doku dla stoczni remontowej w Szczecinie za podobno 150 albo 300 mln zł. Tylko kto da im na to kredyt, jeżeli dzisiaj stocznia remontowa Gryfia jest zadłużona? Apeluję, panie premierze, do pana, żeby nie niszczyć oddziału w Świnoujściu. Tam oni mają swój portfel zamówień, mają swoich kontrahentów, z którymi współpracują od wielu, wielu lat. A dzisiaj chce się ich pozbawić miejsc pracy. Dlatego też my jako posłowie zachodniopomorscy będziemy starali się bardzo mocno apelować, bo wiem, że w tym tygodniu ma zostać podjęta decyzja właśnie o tym, żeby sprzedać ten oddział w Świnoujściu i żeby zamknąć całkowicie remonty statków w Świnoujściu. Panie premierze, apeluję, opamiętajcie się, bo powrotu już nie będzie. Dziękuję bardzo. Nie ma pana posła. Pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W tym roku obchodziliśmy 100-lecie Bitwy Warszawskiej.

To przez Lorda Edgara D’Abernona, ambasadora brytyjskiego w przedwojennej Polsce. W tamtym okresie Polacy uratowali Europę przed falą komunizmu. Plany Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina obejmowały zdobycie Lwowa, następnie Czech, Węgier, Rumunii, Austrii i Włoch. Bitwa Warszawska składała się z trzech faz: walk obronnych na przedpolach Radzymina, bitwy obronnej i manewru zaczepnego 5. armii gen. Sikorskiego nad Wkrą oraz uderzenia grupy manewrowej znad Wieprza i pościgu.

Następnie okrążono i zniszczono sowiecką armię na froncie północnym, co zawdzięczamy szybkości polskiej piechoty i decyzyjności naczelnego wodza. Decyzja ta była spóźniona, ponieważ bolszewicy uciekli w popłochu, o czym poinformowali Józefa Piłsudskiego okoliczni mieszkańcy. Zmierzając do Mińska Mazowieckiego, Naczelny Wódz doszedł do wniosku, że większość Rosjan musi się cofnąć od Warszawy ku wschodowi. Należy zatem jak najszybciej zarządzić zupełną jednolitość działań wszystkich wojsk zebranych pod Warszawą, aby po rozbiciu jednej z sowieckich armii energicznym pościgiem i naciskiem zewsząd rozbić i porazić resztę sił nieprzyjacielskich. Piłsudski przekazał dowodzenie grupom uderzeniowym znad Wieprza gen. Edwardowi Rydzowi-Śmigłowi, sam zaś już w Warszawie wspólnie z gen. Tadeuszem Rozwadowskim, głównym architektem zwycięstwa nad bolszewikami, opracował rozkaz pościgu na liniach Międzyrzec, Białystok, Kałuszyn, Mazowieck, Warszawa, Łomża. Rozpoczęła się kontrofensywa Polaków na całej linii frontu. W wyniku bitwy warszawskiej 15 października zawarto w Rydze zawieszenie broni, a następnie traktat pokojowy. Tym samym aż do agresji na Polskę przez Związek Sowiecki - przypominam, że do dzisiaj obchodzimy tę rocznicę - ustalono polsko-rosyjskie stosunki, ukształtowano granicę wschodnią.

Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom! Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W Polsce od 2 lat wprowadzana jest reforma psychiatrii, która bazuje na opiece ambulatoryjnej zamiast na lecznictwie w zamkniętych szpitalach. Tego rodzaju rozwiązanie daje poczucie bezpieczeństwa i ciągłość leczenia dla pacjentów, a uzyskanie przez nich właściwego wsparcia dobranego do indywidualnych potrzeb powoduje, że osoby te łagodniej przechodzą kryzysy, nie są pozostawione same sobie i wyizolowane od społeczeństwa, a przede wszystkim wiedzą, gdzie szukać pomocy. Bardzo dobrym przykładem placówki funkcjonującej w ramach programu pilotażowego jest działające od 2 lat w moim regionie Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie, dzięki któremu diametralnie polepszyła się dostępność porad specjalistycznych z zakresu psychiatrii w powiecie cieszyńskim. Niestety rozpoczęty pilotaż został zahamowany w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem lockdownu, gdzie wiele organizacji musiało się przebranżowić, by móc nadal funkcjonować. Przykład z Cieszyna pokazuje, że oferowana pomoc leczenia środowiskowego pozwala dotrzeć do osób, które nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej, a wcześniej jedyną formą leczenia była hospitalizacja. Fakt, iż do specjalisty można dostać się bezpłatnie, bez długiego oczekiwania na termin wizyty stanowi niezwykle ważny argument podnoszący sens istnienia takich placówek. Obecnie proces reformowania opieki psychiatrycznej znajduje się w kluczowym dla powodzenia momencie i wymaga pilnych decyzji, jeśli chodzi o kontynuację, szczególnie teraz, kiedy podczas pandemii znacznie powiększyła się liczba osób szukających pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej. Jako kraj nie możemy sobie pozwolić na finansowanie psychiatrii na poziomie przedostatniego miejsca w Unii Europejskiej. Dlatego bardzo ważna jest kontynuacja rozpoczętej reformy i stworzenie systemu opieki, który byłby przyjazny i ludzki oraz to, żeby takie placówki jak ta w Cieszynie mogły nadal skutecznie wspierać chorych w potrzebie. Dziękuję. I bardzo proszę, pan poseł Piotr Adamowicz, Koalicja Obywatelska. Jeżeli pani pozwoli, podziękuję też obecnym pracownikom Sejmu, bo pora lekko późnawa. Otóż Wysoka Izba przyjmuje niemal na każdym posiedzeniu uchwały, które mają upamiętnić, uczcić, przypomnieć pewne ważne postaci lub też pewne ważne wydarzenia w historii naszego kraju. W przeddzień 40. rocznicy polskiego Sierpnia przewodniczący Borys Budka złożył do marszałek Witek projekt uchwały dotyczący właśnie 40. rocznicy polskiego Sierpnia. Niestety, ale tenże projekt został skierowany do tzw. międzyklubowych konsultacji.

Dlatego chciałem przeczytać kilka fragmentów z tejże uchwały - bezspornych: 14 sierpnia 1980 r. wybuchł strajk w ówczesnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Bezpośrednią przyczyną strajku było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz.

Sejm RP dziękuje i wyraża uznanie ludziom Sierpnia za ich działanie na rzecz wolności, a także wszystkim ludziom dobrej woli z całego świata, którzy wspierali ruch solidarnościowy. Jako autor tego projektu przyznam, że bardzo ubolewam, że polski Sejm nie był w stanie przyjąć stosownej uchwały, podkreślam - bardzo neutralnej. Można się z nią zapoznać na stronie internetowej Sejmu. Niestety powiem to, ale chcę przypomnieć koleżankom i kolegom posłom, że dzięki ludziom Sierpnia, dzięki polskiemu Sierpniowi mogą dziś w wolnej, niepodległej Polsce zasiadać w tym miejscu. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam panią poseł Monikę Falej, Lewica. Wysoka Izbo! Oznacza to, że liczba wszystkich przypadków zakażeń w województwie od początku pandemii wynosi 2144. Łączna liczba przypadków śmierci w województwie warmińsko-mazurskim spowodowanej zakażeniem COVID-19 od początku pandemii wynosi 26. W tym samym czasie elblążanki i elblążanie toczą walkę o oddział ginekologiczno-położniczy w szpitalu miejskim w Elblągu.

Szpitale szukają wolontariuszy do obsługi pacjentów, ponieważ zostały wycofane wojska terytorialne.

Pragnę wyrazić zaniepokojenie - i niezrozumienie - utrzymywaniem wydatków na obronność na takim poziomie. W budżecie zapisano 15 mld na wydatki zbrojeniowe. Czy z koronawirusem i zapaścią gospodarczą będziemy walczyć armatami, kupując wojskowy sprzęt za granicą? Czy to naprawdę jest konieczne, szczególnie w czasie, gdy szukamy oszczędności wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, gdy brakuje środków na zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania służby zdrowia? Niepokoi tak wysoki poziom, szczególnie że jest to jeden z najwyższych poziomów w NATO i przekracza o 0,2% wymagany poziom, wymóg, którego i tak wiele państw członkowskich nie spełnia. Apeluję zatem, aby te środki zostały przekazane na walkę z obecnym wrogiem, którym jest pandemia, w tym na służbę zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim. Dziękuję bardzo. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.